Wznawiam posiedzenie. Na sekretarzy dzisiejszych obrad powołuję posłów Agatę Borowiec, Monikę Wielichowską, Jarosława Szlachetkę i Arkadiusza Marchewkę. W pierwszej części obrad sekretarzami będą posłowie Monika Wielichowska i Arkadiusz Marchewka. Protokół i listę mówców prowadzić będą posłowie Monika Wielichowska i Jarosław Szlachetka. Proszę panią poseł o odczytanie komunikatów.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 Nadzwyczajnej do spraw deregulacji - godz. 15.30. Dzisiaj odbędą się także posiedzenia następujących zespołów parlamentarnych: - Parlamentarnego Zespołu ds. wyjaśnienia nieprawidłowości w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej - godz. 10, - Parlamentarnego Zespołu ds. Dziedzictwa Świętego Jana Pawła II - godz. 11, Parlamentarnego Zespołu ds. Organizacji Ochrony Zdrowia - godz. 15, - Parlamentarnego Zespołu ds. Reformy Kodeksu Pracy - godz. 15.30, - Parlamentarnego Zespołu ds. rozwiązywania problemów mieszkańców „Polski powiatowo-gminnej” - godz. 16, - Parlamentarnego Zespołu Szachowego - godz. 20. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pani poseł. Właściwe komisje przedłożyły sprawozdania o rządowych projektach ustaw: - o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, - o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Sprawozdania to odpowiednio druki nr 2713 i 2714. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, marszałek Sejmu podjął decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkty obejmujące rozpatrzenie tych sprawozdań.

Jeżeli nie będę słyszała sprzeciwu, uznam, że Sejm propozycje przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 27. porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Przypominam, że postawienie pytania nie może trwać dłużej niż 2 minuty, zaś udzielenie odpowiedzi nie może trwać dłużej niż 6 minut. Prawo do postawienia pytania dodatkowego przysługuje wyłącznie posłowi zadającemu pytanie. Dodatkowe pytanie nie może trwać dłużej niż 1 minutę, a uzupełniająca odpowiedź nie może trwać dłużej niż 3 minuty.

Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Polska w chwili obecnej jest liderem w branży informatycznej w naszej części Europy. Nasi informatycy, testerzy oprogramowania, architekci systemów IT, menedżerowie cyberbezpieczeństwa stanowią o sile rozwoju naszego sektora i całej branży IT. Jednak wraz z rozwojem branży należałoby podjąć działania, które skutecznie zachęciłyby do zatrzymania obecnych specjalistów w naszym kraju. Przedsiębiorstwa, firmy informatyczne postulują o zmniejszenie podatków nakładanych na informatyków. Nie jest tajemnicą, że naszych specjalistów chętnie przyciągnęłyby do siebie inne kraje. Skutecznym rozwiązaniem mogłyby okazać się obniżenie stawki podatku dochodowego oraz uznanie tworzenia programów komputerowych za działalność badawczo-rozwojową. W związku z powyższym pragnę zapytać: Czy czynione są starania, aby móc skutecznie zachęcić specjalistów z branży informatycznej do dalszego rozwijania swoich przedsiębiorstw? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Na pytanie odpowiada podsekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii pan Marcin Ociepa. Bardzo proszę. Szanowna Pani Marszałek! Panie i Panowie Posłowie! Panie Pośle!

Dzisiaj, kiedy stoimy u progu czwartej rewolucji przemysłowej w gospodarce, opartej na wiedzy i danych, w której kluczową rolę ma odgrywać robotyzacja, rozwój sztucznej inteligencji, magazynowanie energii, rozumiemy, że wszystkie te aspekty diametralnie zmienią obraz gospodarczy świata, w tym także Polski. Jeśli chodzi o kwestie podatkowe, to odpowiedź jest w gestii ministra finansów.

Chcę powiedzieć, że dzisiaj widzimy, że na ten moment Polska jest absolutnym liderem, jeśli chodzi o branżę FinTech i wszystko, co się z tym wiąże. Według rankingów Global Financial Centres Index, które badają konkurencyjność głównych centrów finansowych, zajmujemy na świecie 45. miejsce, w Europie - 12. Jesteśmy wiodącym centrum finansowym w Europie Środkowo-Wschodniej. Z kolei z raportu Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Finansowego wynika, że Polska jest jednym z 14 państw najbardziej wspierających branżę FinTech.

Sama ustawa o innowacyjności wprowadziła do porządku prawnego usprawnienia polegające na zniesieniu opodatkowania podatkiem dochodowym aportu własności intelektualnej i przemysłowej, wprowadziła ulgi podatkowe na badania i rozwój, sukcesywnie rozszerzając listę kosztów kwalifikowanych, wydłużyła z 3 do 6 lat okres, w jakim przedsiębiorca może odliczyć koszty poniesione na działalność badawczo-rozwojową, oraz wprowadziła możliwość zwrotu gotówkowego dla nowo powstających przedsiębiorstw prowadzących działalność badawczo-rozwojową.

Jesteśmy gotowi i otwarci na dialog z branżą po to, by tworzyć jak najlepsze warunki.

Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pana posła o pytanie dodatkowe. Panie Ministrze! Kobiety stanowią połowę populacji świata, tymczasem kobiety w dalszym ciągu w wielu przypadkach są wręcz zniechęcane do rozwoju kariery czy też aspirowania do zawodów stereotypowo postrzeganych jako typowo męskie. W Stanach Zjednoczonych wdraża się już nowe sposoby edukacji i zachęcania kobiet do zainteresowania się nowymi technologiami już od wczesnego wieku nastoletniego.

Szanowny Panie Pośle! Jesteśmy resortem, w którym szefową jest kobieta, która absolutnie wyznacza trendy, jeśli chodzi o działalność innowacyjną. To my staramy się ją gonić w tym profesjonalizmie i zapale z tym związanym. Oczywiście to jest aspekt, powiedziałbym, kulturowy.

Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Przechodzimy do następnego pytania. Pytanie dotyczy działań rządu na rzecz zwiększenia sprawności systemu ratowniczo-gaśniczego oraz wspierania jednostek ochotniczych straży pożarnych. Proszę bardzo pana posła Dariusza Starzyckiego o zadanie pytania. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Występujące liczne zagrożenia o różnorodnym charakterze, takie jak pożary, wypadki komunikacyjne, działania sił przyrody, skażenia środowiska, powodują, że państwo i społeczeństwo potrzebują sprawnych służb ratowniczo-gaśniczych, które będą w stanie szybko i skutecznie reagować na zaistniałe zdarzenia. W Polsce zadania te wykonują Państwowa Straż Pożarna i jednostki ochotniczych straży pożarnych, z których część włączona jest do systemu ratowniczo-gaśniczego, a część pozostaje poza systemem. W związku z powyższym proszę pana ministra o przedstawienie informacji na temat działań Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i rządu w zakresie wspierania tych służb, jeśli chodzi o wyposażenie w niezbędny sprzęt i poprawę stanu niezbędnej do tej działalności infrastruktury. W jaki sposób pod względem finansowym minister spraw wewnętrznych i administracji zadbał o sprawność krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz o ochotnicze straże pożarne? Czy i ewentualnie jakie działania prawne lub organizacyjne zostały podjęte w celu udoskonalenia systemu? Jaka jest wielkość środków budżetowych kierowanych zwłaszcza do jednostek ochotniczych straży pożarnych w poszczególnych latach? Szanowny Panie Ministrze! Jak pan minister ocenia współpracę z samorządami lokalnymi? Chciałbym też zapytać o fundusz ochrony środowiska, Lasy Państwowe.

Bardzo proszę sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji pana ministra Jarosława Zielińskiego o odpowiedź na pytania. Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Straż pożarna jest najbardziej wielofunkcyjną ze wszystkich służb. Wiemy, jakie spełnia dzisiaj zadania.

Nie chcę ich definiować, bo zabrakłoby czasu, a państwo wiecie, czym zajmuje się straż pożarna, jak jest wielozadaniowa, wielofunkcyjna. Powiem może tylko, bo to działa na wyobraźnię, że właściwie nie ma minuty, żeby w jakimś miejscu w Polsce strażacy nie wyjeżdżali do akcji, żeby nie podejmowali interwencji. W 2017 r. wyjeżdżali ponad 520 tys. razy.

Ze względu na rolę systemu ratowniczo-gaśniczego, ze względu na rolę w ochronie przeciwpożarowej jednostek straży pożarnej, ze względu na ich rolę w systemie bezpieczeństwa państwa i obywateli rząd Prawa i Sprawiedliwości wspiera na różne możliwe sposoby jednostki państwowej i ochotniczej straży pożarnej oraz system ratowniczo-gaśniczy. Może warto powiedzieć, że do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego należy 501 jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej, 4404 jednostki OSP włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, 5 zakładowych straży pożarnych, 5 jednostek wojskowej ochrony przeciwpożarowej i 1 lotniskowa straż pożarna. Razem to jest 4916 jednostek. One są wspierane przez ponad 12 tys. jednostek OSP nienależących do tego systemu, bo jednostek ochotniczych straży pożarnych razem jest 16 217. To jest potężny obszar, bardzo liczne jednostki rozlokowane na terenie całej Polski.

Zwiększamy coroczne nakłady budżetowe na jednostki ochotniczej straży pożarnej.

W roku 2018 dotacje budżetowe dla jednostek OSP z krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i spoza tego systemu wynoszą razem 137 585 tys. zł. W tym miejscu chcę podziękować tym posłom, posłom Prawa i Sprawiedliwości, którzy w ramach poprawek do budżetu państwa na rok 2018 zaproponowali konkretne kwoty skierowane do jednostek OSP, a w niektórych przypadkach także do Państwowej Straży Pożarnej. Jest to istotne wzmocnienie finansowania tego systemu. Szanowni Państwo! Ponadto integrujemy wysiłki - jest to odpowiedź na jedno z pytań, które padły - podejmujemy wspólne działania z różnymi podmiotami, aby zakupić jak najwięcej sprzętu, zwłaszcza samochodów ratowniczo-gaśniczych, a także innego rodzaju sprzętu potrzebnego systemowi ratowniczo-gaśniczemu. I tak na 2018 r., a więc rok bieżący, zaplanowaliśmy w ramach integracji wysiłków i tworzenia takiego montażu finansowego różnych podmiotów zakup co najmniej 382 samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP w całym kraju.

Na to składają się środki zarówno Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, jak i - trzeba podkreślić to, że w większej kwocie niż środki budżetowe - jednostek samorządu terytorialnego, narodowego funduszu ochrony środowiska i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, Lasów Państwowych, a czasem także innych podmiotów, również środki pochodzące z odpisu od firm ubezpieczeniowych. Pamiętacie państwo zmianę, jaka dokonana została przez Wysoki Sejm w tym zakresie, żeby ujednolicić system finansowania systemu ratowniczo-gaśniczego [[Dzwonek]] jednostek ochotniczych straży pożarnych.

Bardzo proszę pana posła Jerzego Paula o zadanie pytania dodatkowego. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Panie Generale! Mam pytanie częściowo związane ogólnie ze strażą pożarną: Czy Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej wspiera finansowo i organizacyjnie obozy szkoleniowo-wypoczynkowe dla członków młodzieżowych drużyn pożarniczych? Jakie są środki finansowe przekazywane na te obozy? Jakim cieszą się powodzeniem wśród młodzieży? Dziękuję. I jeszcze raz proszę pana ministra Jarosława Zielińskiego o udzielenie odpowiedzi na pytanie. Nie zdążyłem odpowiedzieć oczywiście z braku czasu na wszystkie pytania, a też chciałem od siebie dodać parę ważnych informacji odnośnie do tego, co zostało podniesione w pierwszej turze pytań. Natomiast tutaj wspomnę tylko o bardzo istotnym wsparciu finansowym, jakiego udzielił minister sprawiedliwości prokurator generalny z tzw. Funduszu Sprawiedliwości jednostkom OSP. Te środki są przekazywane sukcesywnie w poszczególnych województwach. Ten proces jest już bardzo zaawansowany. Dziękując panu ministrowi Ziobrze za takie przeznaczenie tych środków, chcę jednocześnie podziękować pani minister Teresie Czerwińskiej za zgodę na wydatkowanie tych środków na ten cel. Oczywiście wspieramy młodzieżowe obozy pożarnicze środkami finansowymi. W 2017 r. w tych obozach wzięło udział 3300 młodych ludzi, a dofinansowanie wynosiło 2 mln zł.

W latach 2017 i 2018 obozy organizuje Państwowa Straż Pożarna z działaczami, członkami ochotniczych straży pożarnych w terenie, zwłaszcza w powiatach. Chcę wszystkim, którzy w to się angażują, bardzo podziękować, bo to jest bardzo ważny element wychowania ku aktywności, która będzie służyła bezpieczeństwu wszystkich obywateli. Było pytanie - korzystam jeszcze z tego, że mam czas - o współpracę z samorządami i innymi podmiotami. Ta współpraca jest dobra, a nawet, mogę powiedzieć, wyśmienita, dlatego że wszyscy doskonale rozumieją potrzeby jednostek straży pożarnej. Wspieramy je w ramach współdziałania, każdy podmiot, takimi środkami, jakie są dostępne. A dzięki scentralizowaniu decyzji - to jest możliwe pierwszy raz w tym roku - możemy kupić więcej samochodów ratowniczo-gaśniczych, bo uzupełniamy sobie wzajemnie te wkłady. Na koniec dodam jeszcze, przypomnę w zasadzie, jako że państwo to wiecie, bo to przecież była informacja publicznie często przywoływana, że od 2016 r. wprowadziliśmy nowy system udzielania dotacji dla jednostek OSP.

I bardzo proszę, następne pytanie zadają posłowie Sławomir Nitras i Paweł Olszewski, Platforma Obywatelska, w sprawie renegocjacji kontraktów i umów z wykonawcami państwowych inwestycji.

Dziękuję, pani marszałek, i dzień dobry przy okazji. Szanowni Państwo! Sprawa jest niezmiernie poważna. Wtedy po raz pierwszy doszło do takiej sytuacji i brak nam było wówczas pewnego doświadczenia, co z tym robić, dzisiaj mamy zagrożenie podobne, ale mamy już doświadczenie, mamy oprzyrządowanie, mamy zmienione ustawy, wiemy, że jest możliwość renegocjowania kontraktów podpisanych z wykonawcami inwestycji. Przypomnę - ustawa, którą znowelizowaliśmy w roku 2014, pozwala na to w przypadku gwałtownego wzrostu cen, kosztów pracy, kosztów materiałów, zmiany VAT, zmiany podatkowej. Odwrócony VAT to jest to, co najbardziej dotyczy podwykonawców, co zagraża podwykonawcom. Szanowni państwo, dzisiaj - to zjawisko na masową skalę - albo stoją na granicy bankructwa, albo zastanawiają się nad zejściem z realizowanych inwestycji firmy, które podpisywały umowy w roku 2015 i w roku 2016. Mamy do czynienia z sytuacją taką, że wycofują się one z kontraktów czy z negocjacji, wycofują swoje oferty. Ostatnia historia, droga S3, odcinek Kamienna Góra - Lubawka - dziewięć firm wycofało swoje oferty, mając świadomość, że nie jest w stanie ich zrealizować. To jest problem. Pytania: Czy rząd dostrzega ten problem? Czy rząd prowadzi rozmowy z tymi firmami? Czy rząd jest skłonny do negocjacji czy do renegocjacji tych kontraktów, mając świadomość upływającego czasu? To nie jest problem nowy, my ten problem obserwujemy co najmniej od miesięcy i jesteśmy ciekawi efektów działań rządu i planów działań rządów.

Dziękuję, panie pośle. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! My rozpoczęliśmy już w 2016 r. współpracę z wykonawcami przy wszystkich państwowych kontraktach dotyczących tak dróg, jak i kolei. W tej chwili kontynuujemy to w ramach tzw. Rady Ekspertów. Rada ekspertów jest taką platformą współpracy i wymiany poglądów, która ma za zadanie wypracowanie lepszych warunków w relacjach pomiędzy inwestorem a wykonawcą.

Wykonawcy właśnie na forum rady ekspertów podnoszą kwestię znaczącego wzrostu cen, który powoduje, że zawarte z inwestorami, z inwestorem państwowym, jeszcze nieukończone kontrakty przestały być dla nich opłacalne, i może się przyczynić do upadłości wykonawcy. Część zrealizowanych obecnie umów o realizację przewiduje górny pułap waloryzacji na poziomie najwyżej 1% przy zastosowaniu wskaźników opracowanych przez GUS: wskaźnika cen obiektów drogowych oraz wskaźnika cen obiektów mostowych. To nie satysfakcjonuje wykonawców. Wykonawcy chcieliby negocjować z inwestorem waloryzację swojego wynagrodzenia, aby pokryć straty wynikające z ponadprzeciętnych w ich ocenie wzrostów kosztów kluczowych materiałów. Jednak dochodzenie waloryzacji na drodze sądowej uznają za czasochłonne, kosztowne i nierozwiązujące problemu, jakim jest brak środków na bieżące działanie i dokończenie zadań w terminie. Czasem w dyskursie publicznym pojawia się temat różnych kosztów dotyczących ewentualnych roszczeń z tego tytułu, natomiast one są bardzo różne i niepoparte danymi. Chcemy rozmawiać o konkretach, a nie spekulować. Zebranie takich danych wymagałoby od wykonawców zweryfikowania danych dotyczących realizacji poszczególnych umów, konkretnych powodów, przyczyn i wpływu na czas i koszt. W ocenie Ministerstwa Infrastruktury zastosowanie mechanizmów wcześniejszych, niż wynikałoby to z warunków kontraktowych, i większych, bo uwzględniających waloryzację wypłat na rzecz wykonawców, powinno być poprzedzone analizą dotyczącą tego, czy jest to dopuszczalne na gruncie obowiązujących przepisów i jakie to będzie miało konsekwencje prawne i finansowe dla obu stron. W związku z powyższym resort doszedł do wniosku, że trzeba rozważyć następujące sprawy: Czy zmiany wysokości wypłat dla wykonawców nie będą powodowały korekt finansowych w zakresie dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej? Czy możliwa jest zmiana wysokości zobowiązań Skarbu Państwa w zawartych już kontraktach ponad planowane dotychczas wydatki? Czy wypłaty stanowiłyby niedozwoloną pomoc publiczną? To jest bardzo istotne. Czy zwiększenie wynagrodzenia z tytułu waloryzacji od strony już zawartego kontraktu nie stanowi naruszenia Prawa zamówień publicznych? Resort zwrócił się do Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Ministerstwa Finansów, Urzędu Zamówień Publicznych i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z prośbą o opinię co do możliwości zastosowania tego typu rozwiązania, które pozwoliłoby na wypracowanie stanowiska strony rządowej i mogłoby wspomóc strony umów w osiągnięciu porozumienia w tej trudnej sytuacji. Te prace cały czas trwają, ostateczne rekomendacje jeszcze nie zostały przedstawione. Jednocześnie na forum rady ekspertów podniesiona została kwestia tego, że wzrost cen w sektorze budowlanym nie znajduje odzwierciedlenia w danych opracowywanych przez GUS, do którego kompetencji należy szczegółowa analiza cen w oparciu o otrzymywane od jednostek sprawozdawczych dane. W związku z powyższym na spotkanie rady ekspertów zostali zaproszeni przedstawiciele GUS, aby możliwe było zbadanie przyczyny różnic między wskaźnikami opracowanymi przez GUS a faktycznymi cenami na rynku. Przedstawiciele GUS wyjaśnili zasady metodologii stosowanej przez tę instytucję. Okazało się, że firmy będące jednostkami sprawozdawczymi informują GUS o cenach robót budowlanych i obiektów na podstawie już zawartych kontraktów, a nie faktycznych kosztów. W praktyce oznacza to, że wzrost cen. pojawia się w statystykach GUS z opóźnieniem. Przedstawiciele GUS zadeklarowali chęć współpracy i otwartość na ewentualne zmiany w przyjętej dotychczas procedurze. W konsekwencji GUS podjął działania we współpracy z przedstawicielami branży drogowej mające na celu zmianę metodologii, tak aby wskaźniki odzwierciedlały rzeczywiste ceny towarów i usług. W ramach tych działań GUS przeprowadził konsultacje z wybranymi wykonawcami, firmami będącymi jednostkami sprawozdawczymi w celu wypracowania nowej, zmodernizowanej wersji tzw. formularza C4, który panowie posłowie na pewno znacie. Obecnie GUS prowadzi badania we współpracy z wykonawcami, a jeśli wyniki tych badań będą pomyślne, to wskaźnik GUS, na który powołują się w kontraktach inwestorzy państwowi, będzie w lepszy niż dotychczas sposób odzwierciedlać tendencje na rynku. Innym zagadnieniem jest wzrost wynagrodzenia dla pracowników budowlanych. Coraz mocniej jest odczuwalny niedobór pracowników. W Ministerstwie Infrastruktury były prowadzone analizy możliwości ułatwienia zatrudniania w branży budowlanej np. pracowników z wybranych krajów Europy Wschodniej czy Azji. W te potrzeby wpisują się działania Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ułatwiające zatrudnianie cudzoziemców, w tym z branży budowlanej. Według mojej wiedzy rozporządzenie jest przygotowywane przez ministra pracy. Podsumowując: Ministerstwo Infrastruktury jest otwarte na rozmowy z wykonawcami. Nie uchylamy się od rozmów, w tym tych dotyczących waloryzacji cen. Widzimy problemy na rynku, w tym wzrosty cen niektórych materiałów. Nie będziemy natomiast ulegać panice, [[Dzwonek]] jaką próbuje się wywołać. Rozmawiamy i nadal będziemy rozmawiać merytorycznie o poszczególnych, istotnie trapiących wykonawców problemach. Bardzo proszę pana posła Pawła Olszewskiego, Platforma Obywatelska, o zadanie drugiego pytania. Pani Marszałek! Ja pana uwielbiam. 5 minut odpowiadać na pytanie i na nie nie odpowiedzieć, to jest naprawdę wielka rzecz. Z całym szacunkiem dla tego, co pan powiedział. Mówi pan, że od 2016 r. rozmawiacie z wykonawcami. Jest 2018 r., żadnych rozwiązań i pomysłów na rozwiązanie tego problemu nie macie. Rezultat będzie taki, że państwo - jesteście tak niedecyzyjni, tak boicie się podejmować jakiekolwiek decyzje, dostrzegając problem, o czym pan powiedział - doprowadzicie do sytuacji, w której polscy wykonawcy, m.in. polscy wykonawcy, i podwykonawcy, którzy schodzą już z budów - bardzo bliska jest mi droga ekspresowa S5, podwykonawcy schodzą z budów - nie wykonają założeń „Programu budowy dróg krajowych”, który ja przygotowywałem w resorcie i który rząd przyjął 8 września 2015 r. Co gorsza, stracimy pieniądze z Unii Europejskiej. Państwo jako resort infrastruktury doprowadzacie do katastrofy, [[Dzwonek]] za którą zapłacą wszyscy obywatele. Będziemy mieli rozkopaną Polskę z upadłymi polskimi firmami.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Ja z wielkim szacunkiem wysłuchałem pańskiej opinii, ale nie usłyszałem pytania. i te decyzje są w tej chwili wypracowywane. Dziękuję bardzo. Dziękuję panom posłom. Przechodzimy do następnego pytania. Pytanie zadają posłowie Jarosław Sachajko i Norbert Kaczmarczyk, klub Kukiz’15, w sprawie aktualnego stanu rozprzestrzeniania się choroby ASF u dzików oraz w stadach świń hodowlanych, z uwzględnieniem podjętych działań dotyczących zwalczania choroby z urzędu i rozwiązań pomocowych dla poszkodowanych rolników, a także w sprawie przedstawienia wariantów zwalczania choroby w razie rozprzestrzeniania się jej na terenie zachodniej Polski - pytanie do ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Bardzo proszę, pierwsze pytanie - pan poseł Jarosław Sachajko. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Sprawa jest wyjątkowo ważna - wyjątkowo ważna dla polskich rolników, ale i dla wszystkich obywateli. Polscy rolnicy są bardzo dobrzy w produkcji trzody chlewnej, jest zapotrzebowanie na taką produkcję. W ubiegłym roku delikatnie zwiększyła się produkcja trzody chlewnej w Polsce, ponieważ rolnicy wiedzą, jak to robić - wiedzą, jak to robić tak, żeby to w jakiś sposób im się opłacało. Niestety rozprzestrzeniająca się choroba ASF niszczy kolejne gospodarstwa rodzinne, niszczy tę wiedzę, którą mieliśmy, niszczy polskie wsie. Zadałem tutaj przedstawione przez panią marszałek bardzo precyzyjne pytanie i prosiłbym o równie precyzyjną odpowiedź. Choroba ASF jest zwalczana z urzędu i jakie działania są podjęte, aby w końcu skończyć w Polsce z tą chorobą? Panie ministrze, trzeci rok jest przespany, trzecia zima jest przespana. Nie zdołaliśmy jako państwo polskie. Ja również czuję się za to odpowiedzialny, ponieważ może za mało krzyczałem, za mało naciskałem na to, aby doprowadzić do depopulacji dzików w środowisku. Jeżeli okazujemy słabość przy zwalczaniu, wydaje się, bardzo prostej choroby. Oczywiście, możemy mówić, i ja na pewno to za chwilę usłyszę, jak to inni sobie z nią nie poradzili. Uczymy się, powinniśmy się uczyć na błędach innych, dlatego nie powtarzajmy tego, tylko chodzi o to, co zrobimy i jakie są warianty walki, jeżeli za chwileczkę ta choroba pojawi się w Polsce zachodniej, gdzie mamy największe stada. To będą miliardowe straty. Co w tej chwili zrobimy, [[Dzwonek]] aby wyhamować rozprzestrzenianie się tej choroby? Bardzo proszę sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pana ministra Jacka Boguckiego. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie pośle, dziękuję za to pytanie. Problem afrykańskiego pomoru świń jest najpoważniejszym problemem gospodarczym w rolnictwie, obok suszy, innych zjawisk atmosferycznych, które zdarzały się i zdarzają. Ale to jest też, podobnie jak w przypadku suszy, niezależna od człowieka, niezależna od ludzi choroba, wirus, który na szczęście nie szkodzi ludziom, nie przenosi się na ludzi. Draństwem jest to, co robią media ostatnio, pisząc o produktach z terenów ASF. To jest draństwo, to jest w ogóle sabotaż wobec polskiej gospodarki, ponieważ tylko zdrowe zwierzęta trafiają do przerobu, niezależnie od tego, z którego miejsca Polski, wszystkie chore są utylizowane. I o tym trzeba mówić, i o tym trzeba mówić głośno.

Panie ministrze, bardzo proszę ważyć słowa.

Nie wolno choroby. nawet jeśli ta choroba dotyczy zwierząt. i nie dotyczy ludzi. Nie wolno choroby wykorzystywać przeciwko polskiej gospodarce i polskiemu rolnictwu. Szanowni państwo. Walki z tą chorobą, ja to kiedyś powiedziałem, uczymy się ciągle - uczymy się ciągle, bo nie było na świecie przypadku, kiedy choroba wystąpiła jednocześnie u świń, w hodowli, i w środowisku, czyli u dzików. Nie było też przypadku, nie ma kraju na świecie, który ma zmilitaryzowane łowiectwo. Gdybyśmy mieli łowiectwo zmilitaryzowane, w mundurach, wysłalibyśmy tę służbę, żeby wystrzelała wszystkie dziki. Łowiectwo w Polsce jest ochotnicze, jest dobrowolnym zrzeszeniem ludzi. Łowiectwo jest poubeckie, no bo przecież ubowcy byli myśliwymi za komuny, bo normalny człowiek nie dostał pozwolenia na broń.

Po wojnie z myślistwa zrobiono elitarny sport dla ubowców, no bo przecież trzeba było być albo w ORMO, albo w PZPR, albo w PSL-u, albo w jakiejś innej partii, żeby dostać pozwolenie na broń. Przecież ktoś, kto był w opozycji - mój ojciec był żołnierzem Narodowych Sił Zbrojnych, ludzie - jak mój ojciec nie dostał pozwolenia na broń. Nie dostałby, bo miał broń, ale w czasie wojny. Ja też nie jestem myśliwym, bo za komuny nie dostałbym pozwolenia na broń. Z tą chorobą będziemy walczyć, panie pośle, długo i musimy sobie z tego zdawać sprawę. Oczywiście najważniejsze jest ograniczenie populacji dzików.

To jest pierwszy problem, który musimy rozwiązać. I to trwa, jest on rozwiązywany przez ministra Kowalczyka i będzie rozwiązany. A naszym zadaniem jako resortu rolnictwa jest, z jednej strony, wzmocnienie służb weterynaryjnych przede wszystkim, ale też służb granicznych, wszystkich służb odpowiedzialnych za zabezpieczenie gospodarstw i, z drugiej strony, rekompensowanie rolnikom wszelkich strat. Trzeba po prostu rolnikom zrekompensować straty. Mamy zbudowany system, który już działa.

Rolnik będzie miał prawo wystąpić do agencji o zwrot 75% kosztów bioasekuracji. Takiego działania nie było, do tej pory to było 50% i tylko na obszarach z ASF-em. Dzisiaj będzie to obowiązywać na terenie całego kraju, po uchwaleniu przez Radę Ministrów oczywiście.

To są koszty. I ci rolnicy będą mogli korzystać z rekompensaty przez 3 lata za zaprzestanie hodowli.

Przepraszam. Wysoka Izbo! Panie ministrze, jak najbardziej zgadzam się w tej części, w której pan mówił, że jest to obecnie najważniejszy problem polskiego rolnictwa. Nie zgodzę się z tym, że nie mamy na to wpływu, tak jak na suszę, gdzie mamy bardzo ograniczony wpływ, ale też mamy.

Ja składałem poprawkę do ustawy Prawo łowieckie, aby rolnicy mogli swobodnie dostawać się do kół łowieckich. A więc jeżeli legislacyjnie sami pozwalamy na to, to tak to działa.

I bardzo proszę pana ministra o udzielenie odpowiedzi. Wysoka Izbo! Panie pośle, pan źle zrozumiał moją wypowiedź. Jeśli chodzi. o depopulację dzików, to jest to podstawowe zadanie, które musi być realizowane i jest realizowane.

Oczywiście są tam szlachetni ludzie, wielu myśliwych to są szlachetni ludzie, ale ja mówię o całym systemie, który był stworzony za komuny. Nie brońcie tego. Jeśli bronicie draństwa, jeśli bronicie ubecji, to zastanówcie się. Jeśli chodzi o pomoc dla rolników, pani marszałek, panie pośle przewodniczący komisji rolnictwa, Wysoka Izbo, to mówiłem już o tych 136 zł. To nie załatwia problemu, bo wiem, ile to 130 razy 50, umiem liczyć, ale to jest tylko rekompensata za utracone dochody.

To jest jedno rozwiązanie. Drugie rozwiązanie.

A jeszcze w mniejszym procencie gospodarstw wystąpiła choroba. Tam gdzie są chore dziki, ja nie mówię o Polsce, jedno na 70 gospodarstw to jest to, które dotknęła ta najtragiczniejsza sytuacja związana z koniecznością wybicia świń. Jedno na 70, czyli 69 gospodarstw może nadal hodować i radzi sobie z bioasekuracją, nie wpuściło choroby do siebie. Podejrzewamy różne przyczyny przeniesienia. Nie wiemy do końca, jakie są drogi przenoszenia tego wirusa. Nie wiemy, czy nie ma celowego działania człowieka.

Nie bądźcie durniami. Panie pośle, panie ministrze, ja jednak muszę zwrócić uwagę na to, że swoim pierwszym wystąpieniem naruszył pan powagę Sejmu, i będę tę sprawę przedstawiała w Prezydium Sejmu. Przechodzimy do następnego pytania.

Wysoka Izbo! I Polacy, i Unia Europejska, nasi europejscy partnerzy niestety nie kupują kłamstw polityków PiS-u w sprawie wymiaru sprawiedliwości. Dlatego mam konkretne pytania. Jak ma się zamiar zachować obecny rząd w związku z rozpoczętą procedurą na podstawie art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej? Jak rząd PiS zamierza odpowiedzieć na list Komisji Europejskiej wzywający do usunięcia naruszeń w ustawie o Sądzie Najwyższym? Czy będą to te same zużyte już slogany niemające absolutnie nic wspólnego z prawdą, którymi starano się mydlić oczy naszym unijnym partnerom przez ostatnie miesiące? Czy politycy PiS zamierzają respektować ewentualny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydany w tej sprawie na niekorzyść polskiego państwa, tzn. jeśli Trybunał orzekłby w szczególności, że ustawa o Sądzie Najwyższym jest sprzeczna z traktatowymi kryteriami praworządności i niezależności sądownictwa? I ostatnie pytanie: Czy w razie wydania przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej np. nakazu wstrzymania wymiany sędziów w polskim Sądzie Najwyższym lub przywrócenia do pełnienia funkcji sędziowskich sędziów po 65. roku życia, którzy po 3 lipca 2018 r. mają przejść w stan spoczynku, rząd PiS ma zamiar zastosować się do takiego zabezpieczenia czy będzie je ignorował, tak jak to robił w przypadku Puszczy Białowieskiej i zakazu wycinki drzew do czasu wydania ostatecznego wyroku w sprawie, narażając w ten sposób Polaków na poniesienie olbrzymich kosztów? Przypomnę, 100 tys. euro kary za dzień. To, jak ważna jest sprawa łamania przez PiS standardów praworządności, było widać chociażby podczas wczorajszej debaty w Parlamencie Europejskim.

Dziękuję bardzo, pani poseł. Bardzo proszę sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych pana ministra Szymona Szynkowskiego vel Sęka o udzielenie odpowiedzi. Pani Marszałek! Szanowni Państwo Posłowie! Zanotowałem cztery.

Rzeczywiście chciałem stwierdzić, że w dniu 2 lipca Komisja Europejska wszczęła przedsądowe postępowanie, kierując do rządu wezwanie do usunięcia uchybienia. Przypomnę, że nie jest to, tak jak próbowali niektórzy twierdzić, pozwanie Polski przed Trybunał Sprawiedliwości czy też jakiś inny element tej procedury.

To pytanie muszę pozostawić w tej chwili jeszcze bez odpowiedzi, ponieważ do 2 sierpnia mamy czas na sformułowanie tej odpowiedzi, więc trudno mi, pani poseł, prognozować, co dokładnie będzie zawierała treść odpowiedzi rządu.

Kolejne dwa pytania są pytaniami, które zakładają w sobie pewne hipotezy. Pani poseł zakłada, że wyrok Trybunału Sprawiedliwości w ramach tej procedury zostanie wydany, co więcej, pani poseł stawia hipotezy, co ten wyrok będzie zawierał, i prosi o odpowiedź na pytania, co gdyby. Nie będziemy ustosunkowywać się do hipotez, ponieważ rolą rządu i Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które reprezentuję, jest odnoszenie się do faktów. a nie do prognoz czy też hipotez, które stawia pani poseł, bo to nie byłoby, jak sądzę, zasadne. Natomiast chcąc zadośćuczynić państwa pytaniom co do samej procedury, bo to być może państwa interesuje i rozjaśni też nieco sprawę. chciałbym powiedzieć, że postępowanie na podstawie art. 258 to jest jedno z toczących się ok. 750 postępowań prowadzonych na różnych etapach przez Komisję Europejską wobec różnych państw członkowskich. Przeciwko Polsce tego typu postępowań na bazie tego artykułu toczy się w tej chwili 34, ale przeciwko innym państwom, wskażę tu przykładowo, toczy się ich: przeciwko Niemcom - 49, a więc więcej, przeciwko Francji - 35, również więcej, przeciwko Hiszpanii - 58, przeciwko Grecji - 46, przeciwko Włochom - 52. Zwracam też uwagę - już starając się zadośćuczynić państwu i odpowiedzieć na pytanie o procedurę przed Trybunałem Sprawiedliwości, chociaż to jest pytanie hipotetyczne - że Polska wykonuje na bieżąco wszystkie wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i tylko raz w historii Komisja Europejska uruchomiła wobec Polski procedurę dotyczącą niewykonania wyroku. Sprawa ta dotyczyła niewłaściwego wdrożenia dyrektywy azotanowej - obecnie Komisja Europejska planuje zamknięcie tego postępowania. Inne państwa mają problem z wykonywaniem wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

W związku z tym widać dość jasno, jak Polska odnosi się do zaleceń Komisji Europejskiej czy to na pierwszym etapie kierowania, letter of formal notice - na tym etapie jesteśmy w przypadku sprawy, o którą państwo pytacie, czy to na etapie uzasadnionej opinii, czyli w drugim kroku, czy to w sytuacji, w której sprawa trafia przed Trybunał Sprawiedliwości. Polska respektuje wszystkie wyroki Trybunału Sprawiedliwości. Inne państwa niekiedy mają z tym problem. Mam nadzieję, że ta odpowiedź jest dla państwa satysfakcjonująca. Bardzo dziękuję.

Doskonale pan wie, że jeżeli nie usuniecie tych uchybień, to ta sprawa zostanie przed Trybunałem rozpatrzona. Pytanie jest więc proste: Czy odpowiadając na pismo Komisji Europejskiej, usuniecie uchybienia, które dotyczą ustawy o Sądzie Najwyższym? Dziękuję bardzo, panie pośle.

Szanowni Państwo Posłowie! Z ubolewaniem stwierdzam, że być może niewystarczającą uwagę poświęcacie państwo moim odpowiedziom na państwa pytania, ponieważ jasno powiedziałem, że letter of formal notice, czyli wezwanie do usunięcia uchybienia, jest etapem przedsądowym, a więc, panie pośle, nie jest elementem postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, tylko jest etapem przedsądowym. W związku z tym prosiłbym, żeby bardzo precyzyjnie tutaj do tej kwestii się odnosić.

One dotyczą bardzo różnych kwestii, wszystkie. na bazie procedury art. 258. Dotyczą również kwestii oceniających pewne elementy funkcjonowania sądów w różnych krajach, więc jeżeli państwo jesteście tym zainteresowani, to oczywiście bardzo chętnie wszystkie wskażemy, tylko prosimy o to, żebyśmy mieli wówczas trochę czasu. Dobrze, oczywiście jest to możliwe, tylko będzie potrzeba tutaj sporo czasu. Oczywiście zestawienie toczących się 750 postępowań. czego one mogą dotyczyć, dla państwa przygotujemy. Liczymy na państwa rzetelną analizę każdego z tych postępowań i wyciągnięcie odpowiednich wniosków. Dziękuję bardzo, panie ministrze.

Jest to pytanie w sprawie inicjatywy Komisji Europejskiej dotyczącej stanu realizacji programu wsparcia w procesie transformacji regionów górniczych i wysokoemisyjnych (Platforma Wsparcia Regionów Górniczych - do ministra energii. Bardzo proszę, pytanie zadaje pan poseł Grzegorz Matusiak. Dziękuję bardzo. Panie Ministrze! Wysoka Izbo!

Przygotowałem pytania dotyczące tego zagadnienia. Ostatnie posiedzenie grup roboczych w ramach inicjatywy Platformy Wsparcia Regionów Górniczych Komisji Europejskiej odbyło się w lutym 2018 r.

Drugie pytanie. Czy dialog pomiędzy Polską a Komisją Europejską w ramach inicjatywy Platformy Wsparcia Regionów Górniczych został sformalizowany i czy istnieje strategia współpracy w tym zakresie? Trzecie pytanie: Jakie są efekty spotkania z przedstawicielami Komisji Europejskiej podczas europejskiego forum gospodarczego w Katowicach? Dziękuję bardzo. Na pytanie odpowiada sekretarz stanu w Ministerstwie Energii, pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji węgla kamiennego pan minister Grzegorz Tobiszowski. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Panie i Panowie Posłowie! Dziękuję serdecznie panu posłowi za wywołanie tej kwestii, bo faktycznie trwają dość istotne prace nad zagospodarowaniem pierwszy raz terenów poprzemysłowych, głównie górniczych, w województwie śląskim.

Inicjatywa pierwotnie miała być pilotażowa dla naszego kraju, dla wsparcia procesów restrukturyzacyjnych.

Komisja uznała, iż ten program będzie poszerzony i stanie się programem dla innych krajów Unii Europejskiej, nadany mu zostanie charakter właśnie Platformy Wsparcia Regionów Górniczych nie tylko w Polsce. Rozpoczęło ono pewien dialog i wymianę dokumentów, informacji między stroną polską i Komisją Europejską.

W międzyczasie odbyły się spotkania robocze grup, które przygotowały te oficjalne spotkania.

Chodzi o przygotowanie i ocenienie przez Komisję Europejską tego, cośmy zgłosili, bo zgłosiliśmy 36 projektów.

Istotne jest, abyśmy zdążyli z projektami do 24 i 25 października, z zakończeniem, aby na COP-ie móc ogłosić, które projekty będą wsparte stosownymi środkami i ścieżką finansowania z Komisji Europejskiej. Od samego początku opiera się on na trzech szczeblach, poczynając od najwyższego, czyli corocznych spotkań wysokiego szczebla w Strasburgu - to jest grudzień 2017 r. - poprzez dialog ekspercki, czyli grupy robocze Komisji Europejskiej i strony polskiej, tzw. zespoły zadaniowe na szczeblu roboczym powołane do współpracy o charakterze bilateralnym, a więc chodzi o wymianę przygotowanych stosownych projektów i określenie, na jakim są etapie. Powiem tylko tyle, że projekty mają dwa kluczowe kryteria: szybkość inwestycji, szybkość stworzenia i realizacji takiego projektu, takiej inwestycji, jak również jego innowacyjność, a więc element pozwalający stworzyć nową jakość na terenach poprzemysłowych.

Jakie są efekty spotkań z przedstawicielami Komisji Europejskiej podczas europejskiego forum gospodarczego w Katowicach? To było ostatnie spotkanie. A więc przekazaliśmy i potwierdziliśmy te 36 projektów, które zostały przez nas przedłożone. Zostały one ocenione i zaplanowano, abyśmy w ramach takiego planu działania, action plan, otrzymali fiszki wedle sugestii i ram do wypełnienia przez Komisję Europejską. Teraz w lipcu, o czym wspominałem, 11 i 13 lipca odbędzie się spotkanie, na którym będziemy oceniać nasze projekty, niektóre połączone, doprecyzowane, abyśmy następnie mogli przejść do kolejnego etapu finansowania.

Dla nas ważne byłyby ścieżka finansowania, wielkość tego finansowania i kieszenie, w odniesieniu do których będziemy mogli wnioskować, jeśli chodzi o środki: czy to będzie dotacja, czy to będzie pożyczka. Weszliśmy w pewien bardzo istotny etap rozmowy precyzującej, jakie środki Komisja zaangażuje w ten projekt, jakie będzie mieć oczekiwania, jeśli chodzi o kraje, które wejdą do tego projektu.

Bardzo proszę o drugie pytanie. Dziękuję bardzo. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!

Pani Marszałek! Panie i Panowie Posłowie!

Pan minister Kwieciński bardzo mocno zaakcentował to, iż te projekty są wpisane w program dla województwa śląskiego, który jest elementem składowym programu odpowiedzialnego rozwoju premiera Morawieckiego, po czym omówiliśmy następny etap postępowania.

Dziękuję bardzo, panie ministrze. Przechodzimy do następnego pytania.

Pan poseł Tadeusz Aziewicz. Pani Marszałek! Szanowny Panie Ministrze! Od kilku tygodni nad polskim morzem znajdowane są martwe foki i morświny. Oględziny zwłok wskazują, że w istotnej części przypadków przyczyną może być bestialstwo człowieka. Odcięta płetwa ogonowa, rozcięcia w okolicy brzucha wykonane ostrym narzędziem, pętle na szyjach zwierząt to konkretne ślady aktywności zwyrodnialców. Wydarzenia te bulwersują opinię publiczną, która w znacznym stopniu łączy je z niefortunną kampanią posłanki PiS w dość specyficzny sposób nawołującą do zmniejszenia populacji fok w Polsce. Jednocześnie trwa wielka mobilizacja ludzi dobrej woli. Organizacje pozarządowe wyznaczyły nawet wysoką nagrodę za udzielenie informacji umożliwiających zidentyfikowanie i skazanie sprawców tych haniebnych czynów. W tej sytuacji dziwi milczenie i brak aktywności ministra, który jest w końcu odpowiedzialny za ochronę środowiska, w tym chronionych prawem gatunków. Panie Ministrze! Dotychczas nie usłyszeliśmy pańskiego głosu w obronie tych pięknych zwierząt. Nie widzę też realnych działań na rzecz zapobiegania kolejnym aktom bestialstwa. Przypominam, że dysponuje pan potężnym resortem z ogromnymi możliwościami, ma pan narzędzia, aby wpływać na stan świadomości zbiorowej, przekonując ludzi, że foki nie są szkodnikami, że polskie państwo chce i będzie bronić dalszego istnienia tego gatunku. Niestety, w trakcie spotkania w Mławie stwierdził pan, że żyjemy w czasach nadmiernej wrażliwości w ochronie zwierząt. Mocno podważa to pańską wiarygodność jako obrońcy chronionych gatunków, dlatego z niepokojem pytamy: Co zamierza pan zrobić, aby powstrzymać proces mordowania fok i morświnów na polskim Wybrzeżu? Czy rozważa pan przyjęcie programu ochrony foki szarej złożonego w Ministerstwie Środowiska w 2012 r., który zawiera bardzo konkretne rekomendacje? Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo.

przyjął również program ochrony morświna, który kompleksowo zajmuje się zagrożeniami dla tego gatunku oraz metodami przeciwdziałania tym zagrożeniom. W tym dokumencie porusza m.in. kwestie przypadkowego przyłowu morświna w sieci rybackie, stosowania urządzeń odstraszających te zwierzęta, testowania alternatywnych narzędzi rybackich, które są bezpieczne dla morświna. Wiemy, że jeśli chodzi o ten gatunek, dzisiaj populacja jest szacowana na ok. 500 sztuk i jest uznana za populację krytycznie zagrożoną. Jeśli chodzi o foki, to w ministerstwie trwają prace nad planami ochrony obszarów morskich Natura 2000. Przyjęcie tych planów powinno efektywnie zabezpieczyć kluczowe siedliska foki szarej w obszarach, w których ten gatunek jest przedmiotem ochrony. Warto podkreślić, że w odróżnieniu od programów ochrony gatunków, które są dokumentami miękkimi, plan ochrony dla obszarów Natura 2000 zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska będzie stanowił akt mający moc aktów prawa powszechnie obowiązującego.

Dziękuję bardzo, pani minister. Bardzo proszę pana posła Adama Korola o drugie pytanie. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Z niepokojem przyjęliśmy ostatnie wypowiedzi pana ministra Kowalczyka na spotkaniu w Mławie, który powiedział - chciałem zacytować kilka rzeczy, o których mówił pan minister - że żyjemy w czasach nadmiernej wrażliwości w ochronie zwierząt.

Moje pytanie jest takie: Czy tego rodzaju myślenie ma dotyczyć również fok? Bo foka, jak wiemy, również jest zwierzęciem chronionym. Dobrze pan minister wie, że to nie jest rozwiązanie problemu, [[Dzwonek]] gdyż w miejsce odstrzelonego osobnika zaraz pojawi się następny.

Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz proszę panią minister Małgorzatę Golińską o odpowiedź na pytania. Panie Pośle!

Wysoki Sejmie! Jednym z najważniejszych i najmocniejszych punktów programu rządu Prawa i Sprawiedliwości jest niewątpliwie polityka rodzinna. Wszyscy cieszymy się z programu „Rodzina 500+”, który w znaczący sposób wspiera i wzmacnia rodziny z dziećmi na utrzymaniu, dając im poczucie bezpieczeństwa, którego wcześniej nie miały. Kontynuacją tego dobrego kierunku jest zapowiedziany przez pana premiera Mateusza Morawieckiego rządowy program „Dobry start”, dzięki któremu rodzice otrzymają dodatkowe finansowe wsparcie na pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o przedstawienie szczegółowych danych na temat przygotowania do realizacji programu „Dobry start” Wiemy, że program realizują gminy, te same urzędy, które zajmują się przyjmowaniem wniosków do programu „Rodzina 500+” Czy gminy są dobrze przygotowane do tego zadania? Czy ministerstwo nie obawia się kolejek w urzędach? Jak wygląda kwestia finansowania oraz jak ministerstwo rodziny wspiera samorząd w przygotowaniach do startu „Dobrego startu” Dziękuję. Bardzo proszę podsekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pana ministra Bartosza Marczuka o odpowiedź na pytania. Pani Marszałek! Panie Pośle! Tak, rzeczywiście jest tak, że program ruszył czy nabór wniosków ruszył od niedzieli. Wzorem tego, co zrobiliśmy przy okazji programu 500+, postaraliśmy się o to, aby bardzo dobrze przygotować samorządy do obsługi tego programu zarówno od strony organizacyjnej, jak i od strony finansowej. Chciałbym tylko zaznaczyć, że to był dość krótki czas, ponieważ informacja o programie pojawiła się w kwietniu, kiedy ogłosił to pan premier Mateusz Morawiecki, natomiast 1 lipca.

Uruchomiliśmy specjalną stronę internetową czy zakładkę na naszej stronie internetowej.

Ona jest dedykowana samorządom.

Pomyśleliśmy też o tym, by gmin nie obciążać nadmiernie pracą.

Kanał bankowy też jest bardzo istotny.

Jeszcze jedna rzecz: kierownictwo zarówno ministerstwa rodziny, jak i Ministerstwa Edukacji Narodowej wyjechało do wszystkich województw i konsultowało ten program w czerwcu, jeszcze przed jego startem. Można opowiadać o tym, co zrobiliśmy, ale tak naprawdę liczy się na koniec dnia to, jak to wszystko zagrało czy nie zagrało.

Żadnych problemów zgłaszanych przez gminy, żadnych problemów w naszych systemach informatycznych.

Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę pana posła Wojciecha Buczaka o zadanie kolejnego pytania. Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Bardzo dziękuję za odpowiedź na pierwszą część pytania. Też przy okazji naprawdę wielkie uznanie za to, jak program został przygotowany, zarówno poprzedni, „Rodzina 500+”, jak i obecny, „Dobry start”, a szczególnie za to wsparcie, solidarną pomoc ze strony rządu, ministerstwa dla samorządów.

A jeśli są jakieś z tej strony zacięcia czy opóźnienia, to prosiłbym o informację.

Jak jest w przypadku programu „Dobry start”

Dziękuję bardzo. I jeszcze raz proszę pana ministra Bartosza Marczuka o udzielenie odpowiedzi. Panie Pośle! Jeżeli chodzi o samorządy, to my tutaj mówimy, podobnie zresztą jak przy okazji programu 500+, że bardzo szanujemy ich pracę, bardzo dziękujemy za to, że te samorządy, co do zasady oczywiście, chcą z nami współpracować. One też wiedzą i czują, że te świadczenia, które wypłacają, są potrzebne lokalnie, zwłaszcza w tych mniejszych czy najmniejszych miejscowościach. Nasze doświadczenia z programu 500+, tak jak wspomniałem, przenieśliśmy, jeżeli chodzi o współpracę z samorządami, właśnie do programu „Dobry start”, czyli podręcznik, informacja, infolinie, akcja informacyjna, konsultacje w regionach.

Niejako szanując pracę tych ludzi, którzy są tam, na dole, i którzy bezpośrednio zajmują się obsługą tych wniosków, wprowadziliśmy taką zasadę, że te pieniądze, które płacimy samorządom za obsługę - a przypomnę, że to jest 3% całej kwoty programu - są w 80% dedykowane tym pracownikom.

Tak że to jest takie novum i zobaczymy, jak to się sprawdzi, jak to będzie działać.

To jest 10 zł za jeden obsłużony wniosek, bo to jest zadanie zlecone przez rząd, czyli 8 zł, a zatem 80% tych pieniędzy, trafia czy ma trafić bezpośrednio do kieszeni ludzi, którzy zajmują się obsługą tych wniosków. Sam projekt rozporządzenia, który wprowadza program „Dobry start” Tak że szacunek dla samorządów, płacimy samorządom, podobnie jak przy programie 500+, za obsługę tych wniosków, jest nowe rozwiązanie związane z wynagrodzeniem bezpośrednio trafiającym do ludzi.

Dziękuję bardzo, panie ministrze. Przechodzimy do następnego pytania. Pytanie zadają posłowie Anna Czech i Witold Czarnecki, Prawo i Sprawiedliwość, w sprawie działań podejmowanych w zakresie walki z dopalaczami - pytanie do ministra zdrowia. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Dziękuję serdecznie Ministerstwu Zdrowia, że w odpowiedzi na interpelację w sprawie zmiany ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w części dotyczącej definicji nowych środków psychoaktywnych oraz części uprawnień m.in. Państwowej Inspekcji Sanitarnej zostały zadeklarowane oraz podjęte konkretne działania. Powstał projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, zdefiniowano w kierunku ujednolicenia i objęcia przepisami karnymi czyny związane z dystrybucją tzw. dopalaczy. Problem z dopalaczami, jak wiemy, to głównie ciągle modyfikowany skład chemiczny. Handlarze wprowadzają na rynek coraz to nowe, coraz bardziej niebezpieczne substancje. W ten sposób próbują ominąć listę substancji kontrolowanych prawem. Czy i jak zmiana ustawy zakłada radzenie sobie z tym problemem? Ponadto nie ma już oficjalnych, normalnych lub paranormalnych sklepów, które oferują dopalacze, a jeśli policja zidentyfikuje tego typu placówki, natychmiast je zamyka. Natomiast handel dopalaczami zszedł do tzw. podziemia.

Dziękuję bardzo. I bardzo proszę podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia pana Zbigniewa Józefa Króla o udzielenie odpowiedzi. Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Tytułem wprowadzenia, bo dużo było powiedziane na temat problemów, które mamy, i modyfikacji tej dystrybucji.

Mamy mniej więcej 11 przypadków zatruć w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców.

Czyli, po pierwsze, nowe substancje psychoaktywne mają być objęte kontrolą analogiczną jak w wypadku środków odurzających i substancji psychotropowych, pozostawienie odpowiedzialności administracyjnej w zakresie środków zastępczych, tylko przesunięcie w tej chwili ilości, środki zastępcze to są głównie dopalacze, przesuwamy to do narkotyków i środków zastępczych zostanie zdecydowanie mniej. One muszą być ujawnione, muszą być wskazane przez odpowiedni zespół, który działa już kilka lat. Kwestia nadzoru nad środkami zastępczymi nie ulega zmianie. Natomiast substancje w nich identyfikowane będą podlegały ocenie zespołu ds. oceny ryzyka zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzi.

Chcemy, żeby po prostu te substancje identyfikowane jako środki psychoaktywne były tam wpisywane. Dodatkowo zgodnie z przepisami w projektowanej ustawie dopalacze mają być traktowane na równi z narkotykami. Przywóz, wywóz, przewóz, wewnątrzwspólnotowe nabycie lub wewnątrzwspólnotowa dostawa nowych substancji psychoaktywnych będą podlegały grzywnie, karze ograniczenia wolności oraz pozbawienia wolności, tutaj proponujemy do 5 lat, czyli takiej samej jak w wypadku substancji psychotropowych.

Poza tym dyrektywa unijna wskazuje, że powinniśmy w naszej ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii dokonać zmian dotyczących całego rynku wewnątrzwspólnotowego, nie tylko zajmować się obszarem polskim.

Należy podkreślić, że zasadniczym celem tej ustawy jest objęcie przepisami karnymi przede wszystkich czynów związanych z dystrybucją tych substancji i stworzenie instrumentów prawnych umożliwiających pociągnięcie do odpowiedzialności osób z nią związanych.

Serdecznie witamy was w Sejmie. A teraz oddaję głos pani poseł Annie Czech. Dziękuję bardzo, pani marszałek. Dziękuję za podjęcie skutecznych, miejmy nadzieję, działań i za wyczerpującą odpowiedź w pierwszej części.

Czy Ministerstwo Zdrowia planuje rozwinąć ten program w kolejnych latach nie tylko poprzez przeznaczanie coraz większych środków, ale też poprzez inspirowanie do coraz ciekawszych programów, poprzez ogłaszanie konkursów ofert, różnego rodzaju programów profilaktycznych, programów, które pogłębiają wiedzę i dosadnie trafiają do młodzieży, rodziców, a także wychowawców? Dziękuję bardzo. Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Obserwujemy, że problem dopalaczy jest w ogóle niezidentyfikowany w społeczeństwie.

Główny Inspektor Sanitarny doprowadził do utworzenia i funkcjonowania punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, administruje również funkcjonowaniem całodobowej linii będącej w dyspozycji stacji sanitarno-epidemiologicznych, tak aby w każdej chwili można było się skontaktować z perspektywy nie tylko czasami dramatycznych sytuacji na szpitalnych oddziałach ratunkowych, ale również rodziców, również osób, które w swoim otoczeniu dostrzegają ten problem. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Przechodzimy do następnego pytania. Pytanie zadają państwo posłowie Gabriela Masłowska, Czesław Sobierajski i Barbara Bubula, Prawo i Sprawiedliwość, w sprawie sytuacji najemców byłych mieszkań zakładowych i efektów prac legislacyjnych zrealizowanych w tym zakresie przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, które weszły w życie w maju 2018 r. - do ministra inwestycji i rozwoju. Bardzo proszę, pytanie zadaje pani poseł Gabriela Masłowska.

Część tych najemców nadal mieszka w tych mieszkaniach i dopomina się o wyrównanie tego rachunku krzywd. W poprzednich dwóch kadencjach wykonaliśmy ogromną pracę, wraz ze środowiskami najemców, związaną z rozwiązaniem tego problemu, który był przez wiele rządów i przez wiele kadencji pomijany i niechętnie traktowany.

Cały ten cały dorobek przekazałam na początku tej kadencji ministerstwu, uważając, że jest to już jakaś poważna baza w kierunku kontynuacji procesu prac nad ustawą.

Chodzi przynajmniej o część tych najemców, bo pewnie wszystkich nie zadowolimy. Czy pan minister mógłby się odnieść do tego, na jakim etapie są te prace? Bardzo proszę, sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju pan Artur Soboń. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Poseł! Chcę potwierdzić tę trudną sytuację wielu lokatorów mieszkań zakładowych, ponieważ nieruchomości zabudowane tymi mieszkaniami z dniem 5 grudnia 1990 r. zostały z mocy prawa przekazane na własność przedsiębiorstwom państwowym. Fakt uwłaszczenia tych przedsiębiorstw wpłynął na ukształtowanie sytuacji prawnej najemców mieszkań usytuowanych na przekazanych gruntach. Uwłaszczone przedsiębiorstwa mogły w latach 90. dowolnie rozporządzać przekazanym mieniem bez obowiązku informowania najemców mieszkań, ponieważ aż do dnia 7 lutego 2001 r. nie istniały żadne regulacje przyznające najemcom prawo pierwszeństwa w nabyciu mieszkania. Część tych najemców ma już uregulowaną sytuację, znaczna część jednak nie ma. To, co zaproponowaliśmy dotychczas, to coś, z czego za chwilę samorządy będą mogły skorzystać.

Wśród tych zmian w zakresie finansowego wsparcia budownictwa komunalnego uwzględniono postulaty podmiotów wspierających mieszkańców byłych mieszkań zakładowych poprzez następujące rozwiązania. Po pierwsze, zwiększenie bezzwrotnego finansowego wsparcia dla gmin z Funduszu Dopłat na kupno lub kupno połączone z remontem byłych mieszkań zakładowych lub budynku mieszkalnego z byłymi mieszkaniami zakładowymi z 30% do 50% kosztów przedsięwzięcia, a także brak zakazu zbywania lokali mieszkalnych z zasobu mieszkaniowego gminy w przypadku, gdy przedmiotem zakupu jest byłe mieszkanie zakładowe lub budynek z byłymi mieszkaniami zakładowymi. Krótko mówiąc, gmina może dostać 50% finansowania i jednocześnie udzielić bonifikaty, która byłaby dla tych lokatorów adekwatna i możliwa do sfinansowania. W ustawie o finansowym wsparciu zdefiniowano, że przez byłe mieszkania zakładowe należy rozumieć mieszkania stanowiące przed dniem 7 lutego 2001 r. własność przedsiębiorstw państwowych i spółek handlowych, w których Skarb Państwa był podmiotem dominujących w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Tym samym regulacja nie dotyczy mieszkań, które obecnie stanowią mienie przedsiębiorstw państwowych. Ponadto finansowe wsparcie będzie udzielone pod warunkiem, iż osoby, które przed 7 lutego 2001 r. były pracownikami przedsiębiorstwa państwowego lub spółki handlowej, w których Skarb Państwa był podmiotem dominującym w rozumieniu tejże ustawy, a także wstępni, zstępni, małżonek najemcy, osoby przysposabiające i przysposobione oraz osoby, które pozostawały z najemcami w faktycznym wspólnym pożyciu, zamieszkujące w chwili śmierci z najemcą, które wstąpiły w stosunek najmu po śmierci osób wskazanych w pkt 1, które wymieniłem jako osoby, jako tych byłych pracowników przedsiębiorstw państwowych. Jednocześnie chcę powiedzieć, że wnioski o wykup tych mieszkań zakładowych gminy będą mogły składać do Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach najbliższej edycji programu, czyli od 1 lipca do 30 września. Natomiast od 2019 r. wnioski te będą składane w trybie ciągłym aż do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na dany rok.

Natomiast w ramach edycji, która rozpoczyna się już 1 lipca, oczywiście na wszystkie zadania Tyle chcemy przeznaczyć w tym okresie pomiędzy lipcem a wrześniem. Chcemy ocenić, jakie to przyniesie skutki w zakresie rozwiązania tego problemu, o którym mówi pani poseł. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani poseł Gabriela Masłowska. To, o czym pan mówi, te wprowadzone rozwiązania stanowią jakiś mały kroczek w rozwiązaniu tego całego bolesnego, powiedziałabym, okropnego problemu wielu tysięcy ludzi, ale dotyczą tylko pewnej grupy osób. Dotyczą takich sytuacji, kiedy gmina chce nabyć to mieszkanie, bo dopłaty, jak pokazuje doświadczenie, dla gmin na ten cel, które poprzednio wynosiły 30% czy 35%, nie bardzo uruchamiały, nie stwarzały bodźców dla gmin, żeby się zainteresowały wykupem tego mieszkania. Nie sądzę, żeby to było taką zachętą, żeby gminy zdecydowały się kupować te mieszkania.

Pani Marszałek! Pani Poseł!

Wymieniam go, ponieważ on już prowadzi z nami intensywne rozmowy. Ono oczywiście ma mankamenty, ale w tej sprawie - jak pani poseł też doskonale wie, bo mało kto wie o tej sprawie tak dużo jak pani poseł - idealnego rozwiązania nie ma.

To nie jest łatwe, bo te podmioty, które dzisiaj są właścicielami tych mieszkań, to bardzo często ich kolejni właściciele. Moja propozycja jest taka, abyśmy zobaczyli, czy będzie zainteresowanie ze strony samorządów, i jednocześnie zaproponowali rozwiązania systemowe. Myślę, że on jest dobrą podstawą do tego, aby wypracować rozwiązanie systemowe, choć oboje, jak rozumiem, zachęcamy gminy do tego, aby korzystały z tego instrumentu wsparcia, jakim jest Fundusz Dopłat BGK. Bardzo dziękuję. Przechodzimy do następnego pytania.

Bardzo proszę, pytanie pierwsze zadaje pan poseł Bogusław Sonik. Dziękuję. Panie Ministrze! Pytanie dotyczy wdrażania bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, w skrócie zwanej BDO. Szanowny Panie Ministrze!

Biorąc pod uwagę oczywisty fakt, że przejrzysty i w pełni kontrolowany obrót, przemieszczanie odpadów jest warunkiem osiągnięcia tego celu, proszę o odpowiedź na pytanie o stan wdrażania najważniejszego w tym procesie narzędzia, mianowicie bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach przewidywała utworzenie jej w terminie do 23 stycznia 2016 r., tj. 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Realizując zapisy ustawy, w roku 2015 minister środowiska wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zaprojektowanie, wytworzenie i wdrożenie systemu informatycznego pn. Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami”

Jakie kontrakty, na jakie kwoty i na jakiej podstawie prawnej zostały zawarte przez Ministerstwo Środowiska lub podległe mu instytucje? Przypomnę tylko, że pan minister na posiedzeniu komisji mówił, że ministerstwo [[Dzwonek]] będzie to realizować własnymi siłami. Dziękuję bardzo. Na pytanie odpowie podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska pan minister Sławomir Mazurek.

Pani Marszałek! Panie i Panowie Posłowie! Odpowiadając na pytanie pana posła, nie sposób uciec od potrzeby wyjaśnienia ostatnich słów, które pan poseł wypowiedział, mówiąc, że baza danych odpadowych nie jest realizowana. Pragnę na wstępie powiedzieć, że ministrowi środowiska - użyję sformułowania, którego użyła pani poseł Lenartowicz na posiedzeniu komisji - bardzo mocno zależało, w momencie gdy przyszliśmy do ministra środowiska, aby baza danych odpadowych nie była atrapą, nie była kolejnym, bardzo drogim Excelem, ale narzędziem, którego wcześniej nie było, a o którym mój poprzednik w jednej z komisji senackich powiedział, że na to nie są gotowi ani przedsiębiorcy, ani systemy informatyczne, ani inspekcje.

To faktycznie będzie bardzo sprawne narzędzie wykorzystujące najnowsze technologie, które są dostępne na rynku informatycznym, łącznie z tymi najnowszymi, innowacyjnymi rozwiązaniami.

Wpisowi do rejestru podlegają wszystkie podmioty działające w zakresie gospodarki odpadami. Rejestr BDO stanowi, tak jak powiedziałem, pierwszy element bazy danych o produktach oraz o gospodarce odpadami.

Pełne uruchomienie wszystkich funkcjonalności BDO umożliwi skuteczną kontrolę rynku gospodarki odpadami, zgodnie z tym też, co powiedział pan przewodniczący, przyczyni się do efektywniejszego wspierania organów Inspekcji Ochrony Środowiska w walce z nieprawidłowościami występującymi w tym sektorze. Ponadto dzięki BDO organy kontroli będą mogły analizować jednocześnie zgodność faktycznie prowadzonej przez podmioty działalności w zakresie gospodarki odpadami z zakresem zadeklarowanym w rejestrze.

Dodatkowo ze względu na fakt, że organy Inspekcji Ochrony Środowiska będą miały zapewniony dostęp do BDO, umożliwi im to kontrolę ewidencji odpadów, która prowadzona będzie przez podmioty wyłącznie za pomocą dedykowanego w bazie modułu. Powinno się to przyczynić do wyeliminowania nielegalnego przekazywania odpadów wraz z niewłaściwym sposobem ich ewidencjonowania, jakie może występować w przypadku ewidencji prowadzonej w sposób tradycyjny, w formie papierowej. Obecnie w Ministerstwie Środowiska trwają prace nad utworzeniem kolejnej funkcjonalności, tak jak powiedziałem, zgodnie z tą metodą zwinną. Chodzi o opracowanie dokumentacji do przetargu na wyłonienie wykonawcy BDO.

Zamówienie dotyczące rejestru już zostało udzielone specjalistycznej firmie na podstawie Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z obowiązującymi w Ministerstwie Środowiska procedurami udzielania zamówień publicznych. Natomiast aktualnie prowadzony jest dialog techniczny poprzedzający przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i opisu przedmiotu zamówienia dla postępowania dotyczącego realizacji kolejnych etapów. Planuje się ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych w październiku tego roku.

Na bieżąco też odpowiadamy na wszelkie pytania w tej dziedzinie. Dziękuję także za zainteresowanie pani poseł, pana posła tym tematem, ponieważ będzie to sprawne narzędzie, które wspomoże Inspekcję Ochrony Środowiska w tym bardzo ważnym procesie, nad którym dzięki zaangażowaniu osobistemu pana premiera, pana ministra Kowalczyka mogliśmy przyspieszyć prace mające na celu walkę z patologiami w gospodarce odpadami. BDO na pewno tu pomoże. Jednak również pragnę państwa poinformować, że pod kierunkiem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pracuje specjalny zespół i zostały przygotowane specjalne rekomendacje, które po zakończeniu prac też będą ogłoszone. Bardzo dziękuję. I bardzo proszę panią poseł Gabrielę Lenartowicz o zadanie dodatkowego pytania.

Wszystkim nam pan opowiadał, że będzie to robione własnymi siłami ministerstwa. Teraz już pan mówi, że to jest wspomagane zewnętrznie i wymienił pan jedną firmę, w interpelacji nawet z nazwy, zatrudnioną za sto pięćdziesiąt parę tysięcy złotych podobno. A pozostałe moduły, jak pan mówi, już, jak się okazuje, chyba nie będą jednak wdrażane zwinnie przy pomocy pracowników, bo przygotowujecie jakiś dialog techniczny jednak na dokumentację do przetargu.

dziewięć, dziesięć umów w Ministerstwie Środowiska. tejże bazy. I bardzo proszę pana ministra o udzielenie odpowiedzi na pytania.

Sprawdzę dokładnie kwestie związane z umowami. Na pewno wyjaśnimy wszelkie pani wątpliwości na piśmie z tego względu, że oczywiście dla ministra środowiska jest to projekt bardzo ważny, kluczowy, jeśli chodzi o gospodarkę odpadami.

Chcę powiedzieć, że jeśli chodzi o środki, które zostały wydane, to jest to 153 504 zł brutto. I to są te środki, które wynikają z potrzeby wspomożenia Ministerstwa Środowiska w zakresie przygotowania tego pierwszego elementu, który został uruchomiony.

Jestem członkiem komitetu cyfryzacji i pragnę pani powiedzieć, że to jest innowacyjna metoda. Być może pani jej nie zna, dlatego wyjaśnię. To pani niestety nie do końca chyba mnie rozumie, ponieważ metoda zwinna w żaden sposób nie wyklucza używania narzędzi w postaci zamówień publicznych. Ten rząd jest rządem przejrzystym, wszystkie informacje są dostępne. Procedura zamówień publicznych jest narzędziem takim, które umożliwia przejrzyste działanie. I na pewno takich procedur jako rząd ten rząd będzie się trzymał. Jednocześnie bardzo nam zależy na tym, żeby wykorzystywać najnowsze technologie, które pozwolą na optymalizację kosztów i skuteczność działań. Na pewno tego się będziemy trzymać.

To pytanie kończy rozpatrywanie tego punktu porządku dziennego. Przypominam, że na obecnym posiedzeniu Sejmu zostanie rozpatrzona informacja w sprawie przygotowania pilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary oraz sposobu procedowania nad nim, o której przedstawienie wnosił klub Kukiz’15. Przypominam również, że przedstawienie uzasadnienia wniosku przez posła przedstawiciela wnioskodawców nie może trwać dłużej niż 5 minut, a udzielenie odpowiedzi przez przedstawiciela Rady Ministrów - dłużej niż 10 minut. Wystąpienia posłów w dyskusji nie mogą trwać dłużej niż 2 minuty. Na zakończenie dyskusji głos zabierają kolejno przedstawiciel wnioskodawców oraz przedstawiciel Rady Ministrów. Wystąpienie przedstawiciela wnioskodawców nie może trwać dłużej niż 5 minut, a wystąpienie przedstawiciela Rady Ministrów - dłużej niż 10 minut. Marszałek Sejmu może wyrazić zgodę na wydłużenie wystąpienia przedstawiciela Rady Ministrów. Proszę o zabranie głosu przedstawiciela wnioskodawców pana posła Tomasza Rzymkowskiego. Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Po pierwsze, bardzo dziękuję za zgodę na przedstawienie informacji bieżącej w zakresie okoliczności dotyczących przygotowania oraz uchwalenia ustawy z dnia 27 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Mianowicie chodzi o zwykłą notatkę prasową, która została przedłożona jako, powiedzmy, zadośćuczynienie za to, że polski parlament pod dyktando innego państwa przyjął ustawę. Dlatego przejdę od razu do kluczowych, podstawowych pytań dotyczących całego spektrum wydarzeń towarzyszących nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej.

Kolejna rzecz dotyczy zainicjowania negocjacji, które sfinalizowały się rzeczonego 27 czerwca, czyli w ubiegłym tygodniu, w środę. Czy prawdziwe są informacje medialne, jakoby ze strony izraelskiej rozmowy były prowadzone przez funkcjonariuszy Mosadu?

Czy była jakaś groźba ze strony państw trzecich, jeśli nie zmienimy tej ustawy, a tym samym nie przyjmiemy nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej? Kolejna kwestia dotyczy samego trybu procedowania nad ustawą.

Ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej jest właśnie taką ustawą. Kolejna rzecz, która poprzedza w ogóle dyskusję na temat dyspozycji art. 123 ust. 1, dotyczy tego, czy była uchwała Rady Ministrów w sprawie nadania trybu pilnego przedmiotowemu projektowi ustawy rządowej.

Czy to świadczy o suwerenności polskiego Sejmu, Senatu, prezydenta i przede wszystkim rządu, który w taką retorykę wchodzi? Jesteśmy w przededniu rocznicy ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej.

Proszę o udzielenie odpowiedzi sekretarza stanu, szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pana Michała Dworczyka.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Po pierwsze, odpowiadając na pytanie pana posła, chciałbym zwrócić uwagę, że jesteśmy w parlamencie. Można tutaj powiedzieć niemal wszystko, ale rzeczywiście w tych naszych wypowiedziach, panie pośle. w tych naszych wypowiedziach, panie pośle - przepraszam, chciałem pozwolić panu dokończyć, bo jednak odnoszę się do pańskiej wypowiedzi, więc chciałbym, żeby pan usłyszał te słowa - trzeba mieć jednak pewien umiar. Sugerując, że polski rząd i polski parlament działają pod dyktando obcego państwa, obcych wywiadów, obraża pan nie tylko obecny rząd, ale też cały parlament i siebie również. To jest po prostu wierutna bzdura i namawiam pana, bo jest pan osobą wyważoną, rozsądną, żeby w tej krytyce, skądinąd często słusznej, jednak zachować umiar i adekwatnie odnosić się do sytuacji. W tym wypadku przekroczył pan tę granicę.

To wybrzmiało już kilkakrotnie z tej trybuny. Nie doceniliśmy tak naprawdę zaniedbań, które przez kilkadziesiąt lat miały miejsce, jeśli chodzi o dbałość o polskie imię, o dobre imię narodu polskiego poza granicami kraju. Wiedzieliśmy, że ten temat leżał odłogiem, wiedzieliśmy, że polski rząd, zdarzało się, prowadził przeciwskuteczne działania, jeżeli chodzi o budowanie dobrego wizerunku naszego kraju poza granicami Polski - i tutaj przykład, który już podawałem, promowanie Polski poprzez emitowanie takich filmów jak „Pokłosie” w instytutach polskich albo promowanie książek pana Grossa przez instytuty polskie, to są właśnie przykłady z lat rządów Platformy Obywatelskiej, w cudzysłowie, promocji Polski poza granicami, więc zgoda, nie było tej polityki, nie było tej dbałości o wizerunek naszego kraju za granicą - ale rzeczywiście nie doceniliśmy tego, jak daleko te zmiany w świadomości społecznej zaszły.

dlatego taki huraganowy atak, i dlatego nasza odpowiedź, która jednak była, bo przypomnę i dużą kampanię promocyjną - niewłaściwe sformułowanie - dużą kampanię informacyjną przeprowadzoną za granicą jeszcze w lutym i w marcu przez rząd, i działania naszej dyplomacji prowadzone za pośrednictwem ambasad, konsulatów, instytutów polskich. Ale rzeczywiście ten atak był zmasowany i nie doceniliśmy skali zaniedbań. W tym względzie trzeba panu posłowi przyznać rację. Ale nie można zgodzić się z tezą, że byliśmy nieprzygotowani albo że rząd nie podejmował działań, które miały na celu skuteczne poinformowanie zagranicznej opinii publicznej o sytuacji związanej z nowelizacją ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Kto uczestniczył w negocjacjach nad nowelizacją ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej? Nikt, panie pośle, bo nie było żadnych negocjacji.

Jak rozumiem, myli się panu ustawa z oświadczeniem podpisanym przez premierów, premiera Mateusza Morawieckiego i premiera Netanjahu. Tu rzeczywiście toczyły się rozmowy na temat wspólnego oświadczenia - oświadczenia, które pan deprecjonuje, nazywając je notatką prasową. A ja jednak namawiam pana do takiej pogłębionej analizy, ponieważ w naszym przekonaniu ten dokument jest szalenie ważny. Szalenie ważny jest on nie tylko ze względu na jakiś tam bieżący efekt polityczny, ale także ze względu na przyszłą strategiczną i długofalową politykę państwa polskiego i zabieganie o dobry wizerunek i dobre imię narodu polskiego na forum międzynarodowym.

Po raz pierwszy premier Izraela przyznaje, jak duża była rola Polskiego Państwa Podziemnego w zwalczaniu niemieckiego okupanta, w ratowaniu Żydów, w działaniach na rzecz odzyskania niepodległości przez Polskę. Po raz pierwszy jest tak jasno sformułowane w takim dokumencie, kto był rzeczywiście sprawcą i II wojny światowej, i Holokaustu, i wyraźnie są tutaj wskazane faszystowskie Niemcy. Ten dokument z punktu widzenia przyszłych działań wizerunkowych, ale również procesowych jest, uważam, bardzo ważny i naprawdę nie warto go deprecjonować. A jeśli chodzi o wypracowywanie treści tego oświadczenia, to odpowiadam panu, że tutaj prowadził te rozmowy. W kilku długich rozmowach telefonicznych z premierem Netanjahu omawiane były poszczególne elementy tego dokumentu. Ale podkreślę jeszcze raz, bo to wybrzmiało w pierwszej części pańskiego pytania: Dokument, oświadczenie, czyli ten dokument, o którym przed chwilą mówiłem, i nowelizacja ustawy, te dwie rzeczy nie są ze sobą związane, choć oczywiście były tego samego dnia opublikowane. Żyjemy w wolnym kraju, wbrew temu, co niektórzy twierdzą, więc może pan poseł wierzyć, może pan poseł nie wierzyć. Ja odpowiadam zgodnie z moją najlepszą wiedzą na temat tej sytuacji. Jeśli chodzi o tryb, bo zapytał pan poseł o tryb i podawał w wątpliwość to, w jaki sposób została przeprocedowana ta ustawa - to są sprawy prawne. Pan jest prawnikiem, ja jestem historykiem, w związku z tym pozwoli pan, że będę się wspierał notatką. którą prosiłem, żeby sporządził departament prawny, aby panu precyzyjnie odpowiedzieć na to pytanie.

Na podstawie § 98 Regulaminu pracy Rady Ministrów prezes Rady Ministrów zdecydował o odrębnym trybie postępowania z przedmiotowym projektem ustawy, polegającym na wniesieniu tego projektu bezpośrednio do rozpatrzenia przez Radę Ministrów w trybie obiegowym. Tym samym nie było obowiązku przeprowadzenia konsultacji publicznych ani uzgodnień międzyresortowych w odniesieniu do tego projektu. W dniu 26 czerwca szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów skierował pismo do sekretarza Rady Ministrów z prośbą o niezwłoczne skierowanie przedmiotowego projektu ustawy do rozpatrzenia przez Radę Ministrów w trybie obiegowym, jednocześnie wnosząc o uznanie przedmiotowego projektu ustawy za pilny w rozumieniu art. 123 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na konieczność podjęcia niezwłocznych działań służących bardziej efektywnej ochronie dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej i narodu polskiego. Projekt ten został niezwłocznie przedłożony członkom Rady Ministrów do rozpatrzenia w trybie obiegowym i wobec niezgłoszenia uwag w wyznaczonym terminie, tj. do godz. 22 tego samego dnia, na podstawie § 92 ust. 4 Regulaminu pracy Rady Ministrów uznany za przyjęty przez Radę Ministrów jako projekt pilny. Projekt ustawy został następnie przesłany przez prezesa Rady Ministrów na ręce marszałka Sejmu RP z informacją, iż Rada Ministrów uznała wymieniony projekt ustawy za pilny ze względu na konieczność podjęcia niezwłocznych działań służących itd. Na podstawie art. 123 konstytucji Rada Ministrów może uznać uchwalony przez siebie projekt ustawy za pilny, z wyjątkiem projektów ustaw podatkowych, ustaw dotyczących wyboru prezydenta RP, Sejmu, Senatu oraz organów samorządu terytorialnego, ustaw regulujących ustrój i właściwość władz publicznych, a także kodeksów. Krótko mówiąc, w żadnym z tych katalogów ta nowelizacja się nie znalazła, więc mogła być uznana za pilną. Projekt ustawy o zmianie ustawy o IPN mógł być uznany przez Radę Ministrów za pilny, gdyż w szczególności nie regulował ustroju ani nie ingerował w pozostałe obszary. Podsumowując, przedmiotowy projekt ustawy został przygotowany przez Radę Ministrów w zgodzie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i Regulaminem pracy Rady Ministrów. Mam nadzieję, że to jest w miarę wyczerpująca odpowiedź dla pana posła. Wie pan co, nie spodziewałem się po panu tego pytania a propos Wołynia.

Czy ktoś z pań i panów posłów pragnie jeszcze zapisać się do głosu? Otwieram dyskusję. Bardzo proszę o zadanie pytania pana posła Waldemara Budę z Prawa i Sprawiedliwości. Czas wystąpienia - 2 minuty. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pan poseł skupił się na technikaliach, czyli na wskazywaniu na potencjalne nieprawidłowości, co nie potwierdziło się, i mamy tego pewność, to wynika z tej notatki, którą pan minister przytoczył. Natomiast w mojej ocenie trzeba się skupić w tej sprawie na rzeczy najważniejszej, to znaczy, miarą działania są skutki i efekty i ja bym chciał zapytać pana ministra właśnie o te efekty i skutki ustawy wprowadzonej w czerwcu, bo dla mnie te skutki są oczywiście pozytywne i nie mam żadnych wątpliwości w tym zakresie. Gdybyśmy mogli w jakiejś części, bo wiadomo, temat jest rozległy, przeanalizować właśnie te skutki na arenie międzynarodowej, to byłbym bardzo wdzięczny. Dziękuję. Pan poseł Bogusław Sonik, Platforma Obywatelska. Panie Ministrze! Odnosząc się do sprawy tej ustawy, chciałbym powiedzieć, że przypomina to zwyczaje niektórych strażaków ochotników, którzy podpalają domostwa czy łąki, a potem biorą bohatersko udział w ich gaszeniu. Mówię o przestępcach, proszę pana, którzy to realizują. W związku z tym pytanie jest jasne. Powierzono negocjowanie tak ważnej ustawy w sposób skandaliczny, wprowadzono ją w sposób taki, że można by to nazwać podwórkową dyplomacją, która w żaden sposób nie zorientowała się, jakiej wagi sprawę negocjuje. Pytanie jest: Czy są mechanizmy, które w tej chwili pozwolą uniknąć takiej kompromitacji Polski na arenie międzynarodowej?

Rozszerzono ją, pod wpływem klubu Kukiz wprowadzono wątek ukraiński, który w ogóle nie został w tej chwili przeanalizowany i wymagałby również korekty. Otóż myślę, że nauczyliście się państwo, w jaki sposób można szybko, skutecznie negocjować, by zmienić złe ustawy. Wykorzystajcie to doświadczenie w waszych kontaktach z Komisją Europejską.

Panie Ministrze! Na wstępie dziękuję panu ministrowi za udzielenie odpowiedzi na dosłownie trzy pytania, a zwłaszcza na to ostatnie pytanie. Bardzo się cieszę, że rząd nie przewiduje zmian w ustawie penalizującej banderyzm. Odniosę się do słów pana ministra i zaapeluję, aby w tej drugiej części wypowiedzi odniósł się do tych zasadniczych kwestii, do tych informacji, które najbardziej bulwersują polską opinię publiczną.

Bardzo zręcznie pan minister atakuje Platformę Obywatelską - i słusznie - za to, że w czasach, kiedy Platforma rządziła, pan Jan Tomasz Gross, socjolog, atakował Polskę i poniewierał nią na arenie międzynarodowej. Natomiast państwo w tej chwili przekazaliście 750 tys. zł pani prof. Engelking-Boni, która też ma zasługi, powiedziałbym, bardzo duże w tej mierze, wspierając chociażby pana prof. Grabowskiego i jego kłamstwo na temat historii Polski. Jeśli chodzi o mój komentarz do kwestii związanych z art. 123, proszę się wnikliwie wczytać w kwestię dotyczącą ustaw regulujących ustrój i właściwość władzy publicznej.

I ostatnia rzecz w tej krótkiej wypowiedzi. Polacy nie są naiwni.

Pan poseł Robert Winnicki, niezrzeszony. Wysoka Izbo! Tak jak tu zostało powiedziane, pan minister raczy obrażać inteligencję Polaków takimi sformułowaniami, że negocjacje z Izraelem nie dotyczyły ekspresowego tempa, nadzwyczajnego, skandalicznego tempa, w jakim była procedowana ta nowelizacja w ubiegłym tygodniu: bez drugiego czytania, bez debaty, bez odsyłania do komisji, co najważniejsze, bez pytania się Polaków o zdanie, bez pytania się Polaków o zdanie w tej kwestii. Ponieważ baliście się reakcji, ponieważ naopowiadaliście w styczniu, w lutym tego roku tyle dyrdymałów na temat swojej niezłomności, że doskonale sobie zdawaliście sprawę, że teraz król jest nagi, że wy jesteście nadzy. Panie ministrze, ja jeszcze raz proszę, żeby pan odpowiedział na pytanie: Co w takim razie, zgodnie z informacjami, jakie są powszechnie dostępne w Izraelu, jak również w Polsce, było negocjowane w ośrodkach Mosadu w Izraelu, co było negocjowane w Wiedniu, bo takie są potwierdzone na ten temat informacje? Prosiłbym również o odpowiedź na pytanie: Jak mamy traktować to porozumienie, które państwo podpisali z Izraelem i którego tak szumnie nie ogłaszali?

Cała ta debata jest tak naprawdę potwierdzeniem mitologii, jaką tworzy Izrael, czyli, po pierwsze, że II wojna światowa to przede wszystkim prawie wyłącznie cierpienie Żydów, a po drugie, że wszystkie inne narody to narody współsprawców, bo Polacy występują tam głównie również jako współsprawcy. To nie jest żaden sukces.

Była specjalna strona internetowa w językach polskim, ukraińskim i angielskim poświęcona zbrodni wołyńskiej - tak się nazywała - prokuratorzy prowadzili śledztwa, kilkadziesiąt śledztw w sprawie zbrodni na Wołyniu, kwalifikując ją jako zbrodnię ludobójstwa, zebrano kilkaset relacji świadków tych zbrodni. A więc nie było potrzeby nowelizacji tej ustawy, natomiast tak to zrobiono, wymieniając tam siedmiokrotnie Ukraińców, że doprowadziło to do zadrażnienia i popsucia stosunków z Ukrainą. Przecież tam mamy kwestię ustalenia nazwisk wszystkich ofiar zbrodni wołyńskiej. jest kwestia przeprowadzenia tam właśnie ekshumacji, jest kwestia zapewnienia godnego pochówku tym ofiarom, jest kwestia upamiętnienia tych miejsc. Prezydent zakwestionował kilka zapisów dotyczących Ukrainy w tej ustawie i posłał je do Trybunału Konstytucyjnego, ale nawet jak trybunał uzna, że to jest zgodne z konstytucją, to może to Polsce bardzo szkodzić, [[Dzwonek]] chociaż z konstytucją się zgadza.

Wysoka Izbo! Na początek chcę odnieść się do słów pana ministra, który raczył powiedzieć, że poseł Rzymkowski w swojej wypowiedzi obraził Wysoką Izbę. Nic bardziej mylnego, panie ministrze. Otóż poseł Rzymkowski odnosił się do rządu, nie do całej Izby, ponieważ to wy odpowiadacie za ten cały bubel, to was historia oceni i to wy doprowadzacie do tego, że politykę wstawania z kolan zamieniacie na politykę padania na twarz przed innymi krajami. Szanowni Państwo! Zdaniem wielu polityków PiS, a także wspierających ich dziennikarzy styczniowa nowelizacja ustawy o IPN to walka o suwerenność.

Panie Ministrze! Wysoka Izbo!

Wnioskodawca zarzuca rządowi i oczywiście nam jako partii rządzącej, że nie zachowano czujności i nie przyjęto zgłaszanych uwag przez podmioty zewnętrzne.

Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Bardzo szanuję pana zaangażowanie w prace parlamentarne, a teraz również w prace rządowe, niemniej jednak chcę wyrazić z tego miejsca sprzeciw, ogromny sprzeciw. Myślę, że poprą to również inne ugrupowania opozycji.

Mam pytanie: Czym była spowodowana błyskawiczna akcja złagodzenia ustawy o IPN polegająca na wycofaniu się z zapisów karnych? Zgłaszaliśmy poprawki jako opozycja, że to nie będzie miało skutku i zastosowania poza granicami kraju.

Dziękuję bardzo. Panie Ministrze! Sytuacja jest po prostu. Panie ministrze, znamy się już parę lat i powiem szczerze, że pan doskonale wie, o czym my mówimy. Otóż mamy: Bóg, honor i ojczyzna. Na Boga nie macie wpływu, ojczyzna jest nasza, został wam tylko i wyłącznie honor. Pytam się, gdzie on jest, skoro pod wpływem obcego mocarstwa zmieniacie najważniejszy zapis ustawy IPN, który brzmiał w ten oto sposób: kto wbrew faktom zniesławia naród polski. Co takiego jest w tym zdaniu, że aż interwencja zachodnia musiała nastąpić, żeby wyciąć najważniejsze zdanie z całej ustawy?

Nie będę używał tu przymiotników, które należałoby wypowiedzieć w tej kwestii. Natomiast, proszę państwa, Kukiz’15 w tej sprawie zachował się, jak trzeba, w odróżnieniu od Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo. Pan poseł Jan Kilian, Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Styczniowa nowelizacja ustawy o IPN to pewnego rodzaju ważny krok w mówieniu prawdy, pewnego rodzaju nawet egzekwowaniu mówienia prawdy o historii Polski. Opozycja w każdym momencie swej bytności w Sejmie oprotestowuje absolutnie wszystko, każde posunięcie rządu, dzisiaj także, chociaż w tej sprawie akurat wtedy milczała. To oczywiste, że od lat potępiamy antysemityzm w każdej postaci, jest deklaracja podpisana przez przywódcę Izraela o tym, że oni potępiają antypolonizm, który zresztą odkryliśmy, zauważyliśmy, szczególnie intensywny, w ostatnich miesiącach.

To jest w tej deklaracji, że to było państwo, które nie kolaborowało, sprzeciwiało się Holokaustowi, walczyło do końca z Niemcami, utworzyło organizację pomocy Żydom w okupowanej przez Niemców Europie, ostrzegało cały świat przed Holokaustem i prosiło o pomoc.

Czy nie wydaje się, że i sam Izrael nie do końca przewidział tę sytuację? Dziękuję. Dziękuję. Wysoka Izbo! Z przykrością odnotowaliśmy fakt, informacje płynące z prasy izraelskiej o tym, że to służby Mosadu, służby obcego wywiadu podyktowały nam, Polsce, polskiemu parlamentowi, Senatowi, prezydentowi zapisy nowelizacji ustawy o IPN. Chciałem się zapytać, w zasadzie nie pana ministra, tylko premiera Morawieckiego, czy wszystkie ustawy uchwalane większością Prawa i Sprawiedliwości są dyktowane przez służby obcych wywiadów, czy tylko ta jedna. My w pełni jako Kukiz’15 rozumiemy, że jest dyplomacja, jesteśmy za świetnymi relacjami z Izraelem, z Tel Awiwem, z Waszyngtonem, z Brukselą, z Moskwą. Są narzędzia w dyplomacji międzynarodowej, z których można korzystać, ale żadne państwo, które chce być traktowane w sposób podmiotowy, nie pozwoliłoby na wykorzystanie narzędzia, jakim jest dyktowanie prawa przez służby obcego wywiadu. Państwo tym działaniem sprawili, że za państwa rządów Polska stała się państwem podmiotowym, i tak jest postrzegana na arenie międzynarodowej. Państwo sprawili, że Polska postrzegana jako - i być może tak jest - nie suwerenny kraj, tylko jako kondominium pod wiadomym zarządem powierniczym. Dziękuję. Pan poseł Andrzej Kryj, Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ja jednak nie pomniejszałbym znaczenia tej wspólnej deklaracji i starał się zwrócić uwagę na pewne fakty, które wcześniej naprawdę nie wybrzmiewały tak, jak wybrzmiały w tej deklaracji. Otóż w pkt 3 mowa jest o tym, że zawsze byliśmy zgodni, że sformułowania „polskie obozy koncentracyjne”, „polskie obozy śmierci” są rażąco błędne i pomniejszają odpowiedzialność Niemców za tworzenie tych obozów.

Dziś w tej deklaracji po raz pierwszy chyba tak mocno wybrzmiewa stwierdzenie, że to Niemcy odpowiadają za obozy śmierci.

Pamiętają państwo, kto był wnioskodawcą tej uchwały. Tam wnioskodawca napisał, że Polacy próbowali wyzwolić się z pruskiej niewoli. Mam pytanie. Panie ministrze, to jest początek drogi i chciałbym zapytać, jakie działania planuje prowadzić rząd oraz inne podmioty, np. Polska Fundacja Narodowa, aby do opinii publicznej świata przebijała się prawda o postawie polskiego narodu, Polskiego Państwa Podziemnego w czasach II wojny światowej [[Dzwonek]] i w jaki sposób będziemy zwalczać przejawy antypolonizmu, gdyż w deklaracji mówi się o tym, że oba rządy odrzucają antypolonizm, a jednak to przejawy antysemityzmu będą zwalczane. Dziękuję bardzo.

Witamy. Dziękuję, panie marszałku. Pierwsze to jest pytanie o ustawę styczniową, bo wiemy wszyscy, że była notatka MSZ-etu mówiąca o pewnych kontrowersjach, które ta ustawa budzi.

Czy poza wykupionymi artykułami pojawiały się jakiekolwiek inne wzmianki w mediach zagranicznych na temat wspólnej konferencji i przede wszystkim tej rzekomo propolskiej wypowiedzi Netanjahu i czy to w ogóle zostało zauważone, bo można co do tego mieć wątpliwości? I czy rzeczywiście to jest taki olbrzymi sukces, czy ten sukces jest tylko w głowach twórców tego całego zamieszania?

I jakie były przesłanki, żeby stosować to megaszybkie tempo teraz, ostatnio? Dziękuję bardzo. Pan poseł Krzysztof Głuchowski, Prawo i Sprawiedliwość. Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Czy w związku z rezygnacją z penalizowania kłamstwa wobec państwa i narodu polskiego w ustawie o IPN, która to penalizacja nakładała na prokuraturę obowiązek dowiedzenia, że do przestępstwa doszło, został lub zostanie opracowany dokument rządowy, który jednoznacznie określi przypadki wypowiedzi i zachowań, jakie będą przez instytucje państwowe zaskarżane do sądów w ramach powództwa cywilnego? Dziękuję bardzo. Pani poseł Agnieszka Ścigaj, Kukiz’15. Wysoka Izbo! Trybu też dotyczy moje pytanie.

Upłynęło 6 miesięcy i dopiero pan premier uderzył pięścią w stół i powiedział, że dość tego. Nie wiem. Sprawa związana z osobami niepełnosprawnymi.

Dziękuję bardzo. Pani poseł Anna Krupka, Prawo i Sprawiedliwość. Wysoka Izbo! W zeszłym tygodniu Sejm przyjął nowelizację uchwalonej w styczniu zmiany ustawy o IPN. Jaki cel przyświecał pierwotnej zmianie ustawy? Dlaczego zdecydowano się na jej nowelizację? Jaki jest cel tej czerwcowej nowelizacji? Czy ten cel został osiągnięty? Ponadto czy za rządów PO-PSL podjęto działania, które miały zapobiec szkalowaniu dobrego imienia Polski? Jeżeli tak, to jakie? Jakie działania podjęto za rządów Prawa i Sprawiedliwości - jakie działania już zostały podjęte - by bronić dobrego imienia Polski i narodu polskiego? Jakie działania rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego zamierza podjąć? Jakie kolejne kroki wynikające z tej nowelizacji rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego zamierza podjąć? Pan poseł Jerzy Jachnik, Klub Poselski Kukiz’15. Wysoka Izbo!

8 listopada jest sprawozdanie komisji.

Pierwsze. Czy premier, kiedy został premierem, znał notatkę Ministerstwa Spraw Zagranicznych o sytuacji? Czy marszałek Sejmu znał notatkę Ministerstwa Spraw Zagranicznych? To jest pierwsze pytanie. I drugie pytanie - do pana ministra i do całej sali: Czy państwo jako parlamentarzyści VIII kadencji Sejmu nie czujecie się upodleni sposobem procedowania tej ustawy? Bo ja tak. Dziękuję bardzo. Pan poseł Piotr Polak, Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Rządowi pana premiera Mateusza Morawieckiego, jak żadnemu wcześniej, zależało i zależy na obronie dobrego imienia Polski w wymiarze historycznych ocen II wojny światowej. Takie też były cele i tej pierwszej ustawy, i tej nowelizowanej. W związku z tym chciałbym zapytać pana ministra, czy to prawda, że na wspólnej konferencji, która odbyła się już po uchwaleniu i znowelizowaniu tej ustawy właśnie pod koniec czerwca, padły jednoznaczne deklaracje i stwierdzenia, że Polska została uznana za ofiarę II wojny światowej, że nie jest sprawcą Holokaustu. Chciałbym również zapytać, czy w tym samym czasie bądź bezpośrednio po tej konferencji Departament Stanu Stanów Zjednoczonych wydał podobnej treści oświadczenie, stanowisko, w którym też jednoznacznie stwierdza, że określenia obarczające, to jest cytat, państwo polskie odpowiedzialnością za zbrodnie nazistów niemieckich na terenie okupowanej Polski, takie jak polskie obozy śmierci, są nieprawdziwe i krzywdzące. Chciałbym również zapytać, czy został już powołany bądź zostanie w najbliższej przyszłości powołany specjalny polsko-izraelski zespół do spraw dialogu. Była o tym mowa. Była też o tym mowa właśnie na tej wspólnej konferencji. Dziękuję. Pan poseł Grzegorz Wojciechowski, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Zaniedbania są wieloletnie, a nawet powiedziałbym, wielodziesięcioletnie. Chodzi o to, że najpierw to były zbrodnie niemieckie, mieliśmy komisję do spraw badania zbrodni niemieckich.

Muszę powiedzieć, że nie spotkałem się z kimś, kto powiedziałby, że ci zbrodniarze mówili po faszystowsku czy też mówili po nazistowsku, oni mówili po niemiecku.

Chodzi mi o odbiór tego w Izraelu, odbiór opinii publicznej, w mediach. Chciałbym usłyszeć od pana ministra, jak cała sprawa związana z tą ustawą jest odbierana i jak jest odbierane wydanie później wspólnego oświadczenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie marszałku. Również panu dziękuję. Wysoka Izbo! To jest fakt. W takim razie mam pytanie: Co chcemy osiągnąć, tłumacząc się z faktu, że Polska była napadnięta przez Niemcy? To jest oczywista sprawa. Dziękuję bardzo.

Szanowni Goście na Galerii! Moje pytanie to: Czy przyjaźń polsko-izraelsko-amerykańska zostanie wpisana do Konstytucji RP, tak aby projekty ustaw, które mają ją umacniać, mogły być procedowane w trybie pilnym w ciągu kilku godzin, tak aby premier Netanjahu nie spóźnił się na obiad, a prezydent Trump na drugie śniadanie? I jeszcze jedno: Ile razy użył określenia „Niemcy” w swoim ostatnim wystąpieniu departament stanów? Proszę teraz o zabranie głosu przedstawiciela wnioskodawców pana posła Tomasza Rzymkowskiego. Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!

Przypomnę, że ustawę uchwaliliśmy ponad rok później, w styczniu 2018 r. Proszę państwa, czytam fragment. Wobec rozpowszechniania przez część środowisk żydowskich, jak również instytucji i organizacji zajmujących się upamiętnieniem Holokaustu, w tym Instytut Yad Vashem oraz Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie, skrajnie negatywnych opinii na temat projektu ww. ustawy - chodzi o ustawę o IPN - której rzekomym celem ma być: próba zastraszenia i zapobieganie wolnym badaniom naukowym i dyskusji nad przeszłością Polski, konieczne jest podejmowanie aktywnych działań służących prezentacji stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej, w tym zwłaszcza wyjaśnieniu przesłanek dotyczących konieczności wprowadzenia ustawowej penalizacji znieważenia narodu polskiego. O znaczeniu tego typu działań świadczy m.in. fakt osobistego odniesienia się do tematyki nowelizacji ustawy o IPN przez premiera Państwa Izrael pana Benjamina Netanjahu w rozmowie z panią premier Beatą Szydło podczas niedawnych polsko-izraelskich konsultacji międzyrządowych.

Stąd też ponownie zadaję to pytanie: Jak to jest możliwe - pytałem o to również wiceministra sprawiedliwości, który odpowiadał za ten projekt i pilotował ten projekt ustawy - że rząd polski był całkowicie zaskoczony, i dlaczego wybrano tę datę, w przededniu uroczystości w muzeum Auschwitz, na uchwalenie tej ustawy? Nie mieliśmy żadnych działań osłonowych. Nie było żadnych rozmów ze stroną izraelską. Strona izraelska była zaskoczona tą sytuacją. I po 5 miesiącach kapitulujemy, poddajemy się, za rękę jesteśmy prowadzeni przez funkcjonariuszy Mosadu, o czym dzisiaj świadczą przywołane przez nieobecnego tutaj pana posła Szczerbę informacje prasowe. To jest absolutny skandal. Pytanie do rządu jest następujące: Czy państwo planujecie przygotowanie jakiejś białej księgi, wyjaśnienia wszelkich okoliczności? Bo nosi to znamiona jakichś wewnętrznych walk frakcyjnych. To, co przywołał bardzo słusznie pan poseł Jachnik: w grudniu - 13 grudnia - jest powoływany rząd pana Mateusza Morawieckiego i nagle po 15 miesiącach trzymania w zamrażarce ustawy ustawa jest odpalona. Korelacja zdarzeń, brak konkretnych działań związanych z wytłumaczeniem stronie izraelskiej, o co apeluje konkretnie minister spraw zagranicznych, czy ta współpraca była. Ponawiam pytanie o to, kto w tych negocjacjach, o których wiemy, że były prowadzone, i to w Wiedniu i w Izraelu, reprezentował Polskę? Czy prawdą jest, że uczestniczyli w tych rozmowach funkcjonariusze obcych służb specjalnych? Ponawiam to pytanie po raz kolejny, panie ministrze. Chodzi konkretnie o dyskusję nad art. 55a.

Pytanie do rządu: Czy ta kwestia została wyjaśniona? Natomiast rzeczywistość brutalnie pokazała, że jest zupełnie inaczej. Jeśli chodzi o relacje z Ukrainą, pani poseł skierowała to pytanie też do mnie w kontekście tego fragmentu dotyczącego penalizacji banderyzmu. Proszę mi wierzyć, byłem niedawno na Ukrainie i byłem przyjmowany z wszelkimi honorami. Naprawdę Ukraina szanuje państwa, które same się szanują. Szanujmy siebie i szanujmy naszych sąsiadów, w partnerstwie budujmy dobre relacje.

Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu sekretarza stanu, szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pana Michała Dworczyka. Panie Marszałku! Panie pośle, jeszcze raz powtórzę, że nie były prowadzone żadne negocjacje na temat nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Może pan to powtórzyć jeszcze 10 razy, rozumiem, że temat jest chwytliwy medialnie, że chcecie państwo, bo to nie tylko pan takie sugestie wypowiadał z tej trybuny pod część elektoratu, sformułować przekaz, ale nawet jeśli dwudziestokrotnie to powtórzycie, to fakty są takie: nowelizacja ustawy o IPN nie była z nikim negocjowana. Po drugie, jestem trochę zaskoczony, może w mniejszym stopniu, jeśli chodzi o pana posła Szczerbę, ale w większym stopniu, jeśli chodzi o pana posła Rzymkowskiego, że jak prawdę objawioną traktujecie słowa izraelskich polityków, którzy wypowiadają się w sposób dla mnie niezrozumiały i zaskakujący. na temat spraw, o których dzisiaj rozmawiamy. Mogę tylko powtórzyć, mogę tylko powtórzyć: to nie jest prawda.

Naprawdę, my nie musimy brać. My kierujemy się przede wszystkim i wyłącznie, mam nadzieję, polską racją stanu, a to, że komuś się nie zawsze podoba prawo, które jest w Polsce stanowione, to już nie nasza. Mówi się trudno, po prostu. Dla nas jest sprawą nadrzędną polska racja stanu.

Któryś z panów posłów twierdził, że prezydent był ściągany z zagranicy, żeby podpisać ustawę. To bzdura.

Jestem trochę zaskoczony wypowiedzią pana posła Winnickiego.

Zakładam, że nie była to bezmyślność, zajęcie tego miejsca, tylko przemyślana akcja. Chodziło o szybkie dokończenie procedowania, więc dzisiaj wystąpienia pana posła Winnickiego są dla mnie naprawdę niezrozumiałe.

Jeśli chodzi o to, że narracja izraelska - o tym też chyba mówił pan poseł Winnicki - jest jakaś triumfalistyczna, że Polska na tej deklaracji podpisanej przez premiera Morawieckiego i Netanjahu miałaby coś stracić, przeczą temu fakty, i to fakty nie tylko w postaci treści tej deklaracji, ale też publikacji, które się pojawiają w Izraelu.

Nie wygląda to na teksty w duchu triumfalizmu w związku ze znowelizowaną ustawą o IPN. Do wypowiedzi pani poseł Radziszewskiej i pana posła Szczerby naprawdę chyba nie warto się odnosić, bo to wy, państwo, prowadziliście przez lata politykę takiej pedagogiki wstydu i, wielokrotnie przez wasze działania, politykę oczerniania Polski za granicą. Przykłady już w tej Izbie podawałem. Chyba poseł Masłowski zadał pytanie, czy będzie można bezkarnie używać określenia: polskie obozy śmierci.

Ale namawiam, jeżeli niemożliwe jest przeczytanie i zrozumienie, żeby pan spróbował użyć w Polsce publicznie takiego określenia i wtedy zobaczymy. Proszę?

Jeśli chodzi o to, że ta deklaracja jest niewiele warta, takie tu się pojawiły stwierdzenia, i właściwie nic nie mówi na temat sprawców II wojny światowej i sprawców Holokaustu, to ja, jeśli pan marszałek i Wysoka Izba pozwolą, przytoczę kilka cytatów z tej deklaracji podpisanej przez obu premierów: „Oczywistym jest, że Holokaust był bezprecedensową zbrodnią popełnioną przez nazistowskie Niemcy przeciwko narodowi żydowskiemu i wszystkim Polakom żydowskiego pochodzenia” Pierwszy cytat, który chyba nie pozostawia wiele wątpliwości. Kolejny cytat a propos narracji historycznej i rzekomo tego, że deklaracja jest nieistotna i nie ma żadnego znaczenia. Obaj premierzy mówią: „Zawsze byliśmy zgodni, że sformułowania 'polskie obozy koncentracyjne' czy 'polskie obozy śmierci' są rażąco błędne i pomniejszają odpowiedzialność Niemców za tworzenie tych obozów. Jeszcze ostatni cytat: „Nie zgadzamy się na działania polegające na przypisywaniu Polsce lub całemu narodowi polskiemu winy za okrucieństwa popełnione przez niemieckich nazistów i ich kolaborantów z różnych krajów i różnych narodowości. Bardzo dziękuję. Myślę, że to jest najlepsze podsumowanie tego, czym jest ta deklaracja, którą próbujecie państwo zdeprecjonować. Aha, jeszcze pan poseł Apel pytał, czy informacja była powielana w innych krajach przez media. Tak, była.

Absolutnie nie odstępujemy od walki o dobre imię Polski, tylko tak jak już pan premier mówił, powtórzę, polityka polega na skuteczności i pewna dojrzałość polityczna polega na tym, żeby skutecznie dobierać narzędzia, aby osiągać cele. Dzięki tej nowelizacji jesteśmy przekonani, że będziemy mogli skuteczniej walczyć o dobre imię Polski poza granicami kraju. Jeśli chodzi o same przepisy karne, na samo zakończenie zwracam się do pana posła Jakubiaka, to przypomnę, panie pośle, art. 133 Kodeksu karnego: kto znieważa naród polski lub Rzeczpospolitą Polską, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Panie Ministrze! Przede wszystkim chciałbym sprostować. Ja nigdy nie rozmawiałem z panią ambasador Azari. Rozmawiał podobno pan minister Jaki. Mówię „podobno”, bo nadal nie wiem, czy te rozmowy rzeczywiście były, czy ich nie było. Uważam za absolutnie zabronione, aby pod wpływem obcych ambasad pisać polskie prawo. Bardzo proszę ewentualnie o odpowiedź na piśmie na te pytania, które zadałem, a na które odpowiedzi nie otrzymałem. I jeszcze tak a propos prasy, bo pan tutaj powoływał się na prasę izraelską. Przed chwilą pan Barak Ravid poinformował, że stronę polską podobno, pytam, reprezentował pan prof. Ryszard Legutko i pan europoseł Tomasz Poręba. Dziękuję bardzo. Ja wspieram tutaj apel pana posła o to, żeby pan minister przedstawił na piśmie odpowiedzi na te pytania, na które pan minister nie odpowiedział. Ogłaszam 5 minut przerwy.

Wznawiam obrady. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 29. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (druki nr 2667 i 2713) Proszę pana posła Piotra Króla o przedstawienie sprawozdania komisji. Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji o rządowym projekcie ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, druki nr 2667 i 2713. Celem projektu ustawy jest wsparcie realizacji założeń „Narodowego programu mieszkaniowego”, który jest jednym z priorytetowych narzędzi realizacji „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” Jednym z komponentów „Narodowego programu mieszkaniowego” jest program „Mieszkanie+”, który zakłada wsparcie budownictwa na wynajem z możliwością dojścia do własności, budownictwa komunalnego i chronionego. Projekt ustawy wpisuje się w pakiet działań mających na celu wsparcie budownictwa mieszkaniowego dostępnego również dla osób o niskich i przeciętnych zarobkach. Podstawowym problemem polskiego mieszkalnictwa jest statystyczny niedobór mieszkań. Szacowany statystyczny deficyt mieszkaniowy na koniec 2015 r. wynosił w Polsce ok. 897 tys. Nie można zapominać również, że problemem polityki mieszkaniowej w Polsce jest także brak dostępnych mieszkań dla osób, których dochody są zbyt wysokie, aby ubiegać się o mieszkania gminne, i jednocześnie zbyt niskie, aby zaciągnąć kredyt na zakup własnego mieszkania. Szacuje się, że dziś w Polsce w podobnej sytuacji jest ok. 40% społeczeństwa, w tym głównie młode osoby rozpoczynające karierę zawodową.

W niektórych miejscowościach wzrosty są dwucyfrowe. Przykładowo średnia stawka za metr kwadratowy mieszkania w Warszawie w ciągu ostatniego roku wzrosła o prawie 10% i wynosi 7821 zł. Dwucyfrowe wzrosty zanotowano w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach i Szczecinie. Według raport NBP w samym I kwartale tego roku na rynku pierwotnym w Gdańsku ceny transakcyjne wzrosły o ponad 6%, a w Katowicach na rynku wtórnym - o ponad 7%. Projekt jest narzędziem umożliwiającym redukcję deficytu mieszkań i doprowadzenie do sytuacji, w której podstawowe parametry określające poziom zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych nie będą odstawały od przeciętnych wartości rozwiniętych krajów Unii Europejskiej. Projekt ustawy przewiduje przyjęcie rozwiązań deregulacyjnych polegających na upraszczaniu i usprawnianiu procedur administracyjnych związanych z realizacją inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Zaproponowane w projekcie rozwiązania deregulacyjne dotyczą głównie zasad lokalizowania inwestycji. O ustaleniu lokalizacji inwestycji będzie decydowała rada gminy, w drodze uchwały podjętej na wniosek inwestora. Wniosek inwestora o ustalenie lokalizacji inwestycji będzie podlegał upublicznieniu, z możliwością zgłaszania uwag przez zainteresowaną społeczność. Ocena planowanej inwestycji dokonywana będzie przez te same organy i podmioty, które dokonują tej oceny w toku zwykłego postępowania mającego na celu przyjęcie planu miejscowego, z tym że uzgodnienia zastąpiono opiniowaniem - z wyjątkiem wojewódzkiego konserwatora zabytków, zarządcy drogi oraz organu administracji geologicznej. Inwestycji mieszkaniowych lub inwestycji towarzyszących nie będzie można lokalizować na terenach podlegających ochronie przed lokalizowaniem lub zabudową na podstawie odrębnych przepisów, w tym także w otulinach form ochrony przyrody, rodzinnych ogrodach działkowych i obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, chyba że w trybie przepisów przewidujących tę ochronę inwestor uzyska zgodę na lokalizację inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszącej. Projekt ustawy zakłada także pozyskanie nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe, które do tej pory były niedostępne dla inwestycji mieszkaniowych, pomimo atrakcyjnej lokalizacji, wyposażenia w infrastrukturę techniczną oraz społeczną. Chodzi o grunty, które w przeszłości były wykorzystywane jako tereny kolejowe, wojskowe, produkcyjne lub usług pocztowych, a obecnie funkcje te nie są na tych terenach realizowane. Przygotowanie inwestycji mieszkaniowej będzie poprzedzone sporządzeniem koncepcji urbanistyczno-architektonicznej, zawierającej rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne inwestycji mieszkaniowej, z uwzględnieniem charakteru zabudowy miejscowości i okolicy. Koncepcję będą sporządzały osoby posiadające wiedzę specjalistyczną i doświadczenie w planowaniu przestrzennym, w tym urbaniści i architekci, którzy obecnie przygotowują projekty planów miejscowych oraz warunków zabudowy. Inwestycja mieszkaniowa będzie musiała spełniać wysokie standardy urbanistyczne, które ramowo zostały określone w ustawie. Standardy realizacji inwestycji zabezpieczają dostęp inwestycji mieszkaniowej do drogi publicznej, obsługę inwestycji niezbędną infrastrukturą techniczną, dostęp inwestycji do placówek powszechnej edukacji, takich jak szkoła czy przedszkole, dostęp do przystanku publicznego transportu zbiorowego, dostęp do urządzonych terenów wypoczynku oraz rekreacji i sportu. Samorząd gminny będzie miał prawo zwiększyć lub zmniejszyć wymagane od inwestora standardy, o 50% założonych w ustawie wskaźników, określając, w drodze uchwały, lokalne standardy urbanistyczne. Gmina będzie mogła dodatkowo określić również liczbę miejsc parkingowych niezbędnych do obsługi realizowanych inwestycji mieszkaniowej i towarzyszącej oraz obowiązek zapewnienia dostępu do sieci ciepłowniczej. Wybudowane budynki będą wymagać uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Dodatkowo wprowadza się wymóg dostosowania określonej liczby lokali mieszkalnych na potrzeby tych osób. Istotną kwestią jest także rozszerzenie formuły najmu instytucjonalnego o umowę najmu z docelowym przeniesieniem własności. W tym celu zaproponowano stosowne zmiany ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Proponowane rozwiązania maksymalnie redukują obciążenia administracyjnoprawne, co pozwoli na ograniczenie istotnych ryzyk inwestycyjnych. Oczekiwanym efektem będzie zatem przeprowadzenie tych inwestycji w sposób sprawny i efektywny. W ramach ustawy inwestycje mieszkaniowe będą mogły być realizowane znacznie szybciej, bowiem proces uzyskiwania zgody na lokalizację inwestycji będzie trwał do 60 dni, z możliwością wydłużenia o dodatkowe 30 dni. Z projektowanej ustawy będą mogły korzystać wszelkie podmioty realizujące inwestycje mieszkaniowe, o ile będą spełniać standardy urbanistyczne określone ustawą. Jednocześnie projekt ustawy nie wyłącza możliwości przygotowania lub realizacji całości lub części inwestycji na zasadach ogólnych, określonych w obowiązujących odrębnych przepisach. Ustawa będzie obowiązywać 10 lat. Projekt wpłynął do Sejmu 26 czerwca 2018 r., a w dniu 3 lipca 2018 r. został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji z zaleceniem zaopiniowania projektu przez Komisję Infrastruktury oraz Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. W dniu 4 lipca 2018 r. na posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji odbyło się pierwsze czytanie projektu. W posiedzeniu uczestniczyli również przedstawiciele Związku Miast Polskich, Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, posłowie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Podczas posiedzenia omówione zostały wszystkie propozycje przewidziane w projekcie. Przeprowadzono merytoryczną dyskusję nad rozwiązaniami zamieszczonymi w projekcie. Szczegółowo przedyskutowano przepisy umożliwiające realizację inwestycji niezależnie od istnienia lub ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, pod warunkiem że zamierzenie inwestycyjne będzie zgodne ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Rozmawiano również o kwestiach dotyczących ochrony przed zabudową terenów chronionych na podstawie bieżących przepisów - w szczególności chodzi tu o tereny rodzinnych ogródków działkowych - oraz o tzw. uwolnieniach nowych gruntów pod realizację inwestycji. Dyskutowano także o wachlarzu inwestycji towarzyszących, które będą możliwe do realizacji w trybie ustawy, i związanej z tym tematem kwestii renty planistycznej. Przeprowadzono rzeczową dyskusję o udziale społeczeństwa w procesie lokalizacji inwestycji. Dyskutowano także o zbyt krótkim w ocenie samorządów terminie, w którym gmina zobowiązana będzie wydać uchwałę o ustaleniu lokalizacji inwestycji. Poruszono także kwestie dotyczące standardów urbanistycznych, zarówno tych ustawowych, jak i lokalnych, które będzie ustalać gmina, oraz szczegółów dotyczących koncepcji urbanistyczno-architektonicznej. Środowisko architektów uczestniczyło w tej dyskusji. Związek Miast Polskich postulował zniesienie tzw. widełek 50%. W toku procedowania nad projektem przyjęto kilka poprawek o charakterze legislacyjnym i redakcyjnym, zgłoszonych przez Biuro Legislacyjne Sejmu. W trakcie posiedzenia został zgłoszony wniosek formalny o przeprowadzenie publicznego wysłuchania projektu ustawy. Wniosek nie zyskał poparcia komisji. W dniu 4 lipca 2018 r. odbyło się również wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Podczas posiedzenia połączone komisje pozytywnie zaopiniowały projekt ustawy. W imieniu Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji wnoszę o przyjęcie przedkładanego przez komisje projektu ustawy. Dziękuję panu posłowi.

Mam zaszczyt w imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości przedstawić Wysokiej Izbie opinię o rządowym projekcie ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Głównym celem tego projektu jest redukcja deficytu mieszkań i doprowadzenie do sytuacji, w której podstawowe parametry określające poziom zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych nie będą odstawały od przeciętnych wartości w rozwiniętych krajach Unii Europejskiej. Od lat polskie państwo, a właściwie polskie społeczeństwo, boryka się z ogromnym deficytem mieszkaniowym. Według szacunków na koniec 2015 r. statystyczny deficyt mieszkaniowy wynosił 867 tys., czyli tyle gospodarstw domowych potrzebuje swojego mieszkania dla godnej egzystencji. Oprócz ilościowych deficytów mieszkaniowych w kraju występują znaczące deficyty jakościowe mieszkań. Gospodarstwa domowe zajmują mieszkania o niskim stanie technicznym, niedostatecznie wyposażone w instalacje lub mieszkania przeludnione. Występują też deficyty jakości samych zespołów zabudowy: brak adekwatnej obsługi komunikacyjnej, w tym dostępu do transportu publicznego, brak dostępu do niezbędnych usług, w tym usług społecznych, do których zaliczyć należy również tereny rekreacyjne.

W związku z powyższym działania wymienione w projekcie koncentrują się na likwidacji deficytów ilościowych w segmencie mieszkań dostępnych cenowo oraz na rozwoju budownictwa na wynajem. Ta proponowana ustawa to realnie szybki krok na drodze do przeciwdziałania tym problemom mieszkaniowym, o których przed momentem mówiłam. Zakłada się, że potencjalnie głównymi mieszkańcami tworzonego nowego zasobu mieszkaniowego będą osoby z różnych grup wiekowych i pełne rodziny. Projekt określa zatem standard, jakiemu muszą odpowiadać inwestycje mieszkaniowe realizowane w zaproponowanym trybie, aby zapewnić dostosowanie tego zasobu do potrzeb użytkowników. Standardy te zabezpieczają dostęp inwestycji mieszkaniowej do drogi publicznej adekwatny do potrzeb obsługi komunikacyjnej oraz zapewniający miejsce do realizacji infrastruktury technicznej, obsługę inwestycji niezbędną infrastrukturą techniczną, zaspokojenie potrzeb bytowych mieszkańców w drodze zaspokojenia dostępu inwestycji do placówek powszechnej edukacji w odległości nie większej niż 3 tys. m, a w miastach, w których liczba mieszkańców przekracza 100 tys. mieszkańców, nie większej niż 1500 m, i dostępu do przystanku publicznego transportu zbiorowego w odległości nie większej niż 1000 m, a w miastach, w których liczba mieszkańców przekracza 100 tys. mieszkańców - 500 m. Samorząd będzie miał prawo zwiększać lub zmniejszać wymagane od inwestora standardy, ale tylko do 50% założonych wskaźników, określając, w drodze uchwały, lokalne standardy urbanistyczne. W lokalnych standardach urbanistycznych gmina będzie mogła określić również liczbę miejsc parkingowych niezbędnych do obsługi realizowanej inwestycji mieszkaniowej. Pragnę dodać, że ta ustawa jest wyczekiwana, dlatego że, tak jak już powiedziałam, brak mieszkania to brak zaspokojenia jednej z podstawowych potrzeb. Projektowane rozwiązania w związku z możliwością zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych przyczynią się do zwiększenia mobilności osób, w tym rodzin z dziećmi oraz osób niepełnosprawnych, w celu poszukiwania np. odpowiedniego zatrudnienia, co umożliwi zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dzięki zwiększonej dostępności mieszkań na własność. Pani poseł, proszę mi nie przeszkadzać. Proszę nie krzyczeć. To jest po prostu niegrzeczne z pani strony.

Proszę bardzo. Głos ma pani poseł Aldona Młyńczak, Platforma Obywatelska.

Wysoka Izbo! W imieniu Platformy Obywatelskiej przedstawiam opinię o rządowym projekcie ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, druki nr 2667 i 2713. Przedłożona specustawa mieszkaniowa została wprowadzona bocznymi drzwiami przez komisję deregulacyjną i była procedowana w nadzwyczajnym pośpiechu. Ustawa ważna, dotycząca polityki mieszkaniowej oraz planowania przestrzennego i zadań własnych samorządów, była procedowana poza komisjami merytorycznymi i o tym więcej powie wiceprzewodnicząca Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji pani poseł Małgorzata Janyska. Wracając do kwestii merytorycznych, należy stwierdzić, że projekt ustawy umożliwia lokalizowanie inwestycji mieszkaniowej na wniosek inwestora z pominięciem przepisów dotyczących planowania zagospodarowania przestrzennego, z ułomnymi konsultacjami społecznymi, a przede wszystkim z pogwałceniem polityki przestrzennej samorządów. Projekt ustawy wprowadza przepisy obciążające gminy działaniami deweloperów, a także będzie powodować rozlewanie się tkanki miejskiej, zamiast ją zacieśniać, powodując tym samym wzrost transportochłonności miast. Projekt ignoruje jakiekolwiek analizy dotyczące racjonalnego wskazywania terenów pod zabudowę mieszkaniową. Ustawa, szanowni państwo, nie respektuje istniejących planów. Ustawa stwarza warunki do bylejakości i do obniżenia standardów przy zagospodarowaniu przestrzeni. Skutki proponowanych deregulacji doprowadzą, naszym zdaniem, do dewastacji przestrzeni, która jest naszym cennym zasobem i którą należy gospodarować racjonalnie. Projekt ustawy został zaopiniowany negatywnie przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. Podzielając przekonanie o konieczności rozwiązania problemu dostępności mieszkań w naszym kraju, uważamy, że obecny projekt specustawy przyczyni się bardziej do dewastacji przestrzeni niż do pomocy obywatelom w zakresie polityki mieszkaniowej, bowiem ustawa w żaden sposób nie gwarantuje budowy mieszkań czynszowych, społecznych czy komercyjnych dla osób o średnich dochodach.

Nie takie były założenia projektu. Dlatego też, szanowni państwo, nie możemy poprzeć tej ustawy. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Platformy Obywatelskiej składam wniosek o odrzucenie projektu ustawy w całości. Składam również poprawki do projektu ustawy. Dziękuję. Chciałbym jeszcze powitać serdecznie grupę emerytów i rencistów z Doruchowa i Bukownicy, którzy przysłuchują się naszej debacie. Wysoka Izbo! Ten projekt to jest projekt, który można nazwać bardzo krótko: demolka+. Demolka+ z dwóch powodów. Ponieważ tą ustawą zostają zdemolowane podstawowe zasady ładu przestrzennego i teraz będzie można jak w filmach Barei postawić tutaj blok, mimo że jest jezioro, bo jezioro się przeniesie, proszę państwa.

Ta opinia powinna być podczas rozpatrywania tego projektu po pierwszym czytaniu w komisji. A tymczasem, proszę państwa, 3 lipca dowiedzieliśmy się, że następnego dnia będziemy ten projekt analizować w komisji deregulacyjnej. Głosowaliśmy w tym dniu, 3 lipca, do północy. Następnego dnia dostaliśmy specustawę, czyli coś specjalnego, nadzwyczajnego, wielkiego, epokowego, jak opowiadacie, i nie było w ogóle czasu na to, żeby się z nią zapoznać, żeby się do tego przygotować. Zresztą to było widać, bo posłowie z komisji deregulacyjnej, również poseł sprawozdawca i pani posłanka, która wypowiadała się w imieniu klubu. Nie odezwaliście się państwo ani razu, w żadnej kwestii, przy tej epokowej, wielce ważnej ustawie. Proszę państwa, dopiero o godz. 16 odbyły się posiedzenia połączonych komisji: infrastruktury i samorządu, które wydały opinię, która już nikomu nie była potrzebna, bo to już było na takim etapie procesu legislacyjnego, że komisja deregulacyjna już tego nie rozpatrzyła i nie rozpatrzy, proszę państwa. Zostało złamane zalecenie marszałka. Zdemolowaliście zalecenie waszego marszałka. Ale on pewnie wam nic nie zrobi, bo ta ustawa po prostu ma być politycznie przepchnięta, gdyż chcecie ogłosić sukces, powiedzieć: proszę bardzo - jak w serialu „Alternatywy 4”, [[Dzwonek]] proszę państwa, czy w innym filmie Barei - tu się zrobi to, co my zamierzamy. A kiedy, z jakimi skutkami - tego nawet nie chcecie wiedzieć. Dziękuję bardzo. Pan poseł Mirosław Suchoń, Nowoczesna.

Bardzo dziękuję. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam przyjemność przedstawić stanowisko Klubu Poselskiego Nowoczesna w sprawie rządowego projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Szanowni Państwo! O czym jest ta ustawa? Zgodnie z uzasadnieniem - tak jest napisane, trudno w to uwierzyć - ta ustawa jest krokiem w kierunku ograniczania barier administracyjno-prawnych w zakresie budowy mieszkań, spowoduje redukcję deficytu mieszkań. Natomiast założeniem projektowanej ustawy jest wprowadzenie regulacji umożliwiających znaczne przyspieszenie przygotowania i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Zgodnie z tym, co czytamy dalej w uzasadnieniu, projekt zakłada również wprowadzenie szczególnych zasad lokalizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Wysoka Izbo!

W dokumencie czytamy, tu cytuję: W ogólnym brzmieniu projekt ustawy stwarza wrażenie przedkładania interesu prywatnego inwestora ponad interes publiczny, a nawet podporządkowania tego drugiego dla większych zysków inwestora.

No chyba to oznacza, że Prawo i Sprawiedliwość chce coś ukryć. Na pewno w takiej sytuacji należy mieć wzmożoną czujność. Te odpowiedzi, tak jak powiedziałem, znajdujemy już na etapie konsultacji. Przytoczę: Projekt ustawy przedstawiony przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zawiera szereg zapisów, które nieodwracalnie odbiją się w negatywny sposób na ładzie przestrzennym polskich miast. Wprowadzenie ustawy w obecnym kształcie skutkować będzie zmniejszeniem roli planowania przestrzennego, ograniczeniem roli mieszkańców w kształtowaniu przestrzeni miast i podporządkowaniem procesów planistycznych woli politycznej, a co za tym idzie - zwiększeniem ryzyka, uwaga, zachowań korupcyjnych.

Panie ministrze, wstyd. Oczywiście nie jest tak, że ta ustawa zawiera same złe zapisy. Są tam zapisy pozytywne, które gdyby stanowiły element całości zmian systemu, choćby w zakresie parametrów technicznych inwestycji, uwzględniających dostęp do usług edukacyjnych, społecznych i rekreacyjnych. To są oczywiście dobre propozycje. Panie ministrze, gdyby to było elementem zmian całości systemu, a nie wyłomem, który zburzy ład polskich miast, to byłyby to dobre propozycje. Tymczasem jako całość ta ustawa stoi w sprzeczności z takim znanym, myślę, postulatem, z którym wszyscy powinniśmy się zgadzać, otóż z potrzebą uznania przestrzeni publicznej za dobro publiczne, a nie za własność jakiegoś bliżej nieokreślonego dewelopera, który może robić z tą przestrzenią, co mu się żywnie podoba. Zresztą, nawiasem mówiąc, kilka tygodni temu przyjmowaliśmy przepisy, które uniemożliwiają obchodzenie przez deweloperów zapisów planów zagospodarowania. I teraz przedstawiacie ustawę, która robi w tym wyłom, która zniszczy przestrzeń publiczną. Oczywiście to, co mówię, znajduje również potwierdzenie w opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego - co prawda o poprzedniej wersji ustawy, teraz po zmianach w komisji jest nowa, ale jednak - która wydała opinię negatywną. Natomiast trzeba powiedzieć wyraźnie, że te zmiany, które wprowadziliście, nie zmieniły ducha tej ustawy, nie zmieniły materii tej ustawy. Tak nie może być.

Bardzo proszę, pan poseł Paweł Szramka, Kukiz’15. Zgodnie z opinią projektodawcy ustawa pozwoli na uruchomienie gruntów, które do tej pory nie były brane pod uwagę przy budownictwie mieszkaniowym. Chodzi np. o grunty rolne w granicach administracyjnych miast, a także o obszary, które w przeszłości były wykorzystywane jako tereny kolejowe, wojskowe czy produkcyjne. Natomiast zdaniem przedstawicieli strony samorządowej projekt wcale nie gwarantuje, że nowe inwestycje będą powstawały na tych właśnie terenach. Co więcej, możliwość ignorowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego może spotęgować chaos przestrzenny, który i tak jest już dużą bolączką samorządową. Rada będzie mogła podjąć uchwały o ustaleniu lub o odmówieniu ustalenia lokalizacji, ale będzie musiała wziąć pod uwagę stan zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych gminy. To rodzi poważne obawy o ubezwłasnowolnienie rady gminy, która nie będzie mogła odmówić ustalenia lokalizacji bez podania odpowiedniego uzasadnienia, szczególnie w przypadku braku zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Dziękuję bardzo. Pan poseł Kazimierz Kotowski, Polskie Stronnictwo Ludowe - Unia Europejskich Demokratów. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Tak się składa, że w ostatnim okresie już po raz kolejny pochylamy się nad projektem rządowym, który dotyczy szeroko rozumianej gospodarki mieszkaniowej, zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych i - jak czytamy w uzasadnieniu tego projektu - podejścia do rozwiązania tego problemu i zabezpieczenia mieszkań, bo potrzeby są olbrzymie, sięgające ponad 800 tys. mieszkań. To wszystko to działanie w dobrym kierunku, tylko, panie ministrze.

A więc takie pytanie i refleksja nasuwa mi się również jako długoletniemu samorządowcowi: Czy musi być tak, że w tym jednym projekcie, w którym są słuszne cele, słuszne założenia i - uważam - dobre spojrzenie na ułatwienie procesu przygotowania inwestycji.

Czemu to ma służyć? Po pierwsze, panie ministrze, widzę, że jest pan z nami na posiedzeniach, stara się pan, tłumaczy pan nam, tylko proszę mi powiedzieć, po co taki zamęt i nieporozumienia już w czasie trwania procesu legislacyjnego. Komu wczoraj była potrzebna ta wydawana na siłę opinia Komisji Infrastruktury po zakończeniu posiedzenia komisji deregulacyjnej? Można zastanawiać się, można protestować, ale można nic nie mówić. Tylko jakie człowiek sam ma odczucia? Że pracuje w mechanizmie, który służy czemu? Czy projekt, panie ministrze, określa i wskazuje miejsca czy przestrzeń, w której będą budowane te obiekty? Tam jest tyle wątpliwości, że można przypuszczać, że mogą się w to wpisać inwestorzy, którzy mają inne plany, inne cele, a jak się zbuduje, to zgodnie z naszą tradycją. Przecież obiektu się nie przeniesie, musi służyć. Mam takie odczucie, że te samorządy już nie będą potrzebne czy nie będą miały wiele do powiedzenia, bo jest zapis o wpływie społeczności lokalnej na decyzję.

Kolejny temat: standardy urbanistyczne. Dobrze, ale nie ma też zapisów ani nie wskazuje się nigdzie, jakie są te minimalne. Skoro bowiem mówimy, że gmina może obniżyć standardy, to do jakiego poziomu? Przecież chcemy tworzyć akty prawne, które będą zapewniać wszystkim w naszym kraju podobne warunki życia, przynajmniej na tym podstawowym poziomie.

Przechodzimy do pytań. Jeśli ktoś z państwa chce się zapisać do głosu, to zapraszam. Głos ma pani poseł Małgorzata Pępek, Platforma Obywatelska. Wysoka Izbo! To inna ustawa niż przedstawiana kilka miesięcy temu, zupełnie inne założenia. Po konsultacjach resort zdecydował się na znaczną modyfikację swojego pierwotnego projektu. Zgodnie ze specustawą mieszkaniową w obecnym kształcie inwestycję mieszkaniową można byłoby realizować niezależnie od istnienia lub ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jednak nie mogłaby być ona sprzeczna ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jednostki samorządu terytorialnego. Czy to na pewno wystarczy, żeby zapobiec i tak już istniejącemu chaosowi urbanistycznemu w polskich miastach i na ich obrzeżach? Czy państwo nie widzicie, jak to wszystko w skali kraju wygląda? Czy nie okaże się, że grunty rolne w otoczeniu miast zostaną zabudowane blokami deweloperskimi? Dziękuję bardzo. Pani poseł Maria Małgorzata Janyska, Platforma Obywatelska. Mam pytanie do posła sprawozdawcy. Posłowie PiS-u i całej Zjednoczonej Prawicy, czy zdajecie sobie państwo sprawę z tego, że uczestniczycie w manipulacji prawnej, która doprowadza do tego, że będzie przyjęta ustawa z pogwałceniem regulaminu Sejmu? Czyli za ileś lat, jak będzie przywrócona praworządność w Polsce, to będziecie imiennie odpowiadać za negatywne skutki zapisów tej ustawy. Proszę państwa, Polacy przypomną sobie o tym, przypomną. Mimo że prosiliśmy was na posiedzeniach komisji, i komisji deregulacyjnej, i Komisji Infrastruktury połączonej z komisją samorządu terytorialnego, mówiliśmy o negatywnych skutkach, prosiliśmy pana przewodniczącego, który teraz siedzi tam z tyłu, żeby odroczył posiedzenie, skończył na pierwszym czytaniu i poczekał do rozpatrywania całej ustawy na opinie dwóch połączonych komisji, bo to jest obowiązek, niestety nie skorzystaliście z tego, czyli świadomie łamiecie prawo. Świadomie demolujecie tę praworządność. Po co? Co tam jest ukryte, proszę państwa? Czy naprawdę. Pan przewodniczący mówi, że czas?

Proszę, pani poseł Krystyna Sibińska, Platforma Obywatelska. Wysoka Izbo! Szanowna pani poseł, jak się nie zna tematu, to czasami lepiej w ogóle się nie odezwać niż mówić kłamstwa albo głupoty, bo tak inaczej. Nie ma w Polsce deficytu powierzchni pod budowę mieszkaniową. Odwrotnie. Jest bardzo dużo powierzchni pod budowę mieszkaniową zabezpieczonej w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Natomiast ustawa, którą wprowadzacie, specustawa. Trudno nazwać celem publicznym. Od tego zacznijmy. Pozwoli to zbudować wszystko i wszędzie, czyli deweloperzy będą mogli po prostu budować gdziekolwiek. i wcale niekoniecznie mieszkania, dlatego że szeroki katalog inwestycji towarzyszących spowoduje, że deweloper sobie wymyśli, że zbuduje obiekty handlowe, wybuduje jakieś obiekty usługowe czy inne obiekty, z których będzie czerpał korzyści, postawi jeden domek jednorodzinny i wyczerpie inwestycję mieszkaniową. Tak się nie robi.

Dziękuję. Pani poseł Aldona Młyńczak, Platforma Obywatelska. Panie Ministrze! Proszę mi wskazać przepisy, które jasno definiują, iż ten projekt ustawy będzie przeznaczony, będzie spełniał wymogi, które państwo określili w uzasadnieniu, czyli będzie realizował inwestycje mieszkaniowe w formie budownictwa czynszowego, komunalnego i społecznego, a nie będzie możliwości prawnej, tak jak już tutaj wcześniej było to przedstawiane, właśnie dla budowania wszystkich innych mieszkań, tudzież apartamentów, i sprzedaży ich po wysokich cenach, a więc zupełnie niezgodnie z projektem. Proszę mi także powiedzieć, dlaczego projekt nie przewiduje żadnych analiz ekonomicznych ani nie wymaga się prognozy skutków finansowych inwestycji do uchwały o lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub też inwestycji towarzyszących. Przecież to jest absolutnie konieczne. Analizy ekonomiczne i sporządzone prognozy mogą zapobiec właśnie takim inwestycjom nietrafionym, mogą skorygować zapędy niektórych inwestorów czy też gmin, czy też różnych osób prywatnych do budowania tam, gdzie takiej inwestycji nie potrzeba. A więc bardzo proszę o to, aby racjonalnie gospodarować przestrzenią. Tak samo proszę, aby przeprowadzać analizy ekonomiczne przed podjęciem uchwały lokalizacyjnej dla inwestycji [[Dzwonek]] i aby było to zapisane w ustawie, którą należy poprawić, tzn. odrzucić, ale jeśli przejdzie ona do dalszego procedowania, na pewno należy ją poprawiać. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo!

Chcemy, żeby powstawało więcej mieszkań, ale w sposób racjonalny.

Efektem tej ustawy będą osiedla na terenach rolnych, daleko od wszelkiej infrastruktury drogowej i społecznej, przede wszystkim wbrew zapisom miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Dziękuję. Chciałbym serdecznie powitać panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Zarzecza, które przysłuchują się naszej debacie. Proszę, pani poseł Zofia Czernow, Platforma Obywatelska. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Ład przestrzenny jest wartością, którą należy chronić. Ten projekt ustawy, który nie będzie honorował planów zagospodarowania przestrzennego, a więc prawa miejscowego, może spowodować nieodwracalne negatywne skutki dla przestrzeni miast, krajobrazu. Można rozwiązywać sprawy mieszkaniowe bez brutalnej ingerencji w pielęgnowaną od lat przestrzeń. Jestem zaskoczona, że sprawozdawca, wieloletni prezydent Świdnicy, z taką premedytacją popiera te rozwiązania, wiedząc, że one szkodzą miastom. Proszę pana posła i byłego prezydenta o refleksję. To jest po prostu niemożliwe. Mam pytanie. Jakie będą działania deweloperów na obszarach Natura 2000, których na Dolnym Śląsku jest bardzo dużo? Jakie będą działania inwestorów w strefach ścisłej ochrony uzdrowiskowej, a także na obszarach zagrożonych powodzią?

Pan poseł Marek Sowa, Nowoczesna. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Muszę powiedzieć, że jestem zdumiony, że może znaleźć się taki zapis, że inwestycje mieszkaniowe lub inwestycje towarzyszące realizuje się niezależnie od istnienia lub ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Panie ministrze, nie mogę pojąć, jak człowiek, który trafił do Sejmu z samorządu terytorialnego, może tak bezpardonowo niszczyć dorobek samorządu? Czy pan nie ma pojęcia, jak wyglądają osiedla, które zostały zrealizowane bez planów zagospodarowania przestrzennego w latach 90., na początku lat dwutysięcznych? One są dla nas dzisiaj powodem do wstydu, że nie potrafiliśmy racjonalnie zaplanować zagospodarowania krajobrazu. I pan dzisiejszą ustawą znosi ogromny dorobek wielu kadencji samorządowców, którzy w ostatnim czasie z ogromnym wysiłkiem przyjmowali plany zagospodarowania przestrzennego? Ja wiem, że to są bardzo trudne procesy, ale zobaczcie, jak się poprawiła jakość tej infrastruktury mieszkaniowej. Przecież w tych planach określa się wszystko: wysokość budynków, gęstość zabudowy, infrastrukturę publiczną. To wszystko tam się znajduje. Wy to wszystko jednym ruchem tniecie i firmujecie.

Pan poseł Krzysztof Truskolaski, Nowoczesna. Bardzo proszę. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Planowane zmiany w ustawie deweloperskiej wzbudzają ogromne emocje społeczne. Robicie wszystko, żeby jeszcze przed przerwą wakacyjną Sejm to uchwalił, Senat uchwalił i prezydent podpisał, a wy przed wyborami samorządowymi będziecie mogli się pochwalić tym, że budujecie mieszkania.

Teraz będziecie mówić: wybudujemy wszystko, wszędzie, tylko żeby przed wyborami samorządowymi można było to obiecać.

Czy chcecie, aby teraz spółki Skarbu Państwa były deweloperami, żeby PKP budowało mieszkania?

Dziękuję. Pan poseł Cezary Grabarczyk, Platforma Obywatelska. Wysoka Izbo! Panie Ministrze!

Mam pytanie do pana posła Piotra Króla, sprawozdawcy komisji deregulacyjnej. Jakie argumenty padły podczas posiedzenia komisji za odrzuceniem wniosku o wysłuchanie publiczne? Bo procedujemy nad tą ustawą w trybie superpilnym, tak jakby rząd nadał gryf pilności temu projektowi, i nie można przeprowadzić pełnej debaty, nie można spopularyzować jej rozwiązań. Ale także twórcy tej ustawy, tego gniota nie mogą wysłuchać krytycznych ocen. I jeszcze jedno pytanie do posła sprawozdawcy: Czy komisja deregulacyjna uwzględniła opinie? Czy miała okazję zapoznać się przed przygotowaniem sprawozdania na dzisiejsze posiedzenie z opinią, którą miały wspólnie wypracować Komisja Infrastruktury [[Dzwonek]] i komisja samorządu terytorialnego? Dziękuję. Pan poseł Ryszard Wilczyński, Platforma Obywatelska. Wysoka Izbo! Najlepszą miarą zrównoważonego rozwoju jest ład przestrzenny. Jedną z najważniejszych funkcji samorządu jest korzystanie z prawa decydowania o zagospodarowaniu przestrzennym, a decyzje w tym zakresie przesądzają o jakości życia mieszkańców na całe pokolenia. Państwo proponujecie zapis o lokalizowaniu tkanki mieszkaniowej poza ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego bądź sprzecznie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Tego typu zapisy mogą się pojawić niestety tylko w umysłach szaleńców. Mówię to z pełną odpowiedzialnością. Przy tej procedurze, kiedy nie można zważyć wszystkich okoliczności i samorząd będzie działał pod presją dużych inwestorów, co trzeba wiedzieć, każdy konflikt przestrzenny, a będzie ich masa, będzie owocował w przyszłości konfliktem społecznym. Zawsze tak jest. I będziecie za to na trwałe odpowiedzialni.

Pan poseł Mirosław Suchoń, Nowoczesna. Bardzo dziękuję. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Są z nami panie z koła gospodyń wiejskich i tak przypomniało mi się, że u mnie jest taki teren rekreacyjny, gdzie koło gospodyń wiejskich, kilka kół - bo to jest taka fajna impreza - ochotnicza straż pożarna organizują imprezy. jeżeli znajdzie się cwany deweloper i pozyska radnych z jednej, drugiej czy trzeciej gminy, to takich imprez już nie będzie. Nie będzie ich, bo on tam postawi 5-piętrowy budynek. Cztery piętra to będą mieszkania, a na dole będzie piękna powierzchnia handlowa. Taka jest ta ustawa, panie ministrze. Natomiast mam takie pytanie: Czy państwo w ogóle zastanowili się nad kosztami, które samorządy poniosą ze względu na to prognozowane rozlewanie się miasta na podstawie tej ustawy? Czy państwo zastanawialiście się, ile więcej samorządy wydadzą na wszelkiego rodzaju infrastrukturę, która jest konieczna do życia mieszkańców - na drogi, na wodociągi, na inne instalacje, bez których mieszkańcy żyć nie mogą? Jakie to będą koszty, jaka to będzie skala wzrostu? Czy znalazł się choć jeden samorząd, choć jedna malutka gmina, które poparły tę ustawę? Czy znalazła się choć jedna korporacja samorządowa choćby z jednego województwa, która [[Dzwonek]] poparła tę ustawę? Wydaje mi się, że nie. Ale jeżeli pan minister dysponuje choć jednym listem poparcia, to ja bym prosił, żeby pan minister był uprzejmy to zaprezentować i powiedzieć, który samorząd poparł tę ustawę. zapisanych do głosu została wyczerpana. Bardzo proszę o zabranie głosu sekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju pana Artura Sobonia.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Jeśli mówimy o przesuwaniu jeziora, to. był to film „Poszukiwany, poszukiwana”, a nie „Alternatywy 4” Nawet zabawnych filmów trzeba zapamiętywać tytuły, jeśli chce się je potem. przytaczać w debacie. Pan poseł Wilczyński pytał mnie o umysły szaleńców.

przestrzennego. Czy wśród tych szaleńców jest prezydent Lublina, który takich decyzji wydał jednego roku 142? Czy wśród tych szaleńców jest prezydent Poznania, który jednego roku wydał takich decyzji 295? A może prezydent Gdańska, który ich wydał blisko 100, albo prezydent Krakowa, który ich wydał blisko 500? Żyjemy w rzeczywistości, która jest. Panie ministrze, przepraszam. Szanowni państwo, bardzo proszę nie utrudniać wystąpienia ministrowi. Czy nie rozumieją panie po polsku? Bardzo proszę kontynuować, panie ministrze.

Jest ponad 83 tys. decyzji o warunkach zabudowy, które zmieniają polskie miasta w chaos przestrzenny, które doprowadzają do rozlewania się tych miast, prowadzą do kosztów społecznych, prowadzą dokładnie do tego, o czym państwo mówili. Żyjemy w rzeczywistości, którą trzeba poprawić, natomiast państwo przedstawiają tę rzeczywistość jako rzeczywistość idealną. Wystarczy pojeździć po Polsce, by zobaczyć, jak wygląda dzisiaj ta rzeczywistość. Poseł Suchoń w swoim wystąpieniu klubowym powiedział o odstąpieniu od standardów. Szanowni państwo, chcę państwu powiedzieć, o co chodzi z tym odstąpieniem od standardów. Chodzi o umowę z gminą na dowóz dzieci do szkoły w sytuacji, w której gmina wyrazi zgodę na to, aby inwestor podpisał taką umowę na dowóz dzieci do szkoły. Odstąpić od standardów, czyli konkretnie od tego, w tej ustawie można wyłącznie dlatego, że w ustawie zapisane zostały standardy. Dotychczas nikt w Polsce nie wymagał niczego od inwestorów, a my wprost w ustawie zapisujemy standardy, które będą od inwestorów wymagane. To jest zawsze za zgodą samorządu, zawsze za zgodą tzw. wysokich standardów, które zapisaliśmy bardzo precyzyjnie. Nie ma od nich odstępstwa, bo one są uwarunkowane. Chodzi wyłącznie o dowóz dzieci do szkoły, innych nie ma. Dlaczego? Dlatego że one są uwarunkowane pozwoleniem na użytkowanie. Odpowiadam na pytanie, czy wystarczy zgodność ze studium. Zgodność ze studium jest wpisana, dlatego że studia pokrywają całość przestrzeni polskich miast, tzn. wszystkie miasta mają studium. Jeśli mówimy o planowaniu przestrzennym, to plany zagospodarowania przestrzennego, aktualne plany zagospodarowania przestrzennego to jest 16% polskich miast. Mamy przyrost planów zagospodarowania przestrzennego o 1% rocznie. Czy to jest satysfakcjonujące? Czy jest satysfakcjonujące, że statystycznie takie planowanie trwa minimum 3 lata i że co trzeci plan nie obejmuje nawet 1 ha obszaru? To nie jest żadne planowanie przestrzenne, tylko załatwianie pojedynczych spraw. Czy grunty rolne spowodują dewastację przestrzeni? Szanowni państwo, mamy w polskich miastach 900 tys. ha gruntów rolnych. My w tej ustawie dajemy szansę na lokalizację inwestycji mieszkaniowych na terenach rolnych, które są bardzo często dobrze skomunikowane, z dostępem do szkoły w bezpośredniej bliskości osiedla, z dobrym dojazdem, za zgodą samorządów w bardzo uproszczonym trybie. Pracowaliśmy nad tym projektem 4 miesiące. To są uwagi, które uwzględniliśmy w tym projekcie, bo ten projekt, jak słusznie zostało też w tej debacie podkreślone, zmieniał się w wyniku tych uwag, które do nas wpływały. Ci wszyscy, którzy chcieli poprawiać ten projekt, także samorządowcy, poprawiali go wspólnie z nami, tak aby był kompromisem pomiędzy oczekiwaniami, które wiążą się z przestrzenią publiczną, a oczekiwaniem społecznym, którym jest szybsza i tańsza budowa mieszkań.

Pani poseł Sibińska niesłusznie atakowała panią poseł Kwiecień, która przytaczała rzeczywiste dane GUS. Jeśli pani poseł uważa, że gruntów w Polsce pod planami jest tak wiele, to dlaczego ceny tych gruntów są tak wysokie? Tylko uruchomienie dzisiaj większej podaży gruntów może wpłynąć pozytywnie na ten rynek. Mamy dzisiaj sytuację, w której deweloperzy mają banki ziemi. To oni decydują o podaży, oni decydują o marży, oni decydują o tym, za ile Polacy kupują mieszkania, a Polacy przepłacają za mieszkania. Z tym musimy skończyć.

My to zapisaliśmy z proporcjami i odległościami w sposób niezwykle precyzyjny. Czy jeden domek wystarczy, żeby taka inwestycja powstała? Nie, wystarczy przeczytać tę ustawę. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości.

To gmina decyduje o zagospodarowaniu terenu.

Zawsze gmina jest gospodarzem tego terenu. To gmina może i powinna zawierać takie porozumienia z inwestorami, które będą korzystne dla wspólnoty mieszkańców, których dotyczy realizacja tej inwestycji. Do czego jest nam to potrzebne - pytała pani poseł Młyńczak.

Tam muszą być inne funkcje, powinny być inne funkcje, aby ten teren był funkcjonalny, spójny, wygodny do życia. To nie może być wyłącznie budowanie samych bloków. Ta ustawa daje możliwość budowy tak dużych projektów inwestycyjnych w ramach programu „Mieszkanie+”, jakich w Polsce do tej pory się nie budowało. Czy powinny być policzone koszty, skutki ekonomiczne tej czy innej inwestycji realizowanej w ramach tego trybu? Szanowni państwo, my poprzeczkę podnosimy dużo wyżej, niż to jest dzisiaj. Dzisiaj, jeśli inwestor idzie po decyzję dotyczącą warunków zabudowy, nie musi nic. Natomiast my każemy mu przynieść koncepcję urbanistyczno-architektoniczną, która będzie kompletem informacji dla rady gminy, podstawą do podjęcia tej decyzji, co więcej, będzie miała również wszystkie opinie i zgody, będzie przygotowana przez profesjonalistów, będzie czymś, co pozwoli na racjonalne decyzje rady gminy, i ranga tej koncepcji w tej ustawie jest bardzo wysoka.

Tam, gdzie jest plan zagospodarowania przestrzennego, nie ma problemu, nikt nie będzie korzystał z tego trybu, bo dzisiaj będzie szybciej iść zgodnie z planem. Np. program „Mieszkanie+” w Katowicach nie jest realizowany już, tylko rok później, bo rok zajęła zmiana planu, zresztą z mieszkaniówki na mieszkaniówkę, mamy więc do czynienia z sytuacją, w której za zgodą samorządu upraszczamy procedurę, ale w żaden sposób nie ingerujemy w kompetencje samorządu. Udział społeczeństwa jest zapewniony na każdym etapie tego procesu: i na etapie lokalizacji, i na etapie pozwolenia na budowę. Jeśli chodzi o pytanie pana posła Sowy, jakie inwestycje będą mogły być realizowane na obszarach chronionych, to odpowiem: żadne. To przepraszam, w takim razie źle zanotowałem, ale było pytanie o to, jakie inwestycje mogą być na obszarach chronionych - żadne. Tzn. my w tym projekcie chronimy każdy obszar chroniony nawet dużo bardziej, niż to jest dzisiaj.

W projekcie tej ustawy nie ma uwzględnionych żadnych intencji, aby budować gdziekolwiek, chodzi o odblokowanie tańszych terenów, jeszcze raz powiem, po to, aby zwiększyć podaż tych terenów, skrócić procedury. Szybciej oznacza taniej, więcej mieszkań dostępnych cenowo oznacza lepszą ofertę dla Polaków.

Każdego dnia w Polsce powstają osiedla bez planów zagospodarowania przestrzennego, dlatego też rozmawialiśmy o tym, zaproponuję rozwiązania kompleksowe, systemowe w zakresie planowania przestrzennego i do tego się zobowiązuję w ramach tzw. kodeksu urbanistyczno-budowlanego, takie rozwiązania systemowe państwo otrzymają. Niepotrzebne są te uwagi o partyjnych aparatczykach. Natomiast chcę jeszcze raz podkreślić, że ja jako samorządowiec wiem, co znaczy planowanie przestrzenne. panie pośle, panie marszałku, i chcę powiedzieć, że tam, gdzie pracowałem w samorządzie, tam było 100% planu. Rekomenduję to rozwiązanie każdemu: prezydentowi Warszawy, prezydentowi Bydgoszczy, prezydentowi Lublina, prezydentowi Poznania, prezydentowi Gdańska, prezydentowi Krakowa, czyli tym wszystkim, którzy dewastują przestrzeń w swoich miastach, a dzisiaj waszymi głosami próbują odwracać kota ogonem. Czy będziemy zaganiać spółki Skarbu Państwa do budowy mieszkań, pyta poseł Truskolaski.

Tak. Oczekiwanie jest takie, aby te inwestycje były na dużą skalę i były realizowane jak najszybciej. Takie jest oczekiwanie Polaków. Chcemy rozpocząć w roku przyszłym realizację 100 tys. mieszkań w ramach programu „Mieszkanie+”, ale nie zlekceważyliśmy konsultacji społecznych. Rozmawialiśmy z izbami, z ekspertami, z ruchami miejskimi, a 27 kwietnia 2018 r. zrobiliśmy spotkanie podsumowujące konsultacje publiczne, gdzie było kilkaset osób z różnych stron Polski i poważnie rozmawialiśmy o tej ustawie, uwzględniwszy wcześniej niemal wszystkie kierunkowe postulaty i samorządu, i strony społecznej. Co więcej, powiem, że dzięki tej ustawie nie będzie tak, że powstaną wyłącznie bloki, bo będzie tak, że będzie obowiązek przestrzeni wspólnej - to jest wprost napisane w standardach - przy realizacji inwestycji mieszkaniowej właśnie będzie miejsce na tereny rekreacyjne czy na boiska. Dzięki temu w Polsce przestrzeń będzie bardziej spójna, bardziej funkcjonalna i bardziej wygodna dla tych wszystkich, którzy mieszkają w Polsce, bo piękno nas wyzwoli, jak mówił w swoim exposé, cytując Scrutona, premier Mateusz Morawiecki. Bardzo dziękuję. Panie ministrze, pan absolutnie nie zrozumiał, o czym mówiłem.

Teraz wyobraźmy sobie sytuację, w której takie budynki są w okolicy. Zgodnie z art. 19 nowa inwestycja będzie mogła mieć dwie kondygnacje więcej, tak? 50%.

Tak, tak mówimy i tak ewidentnie wynika z przepisów tej ustawy. Rozumiem, o czym pan mówi: że ostateczną decyzję będzie mógł podjąć samorząd, czyniąc wyłom w planie zagospodarowania przestrzennego, ale cały czas mówimy o tym, że ta ustawa jest m.in. właśnie dlatego zła, że tworzy wyłomy [[Dzwonek]] w planie zagospodarowania przestrzennego. Jeśli to jest wyłom, to rzeczywiście nie zrozumiałem, bo jedynym wyłomem jest możliwość dowozu dzieci do szkoły. Panie Pośle! To samorząd jest gospodarzem terenu, to samorząd odpowiada za przestrzeń publiczną. Myśmy w pierwotnej wersji planowali, aby to była decyzja lokalizacyjna wojewody. Samorząd przekonał nas. że jest to kwestia ustrojowa, i myśmy te racje podzielili. Ta zmiana, która zresztą właśnie na wniosek samorządu została wprowadzona do projektu ustawy, daje samorządom możliwość reagowania na lokalne uwarunkowania, tzn. na terenach bardziej zurbanizowanych te standardy mogą być bardziej rygorystyczne, można np. skrócić konieczną odległość do komunikacji publicznej czy szkoły, natomiast na terenach mniej zurbanizowanych samorządy oczekiwały, że damy im możliwość zwiększenia tych odległości, a wczoraj na posiedzeniu komisji deregulacyjnej przedstawiciel Związku Miast Polskich mówił, żeby w ogóle nie było procentowego ograniczania zwiększania bądź zmniejszania tych odległości, bo myśmy wpisali 50%, tylko żeby dać całkowitą swobodę samorządom w określaniu tych odległości, bo to samorząd - jeszcze raz powtórzę - jest gospodarzem miejsca i są samorządy, które będą z tego korzystały i które czekają na tę ustawę. Nie chcę być odpytywany, ale bardzo chętnie przekażę i pisemne stanowisko jednego ze związków samorządowych, i stanowiska wielu prezydentów miast, którzy popierają ten projekt, bo naprawdę nie wszyscy prezydenci w Polsce mają.

W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do przedłożonego projektu ustawy poprawki, proponuję, aby Sejm ponownie skierował ten projekt do Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji w celu przedstawienia sprawozdania.

Dziękuję państwu. 3 minuty przerwy.

Wznawiam obrady. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 30. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2678 i 2714) Proszę pana posła Tomasza Latosa o przedstawienie sprawozdania komisji. Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! W imieniu Komisji Zdrowia mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, odpowiednio druki nr 2678 i 2714. Na posiedzeniu komisji rozpatrzono projekt ustawy. Uzyskała ona pozytywną opinię komisji. Warto podkreślić, że w trakcie procedowania została zgłoszona poprawka, która dotyczy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a która doprecyzowuje przepisy mające na celu stworzenie szczególnych uprawnień dla dzieci między 3. a 16. rokiem życia, jeżeli chodzi o dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności, jeżeli chodzi o dostęp do świadczeń medycznych. Poprawka ta została przyjęta jednomyślnie na posiedzeniu komisji, co przyjmuję też z dużą satysfakcją z racji tego, że tę poprawkę przedstawiałem i dzięki niej nie będzie już żadnych wątpliwości, że również dzieci będą beneficjentami ustawy, która została przez Sejm przyjęta w maju.

Należy podkreślić, że m.in. w efekcie tego podpisanego porozumienia w przypadku rezydentów, którzy zdecydują się na dalszą pracę w granicach Polski, pracę, która będzie tutaj świadczona, będzie możliwość w ramach rezydentury uzyskania dodatkowego dofinansowania: w specjalnościach deficytowych w wysokości 700 zł, a w pozostałych specjalnościach w wysokości 600 zł. Ta ustawa również reguluje inny ważny postulat, jakim jest kwestia wynagrodzeń w przypadku lekarzy specjalistów. I tak w przypadku pracy u jednego świadczeniodawcy - myślę o świadczeniodawcy publicznym - docelowo ta wysokość ma wynosić 6750 zł brutto.

Wszystko to było omawiane w czasie posiedzenia komisji i raz jeszcze rekomendując Wysokiej Izbie przyjęcie tej ustawy, chcę podkreślić, że głosowanie komisji nad całą ustawą odbyło się bez głosu sprzeciwu, były głosy za i głosy wstrzymujące się. Dziękuję bardzo. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół. Jako pierwsza w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość pani poseł Anna Kwiecień. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości przedstawić opinię co do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Przepisy projektowanej ustawy zawierają rozwiązania będące wynikiem dialogu społecznego, którego efektem jest porozumienie ministra zdrowia z przedstawicielami Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy z dnia 8 lutego 2018 r., zwanego dalej porozumieniem. Strony porozumienia jako podstawowy cel swoich działań określiły zwiększenie dostępności świadczeń opieki zdrowotnej oraz poprawę ich jakości poprzez zwiększenie finansowania publicznego systemu ochrony zdrowia oraz zagwarantowanie lepszych warunków pracy kadrom medycznym.

Tym samym w krótszym okresie możliwe będzie sfinansowanie większej liczby udzielonych świadczeń. W ustawie przyjęto, że lekarz odbywający specjalizację w dziedzinie nieokreślanej jako priorytetowa otrzyma zwiększenie wynagrodzenia o kwotę w wysokości 600 zł miesięcznie, natomiast w dziedzinie określanej jako priorytetowa - 700 zł miesięcznie. Aby otrzymać wyższe wynagrodzenie zasadnicze, lekarz będzie musiał złożyć w podmiocie prowadzącym szkolenie specjalizacyjne podpisane zobowiązanie do przepracowania w kraju minimalnego okresu - mówimy tu o łącznie 2 latach w ciągu kolejnych 5 lat następujących po zakończeniu szkolenia specjalizacyjnego. Środki niezbędne do podniesienia wynagrodzenia zasadniczego będą przekazane do podmiotu prowadzącego szkolenia specjalizacyjne w oparciu o umowę zawartą z Ministerstwem Zdrowia. Wprowadzane przepisy realizują jeden z punktów porozumienia i wychodzą naprzeciw problemom dotyczącym zarówno stworzenia mechanizmów zabezpieczających przed emigracją lekarzy wykształconych w Rzeczypospolitej Polskiej, jak i sytuacji finansowej lekarzy odbywających specjalizacje w ramach rezydentury. Oczekuje się, że przyjęte rozwiązania z jednej strony powinny tworzyć większą zachętę dla lekarzy do rozpoczęcia specjalizacji, a jednocześnie przez podpisywanie zobowiązania do przepracowania w kraju określonego czasu po zakończeniu specjalizacji tworzyć lepsze perspektywy w zakresie zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych obywateli. W projekcie zakłada się uwzględnienie programowych dyżurów medycznych w kosztach finansowania umów rezydenckich, co moim zdaniem jest bardzo dobrym rozwiązaniem z uwagi na to, że świadczeniodawcy czy placówki specjalizujące ograniczali, można powiedzieć, dostęp lekarzy rezydentów do tych dyżurów. Takie rozwiązanie z jednej strony poprawi nieco kondycję finansową podmiotów zaangażowanych w kształcenie specjalizacyjne, co powinno również przyczynić się do zwiększenia ich liczby, a z drugiej strony da ministrowi zdrowia dodatkowe narzędzia oddziaływania, jeśli chodzi o prawidłowość realizacji tego elementu szkoleniowego. W projektowanej ustawie określa się sposób przekazywania do podmiotów leczniczych będących świadczeniodawcami, które zawarły z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy obejmujące udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach całodobowych lub całodziennych, środków finansowych na pokrycie kosztów podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych lekarzy specjalistów - to jest kolejny bardzo ważny postulat realizowany na podstawie stosunku pracy - do poziomu 6750 zł oraz kosztów podwyższenia należnego z tytułu dodatku za wysługę lat.

Dziękuję bardzo. Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu Platformy Obywatelskiej w sprawie procedowanego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, druk nr 2678. Jako główny cel tej ustawy przyjmuje się zwiększenie dostępności usług medycznych oraz poprawę ich jakości, w tym także poprawę finansowania kadr medycznych. środków finansowych na ochronę zdrowia jest absolutnie niekwestionowaną pilną potrzebą, ale propozycja przedłożona przez rząd, zakładająca wzrost do 6% PKB przy obecnym finansowaniu na poziomie 4,7%, jest niezadowalająca ze względu na rozłożenie tego w czasie, do roku 2024. Rozwój medycyny, postęp, innowacyjność terapii, ale także starzejące się społeczeństwo, epidemia chorób przewlekłych, cywilizacyjnych nakładają na nas, polityków, obowiązek, a nawet konieczność wprowadzenia nowych rozwiązań systemowych, zwiększenia dostępności świadczeń zdrowotnych, a także finansowania. Przy założeniu wieloletniego i powolnego wzrostu nie zbliżymy się do standardów europejskich, a wręcz będziemy się od nich oddalać.

Chcemy wszyscy jednogłośnie wzrostu finansowania i poprawy jakości usług, ale musi to nastąpić znacznie szybciej.

Tutaj niespodzianka, gdyż wydawałoby się, że sprawa jest oczywista, porozumienie jest podpisane, a jednak wczorajsze stanowisko Naczelnej Izby Lekarskiej było zachowawcze, a młodzi lekarze rezydenci jasno mówili, że nie zostały spełnione wszystkie postulaty zawarte w porozumieniu. Rząd na to odpowiedział: przyjmijmy to, co jest, a rozmowy będą trwały dłużej, może rok, może dwa, nie wiadomo. To nie brzmi dobrze. Ta ustawa niestety nie realizuje wszystkich ustaleń, tak więc obietnice rządowe stały się niewiarygodne. Dodatkowo wrzucono także poprawkę - zresztą bardzo ważną i dobrze, że ona została zgłoszona - dzięki której zapewnia się prawo do bezpłatnego dostępu do wyrobów medycznych dzieciom, ale kuriozalny jest fakt, że wprowadza się to od 1 lipca br. No cóż, zostaliśmy przyzwyczajeni do tego, że szybko, błyskawicznie pracujemy, że łamane jest prawo, że nagina się procedowanie zgodnie z potrzebami interpretacyjnymi. Teraz okazuje się, że nie zawsze obietnice, które są negocjowane przy stole, to jest rzeczywistość i prawda. Rozumiemy więc dobrze stanowisko młodych lekarzy, bo dla nich to nie jest rzeczywiście dobra lekcja. Podsumowując, ten kierunek zmian absolutnie popieramy, wzrost finansowania także, ale obawy budzi ryzyko w postaci przewlekłego czasu i sposobu procedowania. Dlatego też Platforma będzie głosowała za przyjęciem tej ustawy, ale równocześnie składamy poprawki. Mamy nadzieję, że zostaną one przyjęte i że będziemy dalej procedować nad tym projektem. A tymi poprawkami chcemy pomóc zrealizować obietnice złożone przez rząd. Dziękuję bardzo. Składam na ręce pana marszałka poprawki. Dziękuję bardzo.

Wysoka Izbo! Przez wiele, wiele lat zapominano w Polsce o tym, że aby dobrze funkcjonował system ochrony zdrowia, niezbędna jest odpowiednia liczba lekarzy, ale też i pielęgniarek. Nie nastąpiła oczekiwana przez system zmiana pokoleniowa.

Ustawa, która w tej chwili jest przedmiotem naszych obrad, napawa mnie lekkim optymizmem, bo zmiany faktycznie idą w dobrym kierunku.

Rozumiem, że te posunięcia, czyli tak naprawdę podwyższenie płac lekarzom rezydentom, mają taki cel, żeby ten exodus zatrzymać, mam jednak obawy, czy to są podwyżki wystarczające, aby te trendy zmienić na stałe.

Nie jest to spełnienie wszystkich marzeń, ale od czegoś trzeba zacząć. Dziękuję bardzo. Teraz głos ma pan poseł Marek Ruciński, klub

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Wielokrotnie na tej sali plenarnej oraz w trakcie posiedzeń Komisji Zdrowia poruszaliśmy problemy organizacji systemu ochrony zdrowia. Większość tych dyskusji była wymuszona akcjami protestacyjnymi różnych grup zawodowych, których przedstawiciele słusznie domagali się godnych warunków pracy - podkreślam: pracy - i płacy, zwracając jednocześnie uwagę na coraz większy problem związany z brakiem kadry medycznej, który finalnie dotyka polskiego pacjenta, zatem także nas wszystkich. Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, o którym dzisiaj dyskutujemy, powstał na mocy porozumienia z reprezentantami nie całego środowiska, a jedynie jednej grupy, niezwykle ważnej, którą jest Porozumienie Rezydentów OZZL. W lutym, gdy wypracowano 21 punktów wspólnej deklaracji kończącej trwający od wielu miesięcy protest, przekonywano, że to początek dobrych zmian w systemie ochrony zdrowia. Minister deklarował wzrost nakładów na ochronę zdrowia. Mam jednak wątpliwości: Jak włączanie do budżetu odpisu dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz kosztów związanych z Funduszem Rozwiązywania Problemów Hazardowych wpłynie na zwiększenie dostępności świadczeń medycznych dla pacjentów? Jakich świadczeń będzie więcej? Wczoraj na posiedzeniu Komisji Zdrowia zabrakło jasnych odpowiedzi na te pytania. Rozmawiając o tym projekcie ustawy, warto także podnieść inne kwestie. Na co zostaną przeznaczone dodatkowe środki w kwocie ok. 2 mld zł?

Jaki jest harmonogram działań mających na celu urealnienie koszyka świadczeń gwarantowanych oraz ich wyceny zgodnie z § 12 porozumienia? Jaki jest harmonogram realizacji pozostałych zobowiązań przyjętych w porozumieniu? To są pytania z mojej interpelacji, którą skierowałem do ministra zdrowia w dniu 1 marca tego roku. Blisko miesiąc od wejścia w życie porozumienia spodziewałem się już wstępnych planów jego realizacji. Odpowiedzi na te, wydawałoby się, proste pytania nie otrzymałem jednak do dzisiaj. Mimo że naganne w mojej ocenie jest zawieranie porozumienia jedynie z częścią środowiska oraz wykluczanie z dialogu innych przedstawicieli zawodów medycznych i niemedycznych, to jako lekarz praktyk dostrzegam złożoność problemu oraz potrzebę dofinansowania polskiego systemu ochrony zdrowia. Deklarowany przez ministerstwo nawet niewielki wzrost nakładów jest potrzebny, by Polska mogła wyjść z grupy państw Unii Europejskiej, które na ochronę zdrowia przeznaczają najmniej środków. Chcemy wierzyć w złożone wczoraj przez ministra zdrowia deklaracje, że to pierwszy etap zmian, a rozmowy z pozostałymi grupami zawodowymi zostaną wkrótce podjęte. Wiemy też, że projekt ustawy popierany jest przez środowisko medyczne. Będziemy zatem głosować za jego przyjęciem, licząc na to, że Ministerstwo Zdrowia zachowa się w sposób elegancki i podejmie się realizacji złożonych obietnic.

Bardzo dziękuję.

Wysoka Izbo! Wiele moi przedmówcy powiedzieli na temat dochodzenia do tej ustawy, dochodzenia do rozwiązań i do przyjęcia ich w Wysokiej Izbie.

Ale jest ona wywalczona przez środowisko lekarzy rezydentów. Oni w październiku 2017 r. prowadzili prawie miesięczny strajk głodowy, którego efektem było przyjęcie ustawy zwiększającej nakłady na ochronę zdrowia w Polsce do 6% PKB. To jest heroiczna walka, którą młodzi ludzie, decydując się na strajk głodowy, na taką najbardziej ekstremalną, najtrudniejszą formę zwrócenia uwagi, zawalczenia o swoje postulaty, podjęli, ponieważ widzieli bezczynność i bezradność dzisiaj rządzących.

Ponad 50 osób prowadziło strajk głodowy. Chcę przypomnieć te liczby, bo to są prawdziwi autorzy tych rozwiązań.

Dobrze, że dochodzi do refleksji również u rządzących i że doszło do zawarcia porozumienia - już po objęciu przez pana ministra Szumowskiego funkcji ministra zdrowia. Można było to też zrobić jeszcze w listopadzie, gdy głosowano nad pierwszą wersją ustawy.

Patrzę na pana przewodniczącego Latosa. Wiem, że on by chciał być wtedy za. To jest ten zawsze dobry duch w PiS-ie w sprawach medycznych, mam nadzieję, że kiedyś ta dobra intencja obejmie większą grupę posłów PiS-u. Mamy teraz do czynienia z taką samą poprawką. Mam nadzieję, że dzisiaj PiS zachowa się w głosowaniu inaczej. Powody trudnej sytuacji w ochronie zdrowia, które były omawiane i przez pana posła Rucińskiego, i przez pana posła Kozłowskiego, skupiają się w głównych trzech punktach. Starzenie się społeczeństwa, gigantyczne wyzwania opieki nad pokoleniem seniorów, pokoleniem osób w dostojnym wieku, potrzeby medyczne, które z dnia na dzień się zwiększają, nowe technologie medyczne, dostęp do nowych badań, zarówno badań laboratoryjnych, jak i badań obrazowych, do nowej diagnostyki i procesu terapeutycznego powodują, że pomimo wzrostu wydatków, który nastąpił nie od 2 lat, tylko następuje od dekady - przybywa co roku środków w Narodowym Funduszu Zdrowia, wynika to z ilości składek odprowadzanych przez naszych rodaków - wciąż nie mamy potrzeb zaspokojonych na takim poziomie, na jakim oczekują tego Polacy. I problemy kadrowe, to jest rzecz kluczowa również w tym rozwiązaniu. Dobrze, że jest myślenie o tym, jak zatrzymać, jak zachęcić do pozostania w Polsce jak najwięcej lekarzy. Brakuje rozwiązań dla pielęgniarek, brakuje rozwiązań dla fizjoterapeutów, dla ratowników medycznych. To jest ułomność prowadzonej przez was polityki zdrowotnej. Kolejna rzecz, słyszeliśmy wielokrotnie obietnice powrotu Polaków do Polski z Wielkiej Brytanii, z Holandii, z innych krajów europejskich.

Ile pielęgniarek, ilu ratowników medycznych? A ilu wyjechało?

Jako Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego - Unii Europejskich Demokratów popieramy zaprezentowane rozwiązania, ale będziemy też monitorować, czy są kontynuowane [[Dzwonek]] wobec innych grup zawodowych. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Koła Poselskiego Wolni i Solidarni przedstawię stanowisko wobec rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Niedofinansowanie i lata zaniedbań przede wszystkim skutkują niedostateczną ochroną zdrowia i życia naszych obywateli, ale były również przyczyną protestu rezydentów, który po wielu długich i ciężkich rozmowach zakończył się wypracowaniem kompromisu i podpisaniem porozumienia z ministrem zdrowia. Cieszy mnie, że omawiany dziś projekt ustawy wprowadza w życie szereg zawartych w porozumieniu rozwiązań. Wśród nich są: zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia do wysokości 6% PKB do 2024 r., dodatki pieniężne dla lekarzy odbywających specjalizację w wysokości 600 lub 700 zł miesięcznie, w zależności od tego, czy specjalizacja ta jest określona jako priorytetowa, oraz podwyższenie wynagrodzeń zasadniczych lekarzy specjalistów. Ponadto warto wspomnieć o uwzględnieniu, w określonej wysokości, godzin programowych dyżurów medycznych w kosztach finansowania umów rezydenckich, objęciu lekarzy i lekarzy dentystów ochroną prawną należną funkcjonariuszowi publicznemu oraz - co ze względu na obecną demografię naszego społeczeństwa wydaje się szczególnie istotne - zobowiązaniu lekarzy do przepracowania w kraju łącznie minimum 2 lat w ciągu kolejnych 5 lat następujących po zakończeniu szkolenia specjalizacyjnego. Nie dziwię się, że wiele z zaproponowanych rozwiązań obejmować będzie lekarzy, którzy praktykują w podmiotach leczniczych, które mają zawarte umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Podzielam opinię, że celowe jest kierowanie wsparcia i dodatkowego strumienia finansowania tam, gdzie będzie mogło z tego skorzystać najwięcej świadczeniobiorców, a podmioty te są właśnie takim miejscem. Ograniczenie to nie zmienia faktu, że ustawa ta w sposób pozytywny oddziałuje na warunki pracy kadry medycznej, które powinny być godne i bezpieczne. Jest to jeden z kluczowych czynników prawidłowego funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Jestem przekonana, że procedowane dziś regulacje zgodnie z założeniem zwiększą komfort pracy lekarzy, a przez to poprawią również jej jakość. Rozwiązania zawarte w ustawie będą miały także duży wpływ na zwiększenie powszechnego dostępu do świadczeń, m.in. przez zagwarantowanie wykwalifikowanej kadry, która zyskuje dodatkowe zachęty do pozostania w ojczyźnie.

Koło Wolni i Solidarni w pełni popiera procedowany projekt ustawy.

Wysoka Izbo! Warunki porozumienia zawartego z protestującymi lekarzami miały być wypełnione do 1 lipca. Nie dało się wcześniej przygotować i przeprowadzić ścieżki legislacyjnej. Nie bardzo rozumiem, co jest priorytetem, co jest dla was ważniejsze. Czy zdrowie i standardy leczenia Polaków są dla was istotne? Zajrzyjcie do Pszczyny, gdzie zlikwidowano szpital, zajrzyjcie do Żywca, gdzie nowy szpital buduje się już od 8 lat. Mówi się o nim od kilkunastu lat i końca nie widać, a warunki są skandaliczne. Nie wiem, czy ktoś z posłów życzyłby sobie przebywać w takim szpitalu. Mam pytanie: Dlaczego w tej ustawie jest zapis, że część zwiększonych nakładów na służbę zdrowia zamiast na świadczenia dla pacjentów ma być przeznaczona na agencję oceny [[Dzwonek]] technologii medycznych? Proszę o wyjaśnienie. Wysoka Izbo! Właściwie ponawiam pytanie z wczorajszego dnia, ponieważ nie do końca dostałam odpowiedź. Mianowicie interesuje mnie to, w jaki sposób będziecie państwo systematycznie, rok po roku, zwiększone środki wydawać na ochronę zdrowia, biorąc pod uwagę to, że głównym celem jest zwiększenie dostępności i poprawa jakości. W związku z tym chciałabym wiedzieć, jakie macie państwo plany, aby tę efektywność zwiększać i w jakiś sposób poprawiać jakość, ale interesują mnie także priorytety zdrowotne, o których państwo tyle mówicie. Rozpoczęły się, doskonale o tym wiem, debaty na temat zdrowia, ale niestety opozycja nie została zaproszona. Ten głos, który my chcieliśmy w tę dyskusję wnieść, państwa nie interesuje. W jaki sposób państwo zamierzacie zwiększyć dostępność świadczeń zdrowotnych, jeżeli lekarz będzie przypisany do jednego miejsca pracy? Panie Marszałku! Panie Ministrze! Celem projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw jest zapewnienie szerszego dostępu do świadczeń gwarantowanych w ujęciu materialnym. Przy skróceniu o rok okresu osiągnięcia poziomu nakładów w wysokości co najmniej 6% PKB, tj. do 2024 r., oznacza to również ich normalne zwiększenie w tym okresie w stosunku do aktualnie obowiązującej ustawy. Tym samym w krótszym okresie możliwe będzie sfinansowanie większej liczby udzielonych świadczeń. Niewątpliwie bardzo cieszy, że będzie więcej środków na rynku usług medycznych, natomiast chciałbym zapytać: Jaki jest stosunek rządu, pana ministra, do algorytmu podziału tych środków pomiędzy poszczególne oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia, który np. bardzo mocno dyskryminuje województwo opolskie, którego jestem przedstawicielem? Czy zastanawiają się państwo nad tym, [[Dzwonek]] jak to zmienić?

Dziękuję, panie marszałku. Wczoraj na posiedzeniu komisji, gdzie procedowano szybko, bo była wrzutka dotycząca osób niepełnosprawnych i niestety nie wyraziliście państwo zgody na to, żeby powołać podkomisję i spokojnie rozmawiać o tej ustawie, lekarze zwrócili uwagę na to, że ta ustawa nie realizuje porozumienia zawartego pomiędzy lekarzami a panem ministrem Szumowskim. Niestety to wszystko przekłada się na sytuację, z jaką spotykają się pacjenci w placówkach ochrony zdrowia. Coraz częściej słyszymy, że część oddziałów jest zamykanych, część odmawia przyjęcia pacjentów. Ogólnie rzecz ujmując, pacjent nie znajduje w systemie ochrony zdrowia tego, po co tam idzie, czyli opieki medycznej.

Kiedy państwo będziecie rozmawiać z przedstawicielami innych zawodów medycznych, [[Dzwonek]] żeby jesienią służba zdrowia nie stanęła? Pan poseł Zbigniew Pawłowicz, klub Platformy Obywatelskiej. Panie Marszałku! Panie Ministrze! W pkt 2 tego artykułu jest gwarantowane finansowanie dla lekarzy specjalistów do kwoty 6750 zł na pełen etat obliczeniowy. W związku z tym w pkt 3 tego artykułu od razu jest zapis, że lekarz uzyska to finansowanie, jeżeli złoży zobowiązanie, że będzie pracował u jednego świadczeniodawcy. Wynikiem tego jest kolejnych sześć punktów tej ustawy, które generują generalnie biurokrację, bo świadczeniodawca musi składać odrębną dokumentację odnośnie do tych zobowiązań, Narodowy Fundusz Zdrowia, minister zdrowia. Pytanie jest proste. Panie ministrze, korzystając z pewnych doświadczeń z przeszłości, czy nie lepiej byłoby zapisać, że tę kwotę wynagrodzenia brutto otrzymuje lekarz specjalista zatrudniony na pełnym etacie u jednego [[Dzwonek]] świadczeniodawcy. Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze!

Chciałbym w związku z tym zapytać pana ministra, jestem tym, nie ukrywam, zainteresowany, ponieważ od początku brałem udział w pracach nad tym, aby było to zwiększenie finansowania, czy już przed protestem rezydentów były prowadzone prace, były zresztą również określone deklaracje w Komisji Zdrowia, że takie zwiększenie finansowania jest przygotowane, czy też nie. Oczywiście rezydenci ten postulat podnosili i chwała im za to, natomiast chcę, aby była pełna jasność, że ten rząd miał intencję to podwyższenie nakładów wprowadzić, w przeciwieństwie do tego, co działo się w przeszłości. Bardzo dziękuję. Pani poseł Elżbieta Gelert, klub Platformy Obywatelskiej. Panie Ministrze! Moje pytanie dotyczy już poruszanego artykułu, m.in. w jaki sposób państwo chcecie tak naprawdę zwiększyć nakłady na świadczenia zdrowotne, zmniejszyć kolejki do 2020 r., jeżeli cały czas mówimy tylko i wyłącznie o nakładach z narodowego funduszu na personel medyczny. Czymże jest w tej chwili dopłacanie do kwoty 6720 zł, jeżeli nie zembalówką, tak jak poprzednio dla pielęgniarek, co jeszcze jest utrzymywane. Czyli w tej chwili będziemy dopłacać lekarzom specjalistom z narodowego funduszu, a co potem?

Panie Marszałku! Panie Ministrze! To dobrze, że rząd pracuje nad nowymi rozwiązaniami, ale obawiam się, że te rozwiązania są daleko niewystarczające i nie tylko nie zadowolą rezydentów, ale też nie poprawią sytuacji w służbie zdrowia, która jest coraz bardziej nabrzmiała. Mam pytanie. Ilu lekarzy brakuje w polskich szpitalach, w szpitalach publicznych? Informacje bowiem są alarmujące.

Ograniczenie zatrudnienia lekarzy do jednego świadczeniodawcy publicznego pogorszy dostęp do lekarzy specjalistów, który już dziś jest bardzo trudny. Mam pytanie.

Dziękuję. Czy pan minister chce zabrać głos? Bardzo proszę, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia

Najważniejsze jest to, że wreszcie zostanie zapewniony, ustawowo zagwarantowany wzrost nakładów na służbę zdrowia.

Ta ustawa gwarantuje to, że wraz ze wzrostem gospodarczym kraju, wraz ze wzrostem PKB te nakłady nie dość, że będą rosły, to będą rosły coraz szybciej.

Skoro od iluś lat mówimy o tym, że problemem w ochronie zdrowia są pieniądze, to ta ustawa, która gwarantuje stabilny, dodatkowo przyspieszony w stosunku do założeń z tamtego roku wzrost, musi to zapewnić.

Porozumienie określało też działania związane ze zwiększeniem naboru na studia wyższe i działania związane z zawodem asystentki medycznej czy też uwzględniało przegląd koszyka świadczeń gwarantowanych.

Odniosę się do pytań szczegółowych.

Jest to element nierozerwalny.

Ciężko mi sobie wyobrazić, że koszty tego organu nie są ujęte w nakładach na ochronę zdrowia. Padło kilka pytań dotyczących planu wydatkowania środków, podziału środków, skierowania ich do określonych grup świadczeniodawców.

Wydaje mi się, że gremium osób zaproszonych do debaty jest tak szerokie, włącznie z byłymi ministrami zdrowia z różnych opcji politycznych, że jednak ten balans jest zapewniony.

Mówimy o przyspieszonym tempie nakładów.

Oczywiście te rozmowy są prowadzone.

Toczą się rozmowy z różnymi grupami zawodowymi, a to, że te grupy nie zostały ujęte w ustawie, nad którą debatujemy, wynika wprost z zapisów porozumienia. Porozumienie określało zwiększone wynagrodzenia lekarzy rezydentów, lekarzy specjalistów, nie odnosiło się do wynagrodzeń pielęgniarek czy innych zawodów medycznych, co nie znaczy absolutnie, że praca i rozmowy w tych obszarach nie trwają.

Zgodnie z moimi informacjami faktycznie prace związane z ustawowym zwiększeniem nakładów - nie umiem odpowiedzieć dzisiaj, czy mówiliśmy o poziomie 6%, czy o innym, ale wydaje mi się, że o 6% - rozpoczęły się - według mojej wiedzy - w połowie 2017 r.

Przepraszam, powtórzyłem się. Chciałem się jeszcze odnieść do aspektu tego, czemu tyle biurokracji i czy nie dało się tego uprościć i powiedzieć: każdy lekarz specjalista, który pracuje u jednego świadczeniodawcy, powinien mieć zwiększone wynagrodzenie. Zwiększone wynagrodzenie u określonych świadczeniodawców wynika tak naprawdę z największych problemów, które dzisiaj ci świadczeniodawcy mają. Dzisiaj, i było to sygnalizowane również przez lekarzy rezydentów, największy problem mają szpitale. Mają problem z ułożeniem grafiku dyżurów przede wszystkim właśnie z tego powodu, że lekarze pracują w kilku miejscach i nie są chętni do dyżurowania w swojej jednostce macierzystej. Co więcej, odnosząc się i do tego aspektu dotyczącego różnych świadczeniodawców, i do tego aspektu, czy nie zabraknie nam lekarzy specjalistów i czy to nie spowoduje wydłużenia kolejek, chcę podkreślić trzy rzeczy. Po pierwsze, istnieje dobrowolność, jak już państwo zauważyli. Lekarz specjalista dzisiaj nie ma obowiązku podpisywania zobowiązania, że będzie pracował w jednym podmiocie, w swoim podmiocie macierzystym. Zdecydowanie może pracować w wielu, tylko że decyduje się na to świadomie i wtedy nie ma prawa do korzystania ze zwiększonego wynagrodzenia.

W związku z tym to nie przekłada się jeden do jednego na to, że nastąpi kryzys kadrowy w szpitalach.

Dziękuję bardzo. Sprawozdawca komisji też chce zabrać głos. Pan poseł Tomasz Latos. Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Ja przede wszystkim dziękuję wszystkim koleżankom i kolegom z komisji, że mimo tych moim zdaniem wyolbrzymionych zastrzeżeń jednak w ostateczności nikt nie był przeciwko tej ustawie, tej nowelizacji.

Radziwiłł na posiedzeniu komisji. Gdyby pan przewodniczący w poprzedniej kadencji złożył wniosek o zwiększenie nakładów do 6% PKB, wtedy z pewnością bym głosował za tym i przekonałbym klub Prawo i Sprawiedliwość do głosowania za tym. Niestety, w poprzedniej kadencji takiego wniosku nie było. Widać rozwiązanie problemów służby zdrowia czekało na rządy Prawa i Sprawiedliwości. Szanowni państwo, zrozummy jedną rzecz. Jeżeli jest mowa, również w tej ustawie, o zwiększeniu nakładów na ochronę zdrowia i jednocześnie zwiększeniu płac w ochronie zdrowia - mówiliśmy tu o lekarzach specjalistach, lekarzach rezydentach, jednym słowem o tym, że nie idzie to wprost na świadczenia medyczne, idzie na ludzi związanych z ochroną zdrowia, niezwykle ważnych, jako że to jest ważna część tego systemu, bo dobrze wynagradzany pracownik będzie z większą satysfakcją i chętniej wykonywał swój zawód - co do tego nie ma wątpliwości - to pamiętajmy, że podobną funkcję wypełnia agencja, zresztą agencja powołana w przeszłości. Natomiast, szanowni państwo, doceniajcie również to, co zbudowaliście, co było słuszne i jest potrzebne. Ale jednocześnie bez instrumentów, również finansowych, nie będzie mogło to funkcjonować. Ja już pomijam fakt, że to jest tam któryś jeden po przecinku, nie wiem, po iluś tam zerach, jeżeli chodzi o wydatki na ochronę zdrowia, ale dzięki tym wydatkom ileś tam, któraś tam liczba po przecinku, po zerach, dzięki temu mamy zabezpieczoną racjonalność wydawania miliardów w ochronie zdrowia. W związku z tym tak naprawdę per saldo działanie agencji służy pacjentom, służy racjonalności wydatków. Warto o tym pamiętać. I nie krytykujcie państwo tego, co sami akurat słusznie zaczęliście realizować.

Panie Marszałku! Przedłożony projekt ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów jest odpowiedzią na oczekiwania blisko 2,5 mln użytkowników wieczystych, Polaków, tych, którzy dzisiaj są właścicielami swoich mieszkań, swoich domów, ale jednocześnie są użytkownikami wieczystymi gruntów, na których te domy i mieszkania się znajdują. To ma gigantyczne znaczenie społeczne i ogromne znaczenie dla obrotu gospodarczego w Polsce. Wsłuchaliśmy się również w potrzeby samorządów, nie tylko Polaków, ale też tych, którzy sprawują władzę lokalną. Konsultowaliśmy się z nimi, aby ochronić również interesy samorządów. Dlatego dziękuję również stronie samorządowej za te uzgodnienia i za kompromisową postawę. Polacy mają silne przywiązanie do własności. Odpowiadamy na to i proponujemy Polakom, iż 1 stycznia 2019 r. prawo własności gruntów, na których polskie rodziny zaspokajają potrzeby mieszkaniowe, będzie dla tych wszystkich, którzy dzisiaj są użytkownikami wieczystymi. To rozwiązanie wpisuje się w program mieszkaniowy Prawa i Sprawiedliwości, którego najważniejszym komponentem jest program „Mieszkanie+” I to jest część programu „Mieszkanie+” Eliminujemy tym projektem całkowicie nieracjonalną sytuację, w której osoby będące właścicielami lokali i domów nie są jednocześnie właścicielami gruntu pod tym lokalem i domem. Rozwiązujemy palące problemy rodzin zamieszkujących w budynkach wielorodzinnych, w spółdzielniach mieszkaniowych czy we wspólnotach mieszkaniowych, w których dążenie do nabycia prawa własności do gruntu pod mieszkaniem napotyka od lat na poważne przeszkody, bardzo często niemożliwe do rozwiązania na gruncie obowiązującego prawa. Nie zapomnieliśmy również o właścicielach domów jednorodzinnych, którzy wobec braku w poprzednim systemie ustrojowym innych możliwości wybudowali swoje domy na gruntach publicznych obciążonych użytkowaniem wieczystym z obowiązkiem ponoszenia przez wiele lat opłat za korzystanie z tego gruntu. Należy przypomnieć, że prawo użytkowania wieczystego zostało wprowadzone do systemu prawnego w roku 1961 i pełniło wówczas funkcję surogatu prawa własności. W PRL obowiązywała zasada niepodzielności mienia państwowego, która nie pozwalała na przekazywanie własności gruntów państwa na rzecz obywateli. Ustanawiane wówczas prawo nie było przygotowane na zmiany, które szczęśliwie w Polsce zaszły. Także w przestrzeni polskich miast nie było ono przystosowane do tego, że po roku 1990 powstał w Polsce samorząd terytorialny. Dopuszczono bowiem nabywanie własności gruntów od Skarbu Państwa i gmin. Korzystanie z formy prawnej, jaką jest użytkowanie wieczyste, przestało być zatem swego rodzaju przymusem. Jednak ta sytuacja wygenerowała kolejne problemy prawne i praktyczne, które ujawniły się zwłaszcza w przypadkach użytkowania wieczystego pod budownictwo mieszkaniowe. Pierwotnie bowiem prawo to było pomyślane przede wszystkim jako forma przekazywania gruntów spółdzielniom mieszkaniowym i nikt nie myślał wówczas, że w blokach spółdzielczych będzie możliwość wyodrębniania własności lokali. Ułomność konstrukcji prawnej użytkowania wieczystego widać szczególnie wyraźnie w przypadku udziałów w tym prawie związanych z własnością lokali. Obowiązujące przepisy, doktryna i orzecznictwo nie dały dotąd jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy w tej konstrukcji prawem głównym jest użytkowanie wieczyste, czy własność lokalu. Dyskusja ta ma wymiar nie tylko formalny, ale również praktyczny, bo od odpowiedzi na to pytanie zależą losy tych 2,5 mln użytkowników wieczystych, tzn. na pytanie, co się stanie z prawem odrębnej własności lokalu po upływie 99 lat użytkowania wieczystego. Uwłaszczenie obywateli i oddanie im własności oznaczają uniknięcie tego rodzaju komplikacji w przyszłości. Na gruntach zabudowanych budynkami wielolokalowymi dochodzi obecnie do absurdalnych sytuacji, w których mieszkańcy jednego bloku ponoszą opłaty za grunt w różnej wysokości, bo jedni się odwoływali, a drudzy się nie odwoływali do samorządowych kolegiów odwoławczych czy do sądów powszechnych. Wieloletnia praktyka funkcjonowania użytkowania wieczystego na terenach mieszkaniowych dowodzi, że to prawo nie spełnia założonej systemowo funkcji. Jego utrzymywanie jest całkowicie nieracjonalne. Zaproponowane przez rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego ustawowe przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności raz na zawsze zamyka te problemy prawne i problemy praktyczne, ujednolica prawo do gruntów z prawami do lokali oraz domów, zapewniając najsilniejsze prawo rzeczowe: prawo własności zamieszkiwanej nieruchomości. Wzmocnienie prawa do gruntu i skończenie z podwyżkami opłat rocznych zapewnią obywatelom naszego kraju poczucie stabilności prawnej. To jest rozwiązanie, które wpisuje się bezpośrednio w politykę obecnego rządu, także w politykę mieszkaniową w ramach programu „Mieszkanie+” Nie możemy jednak zapominać, że takie próby już podejmowano i one bardzo często były kwestionowane w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Nasz projekt nie powtarza błędów poprzednich inicjatyw ustawodawczych. Dokonaliśmy pogłębionej, pełnej analizy orzecznictwa i wyciągnęliśmy praktyczne wnioski.

Założenie to pozwoliło nam zdefiniować zakres gruntów konieczny do objęcia przekształceniem i uznaliśmy, że w pierwszej kolejności będą to grunty zabudowane budynkami jednorodzinnymi i wielorodzinnymi wraz z towarzyszącą zabudową i infrastrukturą umożliwiającą prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkaniowych. Zasadniczy cel projektu polega na usprawnieniu procesu całkowitej likwidacji prawa użytkowania wieczystego jako pozostałości po okresie realnego socjalizmu. Cel ten realizuje również instytucja zapisana w tej ustawie, tj. opóźnione przekształcenie użytkowania wieczystego z chwilą zabudowania gruntu budynkiem mieszkalnym. Skutkiem tego rozwiązania będzie stopniowe wygaszanie prawa użytkowania wieczystego na cel mieszkaniowy. Tym samym nie będą ponownie generowane problemy, z którymi dziś zmagają się obywatele. Zaproponowaliśmy przyjazny dla obywateli mechanizm odpłatności za przekształcenie.

Wartością dodaną jest to, że okres płatności za przekształcenie będzie krótszy niż okres wnoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego. Ponadto obywatele nie będą już uiszczali tych opłat jako użytkownicy wieczyści, tylko jako ich właściciele. Nie będzie konieczności sporządzania operatów szacunkowych, mieszkańcy nie będą zaskakiwani skokowymi podwyżkami. Jedyna możliwość wzrostu wartości tej opłaty to wskaźnik inflacyjny, to jest jedyna możliwość.

Gdyby skorzystał z ustawy z roku 2005 r., jeśli w ogóle mógłby z niej skorzystać, bo bardzo rzadko jest to możliwe, gdyż musi być powszechna zgoda, to zapłaciłby za to przekształcenie ok. 1400 zł.

Będziemy jako Prawo i Sprawiedliwość zachęcać również samorządy, aby udzielały takiej bonifikaty swoim mieszkańcom, po to aby Polacy chętnie wnosili te opłaty i aby to użytkowanie wieczyste przestało być raz na zawsze tematem, na który rozmawiamy. Potwierdzenie przekształcenia będzie następowało z urzędu w formie zaświadczenia. To zaświadczenie będzie wydawane albo przez starostę, albo przez burmistrza czy prezydenta, w zależności od tego, czy jest to teren Skarbu Państwa, czy teren samorządu. Wpis w księdze wieczystej będzie również następował z urzędu i będzie wolny od opłat sądowych. Mieszkańcy domów i lokali nie będą zatem zobowiązani ani do aktywności, ani do ponoszenia dodatkowych opłat sądowych w związku z ustawowym uwłaszczeniem. Dodam jeszcze, że zabezpieczyliśmy takie pieniądze na księgi wieczyste, że również w zakresie pracy sądów nie będzie z tym żadnego kłopotu.

Dlatego też te 20 opłat rocznych według stanu za 1 stycznia 2019 r. w żaden sposób nie pomniejsza dochodów samorządu z majątku, dochodów, jakie wpływają do samorządu z tytułu użytkowania wieczystego.

Najwięcej jest w Warszawie, gdzie sięgają one ok. 4% wszystkich dochodów. Uwzględniając głosy samorządów, nie objęliśmy przekształceniem z mocy prawa gruntów zabudowanych wyłącznie samodzielnymi garażami niezwiązanymi z zabudową mieszkaniową. Samorządy krytykowały ten pomysł, gdyż istniało bardzo duże ryzyko objęcia przekształceniem również gruntów pod garażami wykorzystywanymi na działalność gospodarczą, wynajmowanymi, a także wielkopowierzchniowymi komercyjnymi garażami wielostanowiskowymi. Pragnę jednak uspokoić właścicieli garaży, gdyż na mocy obecnie obowiązującej ustawy będą mogli skorzystać z tego trybu. A jeśli wprowadzimy rozwiązanie systemowe, co jest naszym zobowiązaniem i kolejnym etapem likwidacji użytkowania wieczystego, dojdzie również do likwidacji użytkowania wieczystego na terenach, na których znajdują się garaże. W ramach planowanych prac chcemy zapewnić, aby wszyscy mieli możliwość stania się właścicielami. Ale część gruntów to grunty, które są w użytkowaniu wieczystym przedsiębiorców. W związku z tym dla pewności prawnej przy rozwiązaniu systemowym będziemy konsultowali takie regulacje z Komisją Europejską. Będziemy również proponowali rozwiązanie w postaci zapewnienia innego prawa rzeczowego, niezbędnego do wprowadzenia w Kodeksie cywilnym, tak aby zapełnić lukę po użytkowaniu wieczystym. Do tego czasu zlikwidujemy użytkowanie wieczyste w odniesieniu do ok. 6% wszystkich gruntów Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste i 44% wszystkich gruntów gmin oddanych w użytkowanie wieczyste. Jestem całkowicie przekonany, że ta operacja przebiegnie sprawnie. Wierzę i w sądy, i w samorząd, i w tych mieszkańców, którzy będą chcieli skorzystać z bonifikat, wierzę, że uda nam się to zrobić sprawnie. Ale te wnioski, które wyciągniemy w pierwszym etapie, bo to jest 2,5 mln, docelowo 4 mln przypadków likwidacji użytkowania wieczystego, z pewnością będą bardzo ważne przy reformie systemowej, którą już dziś zapowiadam. A dzisiaj rozwiązujemy problem społeczny dotyczący, jeszcze raz to powiem, wszystkich właścicieli mieszkań i domów, którzy mają swoje mieszkania i swoje domy - wreszcie będą mieli pełną własność, bo będą mieli również własność tego gruntu, który pod tym domem, pod tym mieszkaniem się znajduje. Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj Wysokiej Izbie rekomendować prace nad tym projektem i przyjęcie tego projektu. I głęboko wierzę, że wszystkie kluby parlamentarne go poprą. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół. Jako pierwszy w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość głos zabierze pan poseł Bogdan Rzońca. Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Rząd opracował i przedłożył projekt ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów. Projekt zakłada zmianę prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i dotyczy gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielorodzinnymi.

Obecnie obowiązujące rozwiązania ustawowe są niewystarczające, a nawet w niektórych sytuacjach nie dają faktycznej możliwości przekształcenia prawa. Dlatego też przedkładany projekt jest szczególnie oczekiwany przez właścicieli lokali mieszkalnych położonych w budynkach wielolokalowych. Właścicielom takich lokali przysługuje udział w prawie użytkowania wieczystego gruntów. W takich przypadkach obowiązujące przepisy wymagają zgody większości dla przekształcenia, a jej uzyskanie jest z różnych względów bardzo utrudnione. Z tego powodu wiele rodzin zamieszkujących budynki wielolokalowe nie może uzyskać prawa własności gruntu pod budynkiem, w którym położony jest lokal. Projektowana ustawa likwiduje te bariery poprzez objęcie ustawowym przekształceniem wszystkich członków wspólnot mieszkaniowych, bez wymogu zgody na zmianę prawa. Ustawa obejmuje również właścicieli domów jednorodzinnych i - co bardzo ważne - kończy również czas niepewności obywateli co do wysokości opłat, jakie ponoszą za grunty pod mieszkaniami i domami. Obecnie bowiem dopłaty roczne za użytkowanie wieczyste są niejednokrotnie podwyższane w sposób skokowy i stanowią bardzo duże obciążenie dla budżetów domowych. Projekt zakłada, że przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności będzie potwierdzone zaświadczeniem wydawanym z urzędu. Przekształcenie będzie odpłatne. Obywatele będą ponosili roczne opłaty przez okres 20 lat od dnia przekształcenia. Przewidziano tutaj także stosowanie ulg w opłatach w formie bonifikat, a także możliwość jednorazowego wniesienia wszystkich opłat przekształceniowych jako opłaty łącznej. W odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w przypadku wniesienia opłaty łącznej zaproponowano bonifikaty obligatoryjne w wysokości od 60% do 10% w zależności od roku, w którym będzie wnoszona opłata roczna. Aby uwzględnić prawa samorządów, rząd zapewnił możliwość dokończenia wszczętych aktualizacji rocznych opłat z tytułu użytkowania wieczystego, w których wysokość ma wpływ na wysokość opłaty za przekształcenie.

Takie rozwiązanie zapewni w przyszłości brak problemów, które obecnie istnieją w związku gruntami mieszkaniowymi oddanymi w użytkowanie wieczyste, szczególnie w dużych miastach. Przedłożony projekt był szeroko uzasadniany, uzgadniany, konsultowany. Jest bardzo oczekiwany i zapewnia po prostu stabilne prawo polskim rodzinom w zakresie gruntów. Klub Prawo i Sprawiedliwość proponuje, by przedłożony projekt poprzeć. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przedstawiam opinię klubu Platformy Obywatelskiej dotyczącą rządowego projektu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów. Rząd PiS przedstawia nam następny projekt ustawy, której założenia są dobre, ale ich szczegółowe zapisy - niekoniecznie. Oczywiste jest, że wielu Polaków zyska dzięki tej ustawie, dlatego ją popieramy. Stracą natomiast swoje dochody samorządy, czyli na końcu też mieszkańcy. W ustawie zapisano, że każdy Polak będący użytkownikiem wieczystym gruntu, na którym posiada mieszkanie lub dom, zostanie właścicielem tego gruntu z mocy prawa po wniesieniu opłaty przekształceniowej. Ustawa daje możliwość uiszczenia tej opłaty przez kolejnych 20 lat lub w całości z góry. W przypadku użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa sytuacja jest jasna, bo za wniesienie opłaty w całości w pierwszym roku po przekształceniu każdy otrzyma 60% bonifikaty. Problem pojawia się w przypadku użytkowania wieczystego gruntu jednostki samorządu terytorialnego. Ustawa nie reguluje wysokości bonifikat. Ustalać je mogą rady gmin, powiatów i sejmiki województw. Część samorządów nie będzie zainteresowana wprowadzeniem bonifikat. Powstanie niesprawiedliwy system, który mieszkańcowi jednej gminy umożliwi uzyskanie bonifikaty, a ościennej, sąsiadowi, już nie.

Rząd nie mógł oczywiście nakazać gminom wprowadzenia bonifikaty, chyba że zaproponowałby sposób na pokrycie tych strat, bo dochody z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów są jednym z dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego. Tą ustawą rząd PiS-u likwiduje ten dochód. Odpowiedzialny rząd powinien zaproponować samorządowi pokrycie strat finansowych w postaci rekompensaty, a nie, tak jak obecny, przerzucać kolejne zadania na samorządy, nie zapewniając im na to środków.

Rekompensując z budżetu państwa straty samorządów, można by ujednolicić wysokość bonifikat na gruncie Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Kolejnym dziwnym rozwiązaniem tej ustawy jest wprowadzenie najwyższych bonifikat za wniesienie opłaty przekształceniowej w pierwszym roku po przekształceniu użytkowania wieczystego tylko od Skarbu Państwa, podkreślam: tylko od Skarbu Państwa, nie gminy. Wprowadziliście zachętę w postaci 60% bonifikaty tylko w pierwszym roku, żeby Polacy jak najszybciej wpłacili całą tę opłatę w 2019 r., gdy będziecie rozdawali publiczne pieniądze w kampanii wyborczej.

To wasza motywacja. Przypominam, że od 2020 r. w dochodach Skarbu Państwa zniknie pozycja: opłaty za użytkowanie wieczyste, ale was nie interesuje, co będzie po 2019 r., bo już teraz wiecie, że przegracie wybory parlamentarne. Potrzebujecie pieniędzy natychmiast, kosztem przyszłych dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Mimo zastrzeżeń, które przedstawiłam, Platforma Obywatelska popiera możliwość przejęcia na własność gruntów, które użytkują Polacy.

Panie Ministrze! Wysoka Izbo!

Każdy, kto ma dom, mieszkanie wie, że ta stara zasada: czyja ziemia, tego własność, jest bardzo istotna i bardzo ważna. Posiadanie mieszkania na własność z ziemią na własność to jest stabilność, pewność i gwarancja, że coś jest mojego i ma sens.

Własność, szczególnie w naszej kulturze, w tradycji polskiej, jest bardzo istotna, bardzo ważna. Tutaj pochylam się nad kwestią podatków. Każdy, kto płaci podatki, doskonale wie, że użytkowanie wieczyste z punktu podatkowego dla mieszkańca jest bardziej kosztowne. Oczywiście jest bardziej korzystne dla gminy, co nie zmienia faktu, że mieszkańcy ciągle są podatnikami i nawet jak będą mieli własność, własność tego gruntu, także będą płacić podatki, ale jednocześnie spadną, zmniejszą się obciążenia dotyczące ich utrzymania i płacenia podatków.

Kolejna sprawa. Ja nie wiem, czy do końca bym się przejmował tym, że mieszkańcy będą mieli lepiej. Z wszelkim szacunkiem, mówię to jako szef sejmowej komisji samorządu, mieszkańcy są po prostu najważniejsi. Mieszkańcy są najważniejsi, bo dla nich jest gmina. Esencją każdej gminy są mieszkańcy. Jeżeli mieszkańcy będą mieli łatwiej, taniej, prościej, to znaczy, że tak naprawdę to jest ten plus. Kolejna kwestia. Ja rozumiem, że w tym momencie spadnie, zmniejszy się liczba obowiązków w gminach z tego powodu.

Jednocześnie mam nadzieję, że to.

Zatem tak naprawdę mówimy o pewnym procesie. To jest dla strony rządowej ważna kwestia. Nie wiem, czy przypadkiem w domyśle nie mówimy już o podatku katastralnym. Jednocześnie myślę, że nowa ustawa o dochodach JST w najbliższym czasie powinna nam dać odpowiedź na pytanie, w jaki sposób gminy będą musiały szukać nowych pomysłów na finanse i swój rozwój. Pamiętajmy, mieszkańcy są najważniejsi.

Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Poselskiego Nowoczesna mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu wobec rządowego projektu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów. Celem projektu jest szybkie umożliwienie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na gruntach zabudowanych budynkami mieszkalnymi w prawo własności, w szczególności przez członków wspólnot mieszkaniowych. Problem przekształcenia użytkowania wieczystego w debacie publicznej jest obecny od dawna.

Warto też podkreślić, że na problemy związane z użytkowaniem wieczystym gruntów zbudowanych na cele mieszkaniowe zwracał uwagę również rzecznik praw obywatelskich w swoich sprawozdaniach.

Przyznała ona osobom fizycznym będącym w dniu 13 października 2005 r. użytkownikami wieczystymi gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe prawo przekształcenia własności wieczystego użytkowania w prawo własności. To prawo przysługiwało także spółdzielniom i właścicielom lokali mieszkaniowych wyodrębnionych w budynkach wielolokalowych, niemniej jednak, zresztą mówił już o tym pan minister, z uwagi na konieczność uzyskania wszystkich zgód właścicieli lokali ta możliwość często była. Musieli się wszyscy zgodzić.

Problem nasilił się po dokonaniu aktualizacji wyceny nieruchomości, która powodowała niejednokrotnie radykalne podniesienie opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie, która musi być ponoszona nawet przez kilkadziesiąt lat. Przedłożony przez rząd projekt ustawy uwzględnia też orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który na połączony wniosek Rady Miasta Szczecin, Rady Gminy Ustronie Morskie i Rady Miasta Poznania badał zgodność z konstytucją ustawy z 2005 r. Nie uwzględnił jednak kwestii podnoszonej przez organizacje samorządowe, które przypominają, że Trybunał Konstytucyjny uznał za niekonstytucyjne odgórne wywłaszczanie gmin. Przypomnę, że Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że w zakresie, w jakim dotyczy nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, jest niezgodny z art. 165 ust. 1 i 2 konstytucji. Ta sprawa była też przedmiotem wielu uzgodnień i prowadzonych rozmów ze środowiskami samorządowymi podczas konsultacji w przypadku tego projektu ustawy.

Jestem głęboko przekonany, że w dobrze pojętym interesie samorządów jest to, aby wprowadzały rozwiązania analogiczne do bonifikat określonych w ustawie dla Skarbu Państwa, że to leży, tak jak powiedziałem, w interesie gmin i reprezentantów, bo realizuje się cele mieszkaniowe wspólnoty swoich małych ojczyzn. Natomiast zgadzam się w pełni, że nie można było tego zastosować wprost w ustawie, bo musiałaby temu towarzyszyć, że tak powiem, pełna rekompensata z tytułu utraconych dochodów. A zatem ministerstwo przyjęło takie, a nie inne rozwiązanie, które w moim przekonaniu w pełni się tutaj broni. Warto też na zakończenie zauważyć, to też było zgłaszane, że jest problem - który się uwidocznił - rozbieżności między Ministerstwem Finansów a Ministerstwem Sprawiedliwości w zakresie pokrycia tych wszystkich kosztów. Trzeba to przypomnieć, bo minister sprawiedliwości stoi na stanowisku, że nie jest w stanie tego zadania zrealizować. Mając na uwadze wagę problemu, Klub Poselski Nowoczesna pomimo szeregu uwag popiera przedłożony [[Dzwonek]] projekt ustawy i opowiada się za dalszą pracą nad tym projektem.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego - Unii Europejskich Demokratów przedstawiam opinię co do procedowanego projektu ustawy z druku nr 2673. Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Jakże inaczej wygląda ten projekt niż projekt nie tak dawno rozpatrywany, jakże inaczej wygląda sama procedura legislacji.

Nie będę powtarzał tych założeń. Uważamy, że projekt ustawy jest w miarę spójny, określa cel, drogi dojścia do tego celu, mówi o okresach, o mechanizmach, mówi o wartościach i kwotach, które będą dotyczyły określonych grup użytkowników. Naszym zdaniem powinien dobrze wpisać się w zrealizowanie tego założenia, aby każdy był właścicielem, mógł być właścicielem swojego mieszkania. Tylko prośba i sugestia, panie ministrze.

Tylko czy nie moglibyśmy też uwzględnić tych, którzy będą chcieli dokonać tych wpłat, a nie dadzą rady w pierwszym roku? To takie ludzkie po prostu. Nie wszyscy będą mogli. Ja odnoszę się do tego, co jest zapisane. Nawet względem ludzi, to takie ludzkie podejście, pomijając inne kwestie.

1% czy 2% - możemy stwierdzić, że może to jest mało istotna, oczywiście niedecydująca o funkcjonowaniu samorządu kwota, ale przy 100 mln to jest 2 mln czy 1 mln, a też pewne zadania można by za to zrealizować.

Dziękuję bardzo. Do pytań zapisało się dziesięcioro pań i panów posłów. Wyznaczam czas pytania na 1 minutę. Nie ma pana posła. Pan poseł Wojciech Król, Platforma Obywatelska. Pani poseł Małgorzata Chmiel, Platforma Obywatelska. Panie Marszałku! Szanowni Państwo!

Rozmawiamy tutaj o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność na cele mieszkaniowe.

W wielu miastach tereny zostały kupione. Poza tym są różne opłaty, w zależności od tego, czy to jest pod usługi, czy to jest pod inne funkcje, szpitale, są różne prawa użytkowania wieczystego. Dziękuję. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Pan minister mówił trochę o tych garażach, ale ja mam bardzo konkretne pytanie. Wiele samorządów przekazywało w użytkowanie wieczyste grunty zabudowane garażami na 40 lat - na najkrótszy okres, na jaki może być ustanowione użytkowanie wieczyste.

Chciałabym zapytać: Jak będzie wyglądało przekształcenie tych gruntów w prawo własności? Czy będzie to możliwe i na jakich zasadach? Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Projekt ten zakłada, że z dniem 1 stycznia przyszłego roku użytkowanie wieczyste dla nieruchomości gruntowych pod budynkami mieszkalnymi tak naprawdę przestanie istnieć. Moje pytanie dotyczy bonifikat, przede wszystkim tych bonifikat, które będzie mógł ustalić samorząd. Jaka może być w tym przypadku maksymalna bonifikata uchwalona przez organy uchwałodawcze samorządu? Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Nie było wówczas woli politycznej ze strony koalicji rządzącej.

Ale tylko jedno pytanie.

Tak więc na pewno taki pomysł przekształcania na mocy ustawy będzie

Co w przypadku, kiedy takie wnioski zostały już złożone, kiedy czekają w gminie na rozpatrzenie?

Panie Ministrze! Jak wiadomo, na mocy tej ustawy zostanie zniesione prawo użytkowania wieczystego dla właścicieli budynków mieszkalnych, którzy staną się właścicielami tych gruntów. Rozumiem, że w momencie transakcji powinno już z automatu być nabywane prawo własności, a nie tylko kupowane prawo wieczystego użytkowania. W tym przedłożeniu nic o tym nie ma, ale rozumiem, że intencja jest taka, abyśmy całkowicie skończyli z wieczystym użytkowaniem na cele mieszkaniowe.

Pan poseł Marcin Święcicki, klub Platforma Obywatelska. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam dwa pytania. Jedno pytanie dotyczy tego, czy dajecie państwo samorządom dostatecznie dużą, powiedziałbym nawet, pełną elastyczność w zakresie stosowania ulg, ich terminów, wysokości, kwoty czy procentów.

Tak więc tutaj, żeby samorząd zastosował jakąś ulgę, musi mieć pełną elastyczność, tak żeby to było w miarę sprawiedliwie w ramach samorządu rozwiązane. Drugie pytanie.

Wysoka Izbo! Nie wiem, czy państwo zwróciliście uwagę, że wreszcie można było tutaj usłyszeć z ust pana ministra, że bardzo ważne jest coś takiego jak budżet domowy.

Czy ministerstwo przewiduje w dalszym ciągu prace nad takimi rozwiązaniami, aby również inne obiekty mogły być włączone w tę podstawę? Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan minister chce zabrać głos?

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dziękuję oczywiście za tę dyskusję, cieszę się z tej deklaracji poszczególnych klubów. Nie wiem, skąd pani poseł Chmiel wzięła 6 mld zł, naprawdę tego nie wiem. gruntów Skarbu Państwa nie ma. Powiedziała pani: 6 mld. Chcę zapewnić i pana przewodniczącego, i pana posła Sowę, że jesteśmy przygotowani do tej operacji. Naprawdę nie tylko z punktu widzenia tej operacji, w której 2,5 mln użytkowników wieczystych stanie się właścicielami, bo to jedno, ale w ogóle będzie dobrze, jak wzmocnimy sądy i księgi wieczyste w sądach, dla obrotu gospodarczego na zawsze. To chcę powiedzieć w sposób jednoznaczny. Chcę tylko powiedzieć, panie marszałku, że nasze środowisko polityczne, Prawo i Sprawiedliwość, będzie namawiać do tego, aby te bonifikaty były atrakcyjne dla mieszkańców Polski.

Tak, o tym za chwilę. Natomiast zwrócę się do pana posła Kotowskiego - oczywiście, że w kolejnych latach będzie można skorzystać z bonifikat w przypadku gruntów Skarbu Państwa, tylko myśmy zapisali ten mechanizm tak, iż w kolejnych latach będą one mniejsze, każdego roku o 10%. Co więcej, jeśli ktoś nie kiwnie palcem i nie wyjdzie z domu, także zostanie właścicielem, jak te raty z tytułu opłaty rocznej się zakończą, po 20 ratach. Nie musimy rekompensować żadnych dochodów, bo samorządy żadnych dochodów nie stracą. Rozumiem, że moglibyśmy mówić o budżecie roku 2040. Jeśli mówimy o innych usługach, to oczywiście stawki są różne. To będzie część rozwiązania systemowego, które zapowiadam. Tak jak powiedziałem, musimy mieć tutaj, po pierwsze, uzgodnienie w zakresie pomocy publicznej, zmiany w Kodeksie cywilnym, szereg rozwiązań, których trzeba dokonać, aby dokonać rozwiązania systemowego.

Pani poseł Masłowska - ja tutaj potwierdzam to, co pani poseł Masłowska powiedziała, i dziękuję jej za to, że w tej sprawie zawsze zabierała głos. Dzisiaj jest to efekt tych prac. Odpowiadam na jej pytanie: to spółdzielnia mieszkaniowa się przekształci w tej sytuacji, o której pani mówiła, ona będzie właścicielem, a dzierżawa będzie funkcjonowała dokładnie tak jak w tej chwili.

Będziemy na pewno przekonywać Polaków do tego, że dobra władza samorządowa ma wpływ na ich życie.

Nie będzie, panie pośle, mówię do posła Sowy, możliwości ustanowienia nowego użytkowania wieczystego w trybie tej ustawy, poza ustawą o KZN. Odpowiedziałem na wszystkie pytania.

Ja wyraźnie powiedziałam, że w 2017 r. do Skarbu Państwa z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów wpłynęło ok. 1 mld zł. A skąd te moje wyliczenia?

Sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju pan Artur Soboń. Mamy 2400 tys. użytkowników wieczystych, z czego tylko 400 tys. na terenach Skarbu Państwa, dlatego te wyliczenia są całkowicie fałszywe.

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić przygotowany przez rząd projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym. Zaproponowana nowelizacja ma uporządkować i ujednolicić w skali kraju zasady opodatkowania gruntów, przez które przebiega infrastruktura liniowa służąca do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów lub energii elektrycznej oraz infrastruktura telekomunikacyjna. W projekcie wprowadzono zasadę, że posadowienie tej infrastruktury na gruntach osób trzecich, z których przedsiębiorstwo liniowe korzysta w sposób ograniczony, nie wpłynie na wzrost podatków gruntowych. Do tej pory nie było przepisów regulujących wprost zasadę opodatkowania tych gruntów. W związku z tym dochodziło do sytuacji, że w sąsiednich gminach takie same grunty mogły zostać opodatkowane inną stawką podatku w zależności od przyjmowanej przez gminę interpretacji prawa. W niektórych gminach organy skarbowe traktowały posadowienie infrastruktury liniowej jako neutralne podatkowo, natomiast w innych gminach grunty, przez które przebiegała ta infrastruktura, były uznawane za zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, co wiąże się z naliczaniem najwyższej stawki podatku od nieruchomości. Taka sytuacja prowadzi do licznych sporów pomiędzy podatnikami, właścicielami infrastruktury liniowej i organami podatkowymi. W ostatnich latach ten problem był szczególnie widoczny w przypadku gruntów będących w zarządzie Lasów Państwowych, na których posadowione są linie elektroenergetyczne. W ostatnim roku organy skarbowe zaczęły klasyfikować grunty pod liniami elektroenergetycznymi na terenach Lasów Państwowych jako grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, a nie jak dotychczas - jako grunty leśne. Z danych Ministerstwa Energii wynika, że w 2017 r. nie więcej niż 5% gruntów pod liniami elektroenergetycznymi na terenach Lasów Państwowych było opodatkowane najwyższą stawką podatku od nieruchomości, natomiast w 2018 r. taka stawka może dotyczyć już nawet ponad 40% gruntów pod liniami.

Koszt podatku zostanie przeniesiony na przedsiębiorstwo energetyczne, które może uwzględnić ten wydatek w taryfie za usługę dystrybucji. W skali całego kraju w większości przypadków posadowienie linii elektroenergetycznych na gruntach osób trzecich nie wpływało i wciąż nie wpływa na zmianę klasyfikacji tych gruntów do celów podatkowych i nie skutkuje opodatkowaniem tych gruntów najwyższą stawką podatku od nieruchomości. Istnieje jednak ryzyko, że zmiana klasyfikacji gruntów rozciągnie się w przyszłości na pozostałe grunty leśne i grunty rolne. Z uwagi na przyjmowaną przez organy skarbowe argumentację zmiana klasyfikacji gruntów może rozpocząć się także w przypadku gruntów, przez które przebiega inna infrastruktura liniowa, np. gazowa, ciepłownicza czy telekomunikacyjna. Przy dokonywanej zmianie klasyfikacji nie jest brana pod uwagę specyfika korzystania z gruntu przez właścicieli urządzeń liniowych. Przedsiębiorstwa liniowe wykorzystują ten grunt wyłącznie w ograniczonym zakresie, odpowiadającym służebności przesyłu. Właściciel nieruchomości zazwyczaj może nadal korzystać z gruntu do podstawowych celów. Na gruntach pod liniami elektroenergetycznymi w lasach nadal może być prowadzona działalność leśna, np. w postaci plantacji choinkowych, natomiast na gruntach rolnych mogą być prowadzone uprawy rolne. W związku z powyższym grunt ten nie powinien zostać opodatkowany w taki sam sposób jak grunt zajęty przez typowe, kubaturowe przedsiębiorstwo. Nie jest przy tym także uwzględniany cel działania przedsiębiorstw dysponujących infrastrukturą liniową wymienioną w ustawie, jakim jest świadczenie usług użyteczności publicznej. Należy podkreślić, że zmiana sposobu opodatkowania gruntów, przez które przebiega infrastruktura liniowa, prowadziłaby do wzrostu cen usług świadczonych przez przedsiębiorstwa wykorzystujące tę infrastrukturę. Ministerstwo Energii szacuje, że o ok. 7 zł miesięcznie dla przeciętnego gospodarstwa domowego mogłaby wzrosnąć opłata za dystrybucję energii elektrycznej, gdyby wszystkie grunty pod liniami elektroenergetycznymi zostały opodatkowane najwyższą stawką podatku od nieruchomości. Wzrosnąć mogłyby także ceny gazu, wody, odprowadzania ścieków oraz usług telekomunikacyjnych. Podwyżki podatków gruntowych z pewnością pozytywnie wpłynęłyby na budżety gmin, na których terenach znajduje się duża ilość linii elektroenergetycznych lub innej infrastruktury liniowej, jednak nastąpiłoby to kosztem wszystkich odbiorców energii elektrycznej oraz innych mediów, w tym mieszkańców mniej zamożnych gmin. Pogłębiłoby to zróżnicowanie rozwoju poszczególnych regionów kraju w zależności od gęstości posadowienia infrastruktury. Wprowadzenie jasnych zasad opodatkowania gruntów, przez które przebiega infrastruktura liniowa, jest także bardzo istotne dla podatników podatków gruntowych. Dzięki tej nowelizacji właściciele lub użytkownicy wieczyści gruntów nie będą zobowiązani do zapłaty wyższego podatku wyłącznie dlatego, że przez ich grunty przebiegają urządzenia infrastruktury liniowej. Naliczanie najwyższej stawki podatku, odpowiedniej dla gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, byłoby w szczególności krzywdzące dla właścicieli gruntów leśnych, rolnych lub nieużytków. Prowadziłoby do sytuacji, w której właściciel sam nie prowadzi działalności gospodarczej ani nie czerpie korzyści w związku z posadowieniem na jego gruncie infrastruktury liniowej, a jest zobowiązany do zapłaty wielokrotnie wyższego podatku od gruntu. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Jestem przekonany, że wejście w życie przygotowanej ustawy jest niezbędne. Społeczne i ekonomiczne skutki ewentualnych podwyżek cen mediów dla obywateli oraz podwyżek podatków dla właścicieli gruntów, na których posadowiona jest infrastruktura liniowa, byłyby wyższe niż ewentualne korzyści, jakie osiągnęłyby gminy. Dlatego wnoszę o pozytywną ocenę tej ustawy i przyjęcie jej w zaproponowanym przez rząd kształcie. Dziękuję. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół.

tego projektu ustawy, ponieważ porządkuje pewne rzeczy, które są różnie interpretowane w różnych miastach. Ale jednak trzeba się zastanowić również nad tym, co pan minister zauważył.

Pan mówi, że 5% właścicieli miało problemy z tą ustawą, a teraz mówimy o 40%.

Bo wójt, który jest pod presją urzędnika skarbowego, szuka zabezpieczenia, czy przypadkiem nie pominął czegoś, co mogłoby być dodatkowym podatkiem. No też pewnie się boi, że działa w interesie... że nie w interesie władzy publicznej podejmuje taką, a nie inną decyzję. My poprzemy ten projekt ustawy, bo to jest działanie strażackie, gaszenie w danym momencie tego ogniska, które płonie. Tak po prostu nie powinno się prowadzić działalności. Wiemy, że inwestycje tzw. infrastrukturalne, liniowe zajmują bardzo dużą powierzchnię kraju, mimo że w pasie są wąskie. Ale też jest ograniczenie dostępu do terenu przez konieczne oględziny, przeglądy, remonty linii przesyłowych, dystrybucyjnych. Z tego dobra, z tej usługi korzystają wszyscy obywatele, więc powinno być to uporządkowane w taki sposób, żeby nie było zgrzytów, żeby nie było tak, że jeden właściciel jest traktowany zupełnie inaczej niż wszyscy pozostali. To trzeba uporządkować.

Bo mamy tutaj do czynienia z ustawą, która porządkuje istniejące obiekty infrastrukturalne. A ile problemów jest w planowaniu takich linii, które zabezpieczają bezpieczeństwo państwa, ciągłość dostawy energii elektrycznej, gazu, paliw płynnych? Ta ustawa jest konieczna i gdyby rząd podszedł poważnie do problemów, a nie działał doraźnie, gasząc to, co teraz płonie, to mielibyśmy czas na przedyskutowanie bez kampanii wyborczej, bez emocji politycznych ustawy, która była już przygotowywana. Przypomnę niektórym zainteresowanym, że były dwa warianty, zgodnie z którymi moglibyśmy dojść do celu. Namawiam pana ministra, aby w resorcie popracować nad tą kompleksową ustawą o inwestycjach rolniczych, o inwestycjach liniowych. Ustawa dotyczy trzech branż. Każda z nich po prostu ma swoje problemy. My jako Platforma Obywatelska poprzemy ten projekt.

Ale pan podziękował, panie pośle. W takim razie, bardzo proszę, głos zabierze poseł Paulina Hennig-Kloska, klub Nowoczesna.

Pani Marszałek! Panie i Panowie Posłowie! Panie Ministrze! Niejednoznaczność jakichkolwiek przepisów, na bazie których pracują czy to przedsiębiorstwa, czy to samorządy, nie jest dobra ani dla obywateli, ani dla gospodarki.

Niestety to pokazuje, dokąd prowadzi zbyt rygorystyczne podejście państwa m.in. do samorządów.

Tak naprawdę inwestor, planując jakiekolwiek inwestycje, nie może bazować na jednym biznesplanie, a w dalszej kolejności okazuje się, że zupełnie inne koszty są mu systematycznie naliczane od eksploatacji danego terenu.

Usługodawców tak naprawdę. Tak że zapewnienie stabilności finansowej przedsiębiorstw zajmujących się czy to przesyłem paliw ciekłych, czy to ciepłownictwem, czy to energetyką jest po prostu konieczne z takiego punktu widzenia, że to powoduje stabilność funkcjonowania samorządów, do których te podatki ostatecznie trafiają, a po drodze oczywiście również osób, które są ostatecznymi odbiorcami danych usług.

W gospodarce nic nie ginie, każda opłata najczęściej jest uiszczana przez obywatela. Dlatego Nowoczesna w gruncie rzeczy poprze dalsze prace nad tym projektem w komisji i oczywiście też na dalszym etapie będziemy mieli do pana ministra bardziej szczegółowe pytania, tak by dopracować projekt, który faktycznie nie tylko będzie odciążeniem sądów, bo pewne nieścisłości w interpretacji zazwyczaj kończą się postępowaniem sądowym, ale także jednocześnie będzie czytelny i ostatecznie rozwiąże wszystkie problemy dotyczące różnic w interpretacjach. Dziękuję bardzo. Teraz głos zabierze poseł Mirosław Maliszewski, Polskie Stronnictwo Ludowe - Unia Europejskich Demokratów. Wysoka Izbo! Zabierając głos w imieniu klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego - Unii Europejskich Demokratów na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym, sygnalizuję na wstępie, że będziemy ten projekt popierać w dalszym procedowaniu. Jest to projekt, który naszym zdaniem rzeczywiście ujednolica pod względem interpretacji sprawę podatku rolnego od urządzeń, które są posadowione na gruntach i które służą mieszkańcom. Chodzi przede wszystkim o urządzenia do przesyłu energii, energii elektrycznej, gazu ziemnego czy energii cieplnej, ale także chociażby o urządzenia telekomunikacyjne.

Ustawa mówi wprost, że jeżeli urządzenie jest zlokalizowane na gruncie niebędącym własnością tego, który tę energię przesyła czy który jest właścicielem takiego urządzenia, to on wtedy tego podatku nie będzie płacić. Jednocześnie jeżeli to urządzenie jest zlokalizowane na gruncie, który jest własnością takiego przedsiębiorstwa - co z kolei również jest zrozumiałe - taki podatek powinien być naliczany. Dobrze, że taki projekt został przedstawiony, bo zwłaszcza w ostatnich kilku latach rzeczywiście mamy problem z interpretacją naliczania podatku.

Bardzo często stojący słup czy urządzenie gazowe służące do dalszego tłoczenia gazu są na gruncie rolnika, na gruncie przedsiębiorcy i nie tylko przeszkadzają mu w prowadzeniu racjonalnej działalności gospodarczej, ale też wprowadzają szereg ograniczeń w zakresie inwestycji właściciela takiego gruntu, bo pod linią energetyczną, na linii gazowej czy nad linią gazową nie można realizować różnego rodzaju inwestycji.

Dlatego warto by się zastanowić, czy w kolejnej nowelizacji tej sprawy nie uregulować. W ostatnim czasie, w ostatnich latach bardzo wiele kontrowersji, oporu społecznego - i słusznie - dotyczyło tzw. specustaw, które mają umożliwić inwestorowi realizację strategicznych zadań.

Ostatnio słyszeliśmy o tym, bardzo mocno to wybrzmiało w przypadku kolejnej specustawy i kolejnego pomysłu, jakim jest budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Dla wielu z nich oznacza to konieczność przesiedlenia się w inne miejsce, ich zdaniem niekoniecznie za ekwiwalentną rekompensatę, a nikogo nie trzeba przekonywać - i o tym dzisiaj mówiono także w poprzedniej debacie - że święte prawo własności zostaje w tym przypadku naruszone. Nie ma nic gorszego, jak odsyłanie z danego terenu kogoś, kto mieszka na nim od pokoleń i stworzył tam on i jego rodzina szereg wartości. Kończąc, panie ministrze, Wysoka Izbo, ponieważ ten projekt wiele kwestii reguluje mimo tych zastrzeżeń, o których mówiłem wcześniej, klub Polskiego Stronnictwa Ludowego - Unii Europejskich Demokratów będzie go popierał. Głos teraz zabierze poseł Jacek Wilk, niezrzeszony. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Miejmy na uwadze to, że to jest łata na łacie na kolejnej łacie. Polski system podatkowy wymaga generalnej przebudowy, a właściwie skasowania go i zbudowania od nowa. Polski system podatkowy to jest chyba jedyna dziedzina prawa, która jest prawem stanowym, czyli takim jak w średniowieczu - zupełnie inaczej jest opodatkowany stan chłopski, zupełnie inaczej stan duchowny i zupełnie inaczej cała reszta, zwłaszcza przedsiębiorcy. Czyste prawo stanowe, jak ze średniowiecza. Mało tego, przecież mamy w Polsce podatek pogłówny. Mało kto o tym pamięta. Każdy przedsiębiorca co miesiąc musi płacić podatek pogłówny w postaci składek ZUS-owskich na ubezpieczenia społeczne w tej samej wysokości. To klasyczny podatek pogłówny. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Mogę się założyć, że pojawią się nowe interpretacje, wykładnie tego, co jest gruntem dla celów gospodarczych. Poza tym w ustawie jest mowa o infrastrukturze liniowej, a co z pozostałą infrastrukturą itd., itd. A drugi problem jest taki, że jakby zła filozofia przyświeca tej całej ustawie, dlatego że uważa się, że trzeba na siłę ujednolicać podatki lokalne. Wręcz przeciwnie, samorządy, władze lokalne powinny konkurować między sobą systemami podatkowymi. Taka powinna być filozofia. W jednych gminach czy na jednych obszarach samorządowych te podatki będą lepsze, w drugich gorsze, w jednych bardziej korzystne dla przedsiębiorców, w innych mniej. I to będzie zdrowa konkurencja podatkowa, dzięki której tak naprawdę system podatkowy w całości będzie się poprawiał. Głos teraz zabierze poseł Andrzej Szlachta, Prawo i Sprawiedliwość. Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość przedstawiam stanowisko wobec rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym. Potrzeba dokonania zmian tych ustaw wynika z konieczności doprecyzowania przedmiotu opodatkowania i sposobu jego klasyfikacji. Według projektu posadowienie infrastruktury służącej do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów lub energii elektrycznej oraz infrastruktury telekomunikacyjnej na gruntach nienależących do przedsiębiorstw, w skład których wchodzi ta infrastruktura, nie zmienia sposobu opodatkowania tych gruntów. Wobec braku jednoznacznych przepisów odnoszących się do sposobu opodatkowania gruntów dochodzi często do rozbieżności w ich stosowaniu przez organy podatkowe, czyli w tym przypadku przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta. W konsekwencji tego stanu rzeczy dochodzi do odmiennego opodatkowania tych gruntów w zależności od ich położenia. W ostatnim okresie ukształtowała się niekorzystna linia orzecznicza sądów administracyjnych, zgodnie z którą grunty, na których posadowiona została rzeczona infrastruktura, powinny być opodatkowane podatkiem od nieruchomości w wysokości przewidzianej dla gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. W oparciu o te orzeczenia przyjmowana jest przez organy skarbowe interpretacja, że sam fakt posiadania tej infrastruktury jest wystarczającą przesłanką dla klasyfikowania gruntów jako zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej. Taka interpretacja skutkuje tym, że podatnicy, czyli właściciele nieruchomości, pomimo że nie prowadzą działalności gospodarczej i nie czerpią z niej zysków, zobowiązani będą do opłacania wyższego podatku tylko przez sam fakt, że zgodzili się na udostępnienie gruntu na cele przesyłowe. Proponowane zmiany ustaw mają zniwelować wątpliwości w doktrynie i w orzecznictwie. Intencją dokonania zmian ustawowych jest wprowadzenie zasady, że ulokowanie na gruntach osób trzecich infrastruktury przesyłowej, z której przedsiębiorstwo będące właścicielem tej infrastruktury korzysta w sposób ograniczony, nie skutkuje zmianą sposobu opodatkowania tych gruntów. W przypadku gdy na tych gruntach oprócz umieszczonej infrastruktury prowadzona jest działalność gospodarcza, od tych gruntów będzie pobierana najwyższa stawka podatku od nieruchomości na dotychczasowych zasadach. Drugim celem regulacji jest zapobieżenie wzrostowi obciążeń finansowych przedsiębiorców posiadających infrastrukturę liniową. Propozycja zmian legislacyjnych jest zgodna z zapisaną w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasadą powszechności opodatkowania oraz zasadą równości i nie jest sprzeczna z prawem Unii Europejskiej. Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość popiera zaproponowane zmiany legislacyjne i wnosi o skierowanie przedmiotowego projektu ustawy do dalszego procedowania do Komisji Finansów Publicznych. Bardzo dziękuję za uwagę. Czy ktoś z pań i panów posłów chciałby się jeszcze dopisać do listy? Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Rządowe Centrum Legislacji oceniło, że projekt tej ustawy budzi wątpliwości co do zgodności z konstytucją, m.in. z art. 167 ust. 1, zgodnie z którym jednostkom samorządu terytorialnego zapewnia się udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań. W tym projekcie uszczupla się dochody samorządów, bez równoczesnego zmniejszenia ich zadań. Co więcej, w ocenie skutków regulacji ustawodawca przedstawił korzyści, jakie odniosą przedsiębiorstwa energetyczne na skutek wprowadzonych tą ustawą zmian, pominął jednakże całkowicie skutki finansowe tych zmian dla jednostek samorządu terytorialnego; skutki zostały oszacowane na 0 zł. Czy pan minister zgadza się z taką oceną RCL-u? Czy prawdą jest, że skutki tej ustawy będą bezpośrednio wpływały na wysokość dochodów jednostek samorządu terytorialnego, prowadząc do ich zmniejszenia? Jakie będą skutki finansowe dla samorządów na skutek wejścia w życie ustawy w ciągu najbliższych lat? Pytanie zadaje poseł Krzysztof Gadowski, Platforma Obywatelska. Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Panie ministrze, dobrze, że ta ustawa się pojawia w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy. Czy to były państwowe spółki, czy ten obywatel, który był właścicielem tego terenu? Czy po prostu organy, które ten podatek ustanawiały? Czy państwo wykonaliście jakieś inne ruchy, poza przygotowaniem tej ustawy? Potrzebna była może wykładnia dokonana przez urzędy skarbowe tego prawa podatkowego, jakaś interwencja regionalnych izb obrachunkowych, które kontrolują budżety gmin. Czy państwo wykonaliście taki ruch, czy po prostu była to informacja medialna, prasowa, która miesiąc czy półtora miesiąca temu pojawiła się w Polsce, o tym, że sądy zasądzają, że pojawiały się takie trudne sytuacje? Pytanie zada poseł Mirosław Maliszewski, Polskie Stronnictwo Ludowe - Unia Europejskich Demokratów. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W minionych 2 latach bardzo wiele emocji wzbudzały nowe inwestycje energetyczne, które były zapowiadane, m.in. jedną z nich była budowa nowej linii 400 kV, która miała połączyć nowy blok w elektrowni Kozienice z aglomeracją warszawską, określona jako linia Kozienice-Ołtarzew. Lokalizacja tej linii wzbudzała wiele kontrowersji, było masę protestów społecznych, zwłaszcza tych, na których działkach miały być posadowione słupy energetyczne, nad którymi miała przebiegać ta linia czy wreszcie tych, którzy znajdują się albo znajdowali się w bezpośrednim sąsiedztwie. Chciałem zapytać w związku z tym, korzystając z obecności pana ministra: Co z tą inwestycją dzieje się w tej chwili, na jakim ona jest etapie? Co z ustawą, w której ona jest zapisana? Czy ta inwestycja jest przewidywana w najbliższym czasie? Dziękuję bardzo.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Spoglądam na te pytania, które zostały zadane. Pan poseł Bańkowski: uszczuplenie dochodów gmin, niezrozumiałe wyjaśnienie i rozbieżności pomiędzy RCL-em. Takie wątpliwości były, dyskusja, która poprzedziła skierowanie tej ustawy w to miejsce, gdzie w tej chwili jesteśmy, spowodowała, że spojrzenie, optyka była następująca. My spoglądamy na uszczuplenie dochodów gmin w ten sposób: nie na jako hipotetyczne dochody gmin, które mogłyby się pojawić, tylko rzeczywiście na te, które faktycznie miały miejsce. Padło pytanie, że było tego mało przez wiele lat, pan poseł Czerwiński mówił, że dało się z tym żyć. orzeczenia sądu wskazujące na to, że można czerpać z tego tytułu korzyści.

Z tego powodu kierujemy do państwa ten projekt. Ona nie jest w gestii ministra energii bo to są Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Postaramy się zdobyć odpowiedź na to pytanie od właściciela, bo ta linia akurat nie podlega Ministerstwu Energii. Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję.

Wznawiam obrady. Prezydium Sejmu, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów, przedłożyło wniosek w sprawie zmian w składach osobowych komisji sejmowych, druk nr 2717. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjąłem decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego wniosku.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 W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjąłem decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący głosowanie nad tym projektem uchwały. Właściwe komisje przedłożyły sprawozdania o uchwałach Senatu w sprawie ustaw: - o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw, - o zmianie ustawy o własności lokali, - o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw, - o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, - o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw.

W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjąłem decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkty obejmujące rozpatrzenie tych sprawozdań. Właściwa komisja przedłożyła sprawozdania o uchwałach Senatu w sprawie ustaw: - o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, - o tachografach. Sprawozdania to odpowiednio druki nr 2704 i 2703.

Proponuję, aby w tych przypadkach Sejm wyraził zgodę na zastosowanie art. 54 ust. 5a regulaminu Sejmu oraz w przypadku sprawozdań komisji zawartych w drukach nr 2690, 2695, 2694, 2691 i 2715 wyraził zgodę na zastosowanie art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu. Sprzeciwu nie słyszę. Komunikat. Marszałek Sejmu zaprasza w dniu jutrzejszym, tj. 6 lipca, o godz. 14 na uroczyste otwarcie w Zamku Królewskim wystawy pt. „550-lecie Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej” Dziękuję. Dziękuję. Przypominam, że kluby złożyły wnioski o uzupełnienie porządku dziennego o punkty: - Informacja Rady Ministrów na temat społecznych skutków wprowadzenia w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin - zgłoszony przez Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego - Unii Europejskich Demokratów, Informacja prezesa Rady Ministrów na temat przyczyn rozwiązania zespołu śledczych zajmującego się śledztwem w sprawie wypadku samochodowego z dnia 10 lutego 2017 r. w Oświęcimiu, na skutek którego ucierpiała premier Beata Szydło - zgłoszony przez Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska. W związku ze zbliżaniem się terminu, o którym mowa w art. 173 ust. 5 regulaminu Sejmu, poddam pod głosowanie wniosek o uzupełnienie porządku dziennego o te punkty. Przypominam, że zgodnie z art. 173 ust. 4 regulaminu Sejmu głosowanie to nie jest poprzedzone debatą ani zadawaniem pytań. Możemy przystąpić, tak? Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem dotyczącym informacji o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy. Kto z państwa posłów jest za uzupełnieniem porządku dziennego o punkt: Informacja Rady Ministrów na temat społecznych skutków wprowadzenia w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy instytucji, które wcześniej wymieniłem, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek odrzucił. Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem dotyczącym informacji w sprawie wypadku samochodowego w Oświęcimiu. Kto z państwa posłów jest za uzupełnieniem porządku dziennego o punkt obejmujący przedstawienie tej informacji, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił. Powracamy do rozpatrzenia punktu 1. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim. Proszę pana posła Michała Jacha o przedstawienie tego sprawozdania. Szanowny Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Połączone komisje: Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w dniu 4 lipca br. rozpatrywały zgłoszone w drugim czytaniu poprawki do ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim. Komisje rekomendują przyjąć poprawkę nr 1 i odrzucić poprawkę nr 2. Wysoki Sejm raczy przyjąć ustawę. Dziękuję panu posłowi. Przypominam, że chodzi o projekt ustawy z druku nr 2666. Przypominam, że komisje wnoszą o uchwalenie tego projektu. W dodatkowym sprawozdaniu komisje przedstawiają również poprawki, nad którymi głosować będziemy w pierwszej kolejności. Komisje wnoszą o przyjęcie tej poprawki. Głosujemy. Kto z państwa posłów jest za przyjęciem 1. poprawki, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę przyjął. Pytanie zadaje poseł Marek Hok, klub Platforma Obywatelska. Wysoka Izbo! Jeżeli tak naprawdę jest doskonała sytuacja finansowa budżetu państwa, o której się mówi, że jest najlepsza od 30 lat, jeżeli w takim razie stać nas na wiele rzeczy, to mam prośbę do posłów z Prawa i Sprawiedliwości, a zwłaszcza do parlamentarzystów z województwa zachodniopomorskiego, do panów ministrów Brudzińskiego i Szefernakera, aby pomogli mieszkańcom Drawska Pomorskiego i Złocieńca, pomogli tym biednym gminom, które biorą na siebie odpowiedzialność. Serce nie wystarczy, panie ministrze. Słuchacie suwerena, słuchacie Polaków, to słuchajcie mieszkańców biednych gmin, które biorą na siebie odpowiedzialność, łącząc gminy, biorą tę całą spuściznę po Ostrowicach.

Panie Pośle! Byłem przekonany, że pan nie wyjdzie z tym pytaniem, bo trzeba być wyjątkowym hipokrytą. żeby zadawać tego typu pytania. Przypomnę, że pierwszy wniosek wojewody zachodniopomorskiego o wyznaczenie zarządu komisarycznego w upadającej gminie był w 2010 r., kolejny - w 2015 r. W tym czasie rządziliście Polską. Uwaga, bo może nie wszyscy państwo wiedzą. Wójt, który dopuścił do 50-milionowego zadłużenia.

premiera i tego zarządu nie wyznaczyliście.

które się dobrowolnie łączą.

Proszę państwa, nie było pytania. Było wystąpienie posła Hoka. A minister jako przedstawiciel rządu zgodnie z art. 186. Sprostowanie, przypominam państwu.

Kto z państwa posłów jest za przyjęciem 2. poprawki, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił.

Wysoka Izbo! Chciałbym przypomnieć panu ministrowi Szefernakerowi, zapytać go o coś.

Wysoka Izbo! Gdyby szybciej się zabrali do tej pracy, na pewno tego długu by nie było. To jest jedna sprawa. Obiecaliście, że uratujecie gminę Ostrowice. Dzisiaj mówimy o drobnej sumie 1300 tys., żeby można było wyegzekwować środki na funkcjonowanie tych biednych gmin. O głos prosi wiceminister spraw wewnętrznych Paweł Szefernaker. Szanowni Państwo! Chętnie odpowiem na to pytanie. Ten dług, o którym pan mówi, był zaciągnięty za wójta z Platformy Obywatelskiej, który zaciągał te zobowiązania w parabankach. One lawinowo rosły przez ostanie 2 lata. A komisarz rządowy.

I uwaga: komisarze nie podejmowali zobowiązań w parabankach, tak jak za Platformy Obywatelskiej. Kto z państwa posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 2666, wraz z przyjętą poprawką, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Powracamy do rozpatrzenia punktu 2. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Przystępujemy do trzeciego czytania. Proszę pana posła Wiesława Krajewskiego o przedstawienie tego sprawozdania.

Wysoka Izbo! W imieniu Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa przedstawiam dodatkowe sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, druk nr 2377.

Komisja wnioskuje o odrzucenie poprawek 2. i 3. Komisja rekomenduje przyjęcie projektu ustawy w całości. Dziękuję panu posłowi. Przypominam, chodzi o druk nr 2537. Nad poprawkami, które komisja przedstawia w dodatkowym sprawozdaniu, głosujemy w pierwszej kolejności. Poprawki od 1. do 4. zostały zgłoszone do art. 1 projektu ustawy nowelizującej zawierającego zmiany do ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Nad nimi głosować będziemy łącznie. Komisja wnosi o ich przyjęcie. Pytanie zadaje poseł Paweł Bańkowski, klub Platforma Obywatelska. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Czy prawdą jest, że węgiel brunatny, który jest jakościowo dużo gorszy niż węgiel kamienny i charakteryzuje się pięciokrotnie wyższą emisją pyłu podczas spalania, siedmiokrotnie wyższą emisją węglowodorów aromatycznych i trzykrotnie wyższą emisją benzopirenu, do czasu złożenia tych poprawek przez klub PiS był wykluczony jako paliwo przeznaczone do spalania w sektorze komunalno-bytowym? Czy prawdą jest, jak uzasadniał pan minister Tobiszowski, że ta poprawka, te poprawki zostały złożone i przygotowane pod Kopalnię Węgla Brunatnego Sieniawa? Czy Skarb Państwa ma udziały w tej kopalni? Czy ministerstwo oszacowało, jaki wolumen węgla brunatnego będzie spalany w gospodarstwach domowych na podstawie tych poprawek do 1 czerwca 2020 r. Jak zapisy tej ustawy, które pozwalają dzięki tym poprawkom spalać węgiel brunatny w gospodarstwach domowych, będą się miały do przyjętych uchwał antysmogowych zakazujących spalania tego węgla przez dużą część sejmików wojewódzkich?

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawki przyjął. W 2. poprawce do art. 3a ust. 2 wnioskodawcy proponują, aby określenie wymagań, o jakich mowa w tym przepisie, następowało w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw energii w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Jej przyjęcie spowoduje bezprzedmiotowość poprawki 3. Pytanie zadaje poseł Marek Sowa, klub Nowoczesna. To jest bardzo ważna poprawka. Trudno sobie wyobrazić, aby przy częstych sporach ministra energii z ministrem środowiska, który odpowiada za czyste powietrze zgodnie z ustawą o działach, takie rozporządzenie wydawał jedynie minister energii. Dlatego bardzo państwa proszę, abyście przyjęli tę poprawkę, którą zgłosiliśmy, tak by to rozporządzenie zostało wydane w porozumieniu z ministrem środowiska i z ministrem właściwym do spraw gospodarki. Zresztą uważam, że to jest kluczowy element i że to jest też odpowiedź na oczekiwanie środowisk, które bardzo wiele zrobiły na rzecz zmian legislacyjnych, również wprowadzenia regulacji dotyczących jakości paliw. Pan minister Grzegorz Tobiszowski odpowie na to pytanie. Panie i Panowie Posłowie!

Dlatego że w art. 3a ust. 2a mamy zapis, że minister właściwy do spraw energii w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska i ministrem właściwym do spraw gospodarki co najmniej raz na 2 lata dokonuje przeglądu wymagań jakościowych określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 2 w celu oceny wpływu ich stosowania na ochronę środowiska, zdrowie ludzi oraz interesy konsumentów i że wyniki tego przeglądu stanowią podstawę do zmiany tych wymagań. A więc mamy to ujęte w naszej ustawie, stąd proponujemy, aby tych poprawek nie przyjmować. Proszę bardzo. Panie ministrze, z pełnym szacunkiem, pan doskonale przytoczył przepis o tym, jak będziecie dokonywali oceny. Skoro to robicie w porozumieniu z ministrem środowiska i z ministrem właściwym do spraw gospodarki, to dlaczego nie chcecie wspólnie podjąć pracy nad rozporządzeniem?

Kto z państwa posłów jest za przyjęciem 2. poprawki, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Ale zgodnie z regulaminem, panie pośle. Regulamin mówi, że marszałek najpierw zapozna się z wnioskiem na piśmie, a potem. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Yaakov Nagel, jeden z doradców premiera Benjamina Netanjahu, powiedział, że rząd polski wycofał się z zapisów ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej z podkulonym ogonem. Zmieniliśmy prawo, nie dając im nic w zamian - powiedział Nagel w „The Times of Israel” Okazuje się, Wysoka Izbo, że wstawanie z kolan kończy się podkuleniem ogona. Ten anons świadczy o tym, że Polska doznała ogromnego upokorzenia na arenie międzynarodowej, ale także w oczach wszystkich rodaków.

Jest to wniosek formalny o przerwę, więc poddam ten wniosek pod głosowanie. Kto z państwa jest za zarządzeniem przerwy w obradach, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

W 3. poprawce do art. 3a ust. 2 wnioskodawcy proponują, aby określenie wymagań, o jakich mowa w tym przepisie, następowało w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw energii w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska. Kto z państwa jest za przyjęciem poprawki 3., proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił.

Wysoka Izbo! Panie Ministrze!

Ceny ogrzewania wzrosną. Tymczasem zalewa nas węgiel z importu. Mam pytanie, panie ministrze, jakie propozycje ma rząd Prawa i Sprawiedliwości dla 5,5 mln gospodarstw domowych, żeby zrekompensować wzrost kosztów ogrzewania i zminimalizować ubóstwo energetyczne, które wzrasta w naszym kraju. Minister Grzegorz Tobiszowski odpowie na pytanie. Panie i Panowie Posłowie! Chcę tylko przypomnieć, że już decyzje sześciu marszałków poszczególnych województw w tamtym roku wyprzedziły nasze decyzje zawarte w ustawie o jakości paliw, co spowodowało, że proces podwyżki cen rozpoczął się w zeszłym roku.

Kto z państwa posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy z druku nr 2537, wraz z przyjętymi poprawkami, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Powracamy do rozpatrzenia punktu 3. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw. Trzecie czytanie. Proszę pana posła Wojciecha Murdzka o przedstawienie tego sprawozdania. Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić dodatkowe sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw, druk nr 2549.

Dziękuję bardzo. Dziękuję.

Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Kto z państwa jest za przyjęciem 1. poprawki, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę odrzucił. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Kto z państwa jest za przyjęciem 2. poprawki, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Za głosowało 419, 1 - przeciw, 1 wstrzymał się. Sejm poprawki przyjął. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z państwa jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 2612, wraz z przyjętymi poprawkami, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Powracamy do rozpatrzenia punktu 4. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz Komisji Obrony Narodowej o rządowym projekcie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 2659-A. Trzecie czytanie. Proszę pana posła Tadeusza Dziubę o przedstawienie tego sprawozdania. Szanowni Państwo! Sejmowe Komisje: Obrony Narodowej oraz Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii rekomendują przyjęcie projektu ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa wraz z dwiema poprawkami, a mianowicie z poprawkami 10. i 11. Komisje rekomendują odrzucenie pozostałych dziesięciu poprawek, tak jak to wyszczególniono w druku nr 2659-A.

Komisje wnoszą, przypominam, o odrzucenie tej poprawki. Kto z państwa jest za przyjęciem 1. poprawki, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę odrzucił. Komisje wnoszą o odrzucenie tej poprawki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Komisje wnoszą o odrzucenie tej poprawki. Pytanie zadaje poseł Paweł Pudłowski, klub Nowoczesna. Ponieważ domyślam się, że macie państwo nakaz głosowania przeciwko tej poprawce, chciałbym zapytać, czy ją dobrze rozumiecie. W naszej poprawce sugerujemy, aby zamiast powoływania pełnomocnika, który to pełnomocnik będzie reprezentantem pana premiera i będzie koordynował działania pomiędzy Ministerstwem Cyfryzacji, Ministerstwem Obrony Narodowej i MSWiA, dać tę prerogatywę ministrowi właściwemu do spraw cyfryzacji, do spraw informatyzacji kraju. Uważamy, że te kompetencje w tym ministerstwie są i to właśnie ta osoba powinna wypełniać te zadania koordynacji. Po co powoływać dodatkową osobę, która będzie dodatkowym elementem w tym głuchym telefonie? Są sytuacje, w których być może powołanie pełnomocników jest wskazane. Nie może jedna osoba być jednocześnie prezydentem i premierem. Dziękuję. Kto z państwa jest za przyjęciem 3. poprawki, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Głosujemy. Kto z państwa jest za przyjęciem 4. poprawki, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Kto z państwa jest za przyjęciem 5. poprawki, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę odrzucił. Komisje wnoszą o jej odrzucenie. Pytanie zadaje poseł Piotr Cieśliński, klub Platforma Obywatelska. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Nie ma wątpliwości, że odpowiedzialność za cyberbezpieczeństwo spoczywa na barkach państwa, a to dlatego że jest to jego obowiązek wobec suwerena rzecz jasna. Jednym z elementów podniesienia poziomu tego bezpieczeństwa jest szeroko rozumiana edukacja społeczeństwa w tym właśnie zakresie.

Chcę wyraźnie podkreślić, że mówimy tutaj o uprawnieniach, a nie o obowiązkach, ale chociażby w takim zakresie państwo powinno wziąć na siebie odpowiedzialność za tak ważny obszar z punktu widzenia realizacji celów projektu. Dziękuję. Kto z państwa jest za przyjęciem 6. poprawki, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Komisje wnoszą o odrzucenie tej poprawki. Kto z państwa jest za przyjęciem 7. poprawki, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę odrzucił. W 8. poprawce do art. 55 wnioskodawcy proponują m.in. nowe brzmienie wprowadzenia do wyliczenia. Komisje wnoszą o odrzucenie tej poprawki. Pytanie zadaje poseł Piotr Cieśliński, klub Platforma Obywatelska. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Czy nie jest to furtka dla takich działań jak w 2015 r., kiedy to na polecenie pana ministra Macierewicza niejaki Bartłomiej Misiewicz za pomocą dorobionego klucza, bez żadnych prawnych umocowań włamał się czy, jak kto woli, wszedł zwyczajnie z buta do pomieszczeń centrum kontrwywiadu NATO? Jeżeli odrzucacie poprawkę obligującą osobę kontrolującą do posiadania przepustki, to pozbawiacie podmiot kontrolowany, kontrolujący jakiegokolwiek wpływu na to, co będzie się działo z tą osobą w trakcie kontroli. Kto zatem weźmie odpowiedzialność za nieprzeszkoloną stanowiskowo osobę kontrolującą np. elektrownię lub petrochemię, gdzie nieznajomość zasad bezpieczeństwa obowiązujących w obiekcie [[Dzwonek]] może prowadzić do utraty zdrowia. Kto z państwa jest za przyjęciem 8. poprawki, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Komisje wnoszą o jej odrzucenie. Pytanie zadaje poseł Arkadiusz Marchewka, klub Platforma Obywatelska. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Skoro rozmawiamy o ustawie, która ma poprawić bezpieczeństwo w sieci, to warto zapytać, czy ktoś przypadkiem nie zhakował strony ministerstwa. Bo w projekcie ustawy jest zapisane, że musi powstać strategia cyberbezpieczeństwa i powstanie ona najpóźniej za 1,5 roku. To ta strategia jest, czy jej nie ma? W jakim celu chcecie przyjmować kolejne strategie, jeśli dopiero co premier Szydło podpisała uchwałę o przyjęciu strategii cyberbezpieczeństwa? Czy ta strategia jest, czy jej nie ma? Pytanie zgłasza poseł Paweł Pudłowski, klub Nowoczesna. Zanim pan minister, bo widzę, że już się czai do odpowiedzi, powie nam, że ta strategia to tak naprawdę są „Krajowe ramy polityki cyberbezpieczeństwa”, chciałem zwrócić państwa uwagę na to, że ta poprawka, którą zgłaszamy, jest bardzo łatwa. Dajemy wam pół roku na przygotowanie strategii dotyczącej cyberbezpieczeństwa, zamiast, jak państwo wnioskujecie, 1,5 roku. NIK raportował: Działania prowadzone są bez przygotowania i bez wspólnej wizji. Instytucje w zasadzie ze sobą nie rozmawiają. Państwo potrzebowaliście 3 lat, żeby złożyć ustawę, w której proponujecie, że za 1,5 roku zrobicie strategię ds. cyberzagrożeń. Wszystko jest dobrze, dopóki komputery pracują, dopóki nie ma, tak jak 2 miesiące temu, wielkiej awarii ePUAP-u, gdy nie można w zasadzie w ogóle skorzystać z e-administracji.

Proszę. Panie Marszałku!

Ten dokument ma inną nazwę, ale to ze względów proceduralnych, a nie żadnych innych, natomiast jest jasne, że musimy go co jakiś czas aktualizować i będziemy to robić. Data wyznaczona na przyszły rok ma umożliwić nam m.in. zebranie doświadczeń z wdrożenia tej dyrektywy NIS i implementacji w Polsce, żeby nie wydawać niepotrzebnie pieniędzy i nie tworzyć pustych dokumentów. Dziękuję. Kto z państwa jest za przyjęciem 9. poprawki, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę odrzucił. Komisje wnoszą o przyjęcie tej poprawki. Kto z państwa jest za przyjęciem 10. poprawki, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę przyjął. Komisje wnoszą o przyjęcie tej poprawki. Pytanie zadaje poseł Paweł Pudłowski, klub Nowoczesna. Wysoka Izbo! Co prawda chciałem się wypowiedzieć przy tej poprzedniej poprawce, ale tak naprawdę to komentarz, pytanie dotyczące tych poprawek jest takie samo. Czy nie uważacie państwo, że za mało środków jest przeznaczane na cyberbezpieczeństwo? Już w październiku 2016 r. ówczesna minister stwierdziła na spotkaniu publicznym, oficjalnym, otwartym, że podległy jej resort nie dysponuje ekspertami, wiedzą ani środkami finansowymi na skuteczne wdrażanie strategii bezpieczeństwa w naszym kraju.

To naprawdę nie jest dużo na przygotowanie i zrealizowanie właściwych działań w zakresie cyberbezpieczeństwa. Proszę. Kto z państwa jest za przyjęciem 11. poprawki, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę przyjął. Komisje wnoszą o odrzucenie tej poprawki. Pytanie zadaje poseł Paweł Suski, klub Platforma Obywatelska. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Jest to obrót bezgotówkowy, który jest najbardziej narażony na cyberataki. Krajowy system bezpieczeństwa, który dziś rząd chce przygotować, nie obejmuje ochroną transakcji bezgotówkowych. Dlaczego nie chcecie ochronić pieniędzy Polaków? Incydentów dotyczących naruszeń właśnie bezpieczeństwa transakcji bezgotówkowych jest najwięcej. Ta poprawka właśnie reguluje tę kwestię. Pan minister odpowiada, że KNF albo banki sobie z tym poradzą. Zintegrowany powinien również chronić pieniądze Polaków.

Panie Marszałku!

Jeśli chodzi o obszar usług płatniczych, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby również te usługi po tym, jak zostaną zgłoszone do KNF-u, były również zgłoszone później dalej do CSIRT-ów. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę odrzucił.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Projekt tej ustawy powstawał w chaosie i w atmosferze konfliktu pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej i Ministerstwem Cyfryzacji. Niestety chyba taki chaos po wprowadzeniu pozostanie. Przytoczę tylko kilka wątpliwości, które pojawiały się w konsultacjach społecznych i dotyczyły takich spraw jak: brak precyzyjnych zasad funkcjonowania jednostek zależnych od organów państwowych, brak ograniczenia zakresu uprawnień nadzorczych organów nadzoru i kontroli, brak publikacji kluczowych aktów wykonawczych, brak jednego punktu zgłoszeń incydentów na poziomie krajowym itd. Cyfrowe państwo musi być bezpieczne, ale bezpieczeństwa w sieci nie zagwarantuje się tylko na papierze. Na koniec tamtego roku, kiedy był przygotowywany budżet na 2018 r., Ministerstwo Cyfryzacji zawnioskowało o 76 mln zł na realizację strategii cyberbezpieczeństwa. Dostało ile? 0 zł. W jaki sposób w takim razie będą przez ministerstwo realizowane te [[Dzwonek]] działania, skoro nie ma na to pieniędzy w budżecie? Głos ma poseł Paweł Pudłowski, klub Nowoczesna. Wysoka Izbo! Ustawa, nad którą głosujemy, jest bardzo ważna i problem, który omawiamy, jest bardzo ważny. W światowym indeksie cyberbezpieczeństwa Polska zajmuje 40. miejsce. Są tam brane pod uwagę podstawy prawne, zdolność operacyjna, środki organizacyjne, czyli polityki i procedury, kwalifikacje, czyli czy są standardy, czy mamy kadrę, która może to realizować, i współpraca międzynarodowa z innymi. 40. miejsce - za takimi krajami jak Stany Zjednoczone, Singapur, Wielka Brytania, Francja, Kanada czy Rosja. Być może to nie dziwi, ale przed nami jest również Grecja, Estonia, Egipt, a nawet Mauritius. Nie możemy odpowiedzialnie poprzeć państwa ustawy. Uważamy, że jest za mało ambitna, że za małe nadaje tempo i za mało środków dedykowanych jest na obronę cyberbezpieczeństwa. NIK swój raport kończy tym, że właśnie za mało środków jest na to dedykowane. Tak że z przykrością muszę stwierdzić, że pomimo że w tej ustawie jest kilka elementów właściwych, będziemy głosowali przeciw. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z państwa posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy z druku nr 2659, wraz z przyjętymi poprawkami, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Powracamy do rozpatrzenia punktu 5. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 2547. Kto z państwa jest za przyjęciem w całości projektu z druku nr 2547, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Powracamy do rozpatrzenia punktu 6. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 2588. Pytanie zadaje poseł Sławomir Neumann, klub Platforma Obywatelska. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Głosujemy nad projektem ustawy, która pozwala, żeby ze środków Funduszu Rezerwy Demograficznej inwestować nie tylko w obligacje bezpieczne, czyli obligacje Skarbu Państwa, ale także obligacje różnych prywatnych firm. Wasze ekscesy, waszych urzędników czy waszych partyjnych nominatów, którzy zachęcali w bankach państwowych do inwestowania w GetBack i ich obligacje. Do dzisiaj nie chcecie tego wyjaśnić. I po aferze SKOK, kiedy kilka miliardów złotych także było straconych - w tym przypadku zapłacił Bankowy Fundusz Gwarancyjny - nie możemy się zgodzić na to, żeby tacy eksperci od finansów, od inwestycji, jak wasi ludzie ze SKOK-ów czy z GetBack zajmowali się funduszami emerytów z Funduszu Rezerwy Demograficznej. Głosujemy. Kto z państwa posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy z druku nr 2588, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 431 posłów. Powracamy do rozpatrzenia punktu 7. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

Dziękuję bardzo. Wysoka Izbo! W drugim czytaniu do projektu zawartego w druku nr 2661 złożono 27 poprawek.

Wysoka Izbo!

Komisja poparła te poprawki, które umacniają uszczelnienie przepisów, a nie poparła tych poprawek, które rozszczelniają przepisy.

Komisja wnosi o jej odrzucenie. Kto z państwa jest za przyjęciem 1. poprawki, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Nad nimi głosować będziemy łącznie. Komisja wnosi o ich przyjęcie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawki przyjął. Komisja wnosi o jej przyjęcie. Kto z państwa jest za przyjęciem 3. poprawki, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Komisja wnosi o jej odrzucenie. Kto z państwa jest za przyjęciem 4. poprawki, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę odrzucił.

Komisja wnosi o jej odrzucenie. Kto z państwa jest za przyjęciem 5. poprawki, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Sejm poprawkę odrzucił. Nad nimi głosować będziemy łącznie. Komisja wnosi o ich odrzucenie.

Wysoka Izbo! Miałem nie zadawać pytania, a właściwie nie wyjaśniać tego państwu posłom tu obecnym, ze względu na to, że ta poprawka jest w pewnym sensie skonsumowana przez kolejną poprawkę, zaproponowaną przez Prawo i Sprawiedliwość, w której jest pewna zmiana, mianowicie wprowadzona jest pewna sankcja. Natomiast muszę to zrobić, muszę wyjaśnić pewną rzecz ze względu na to, że pani sprawozdawca mija się z prawdą. My proponujemy poprawki, które nie rozszczelniają systemu związanego z gospodarką odpadami. To jest nieprawda. Nasza poprawka była właśnie po to, żeby ten system uszczelnić, a jednocześnie umożliwić działalność gospodarczą w ramach gospodarki odpadami. Proszę bardzo. Kto z państwa posłów jest za przyjęciem poprawek 6. i 8., proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawki odrzucił.

Nad nimi głosować będziemy łącznie. Ich przyjęcie spowoduje bezprzedmiotowość poprawki 24. Komisja wnosi o ich przyjęcie. Kto z państwa jest za przyjęciem poprawek 7., 10. i 25., proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawki przyjął.

Komisja wnosi o jej przyjęcie. Kto z państwa jest za przyjęciem 9. poprawki, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę przyjął.

Konsekwencją przyjęcia poprawki będzie zastąpienie w projekcie ustawy występującego w różnych przypadkach wyrazu „udziałowiec” wyrazem „prokurent”

Komisja wnosi o jej odrzucenie. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Niestety PiS przez swoją niekompetencję sparaliżuje zapisami w tej ustawie inwestycje przede wszystkim na autostradach i liniach kolejowych, bo nie wie o tym, jaka jest rzeczywista definicja odpadu w Polsce, że odpad to także ziemia z wykopów, a przekształcanie odpadu to jest konstruowanie nasypów i wymaga w kraju, w którym 70% powierzchni nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, takich planów albo warunków zabudowy, podczas gdy w przypadku tych inwestycji infrastrukturalnych są specustawy i nie ma takiego wymogu. I tylko dlatego, że PiS upiera się ideologicznie i partyjnie, żeby odrzucać wszelkie poprawki opozycji, nawet jeśli są sensowne i logiczne, tylko dlatego ta poprawka jest odrzucona.

Dziękuję. Kto z państwa jest za przyjęciem poprawki 12., proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto z państwa jest za przyjęciem 13. poprawki, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę przyjął. Komisja wnosi o jej odrzucenie. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ta poprawka z naszej strony zmierza do doprecyzowania i zobowiązania ministra środowiska, by bardzo wysoko wyszacowane zabezpieczenia były zgodne z ich celem i odpowiadały nie tylko wartości odpadów, ale także przede wszystkim skutkom, jakie może wywołać ich porzucenie, np. będą bardzo drogie zabezpieczenia na odpady, których nikt w życiu nie porzuci, bo to są metale nieżelazne, i to sparaliżuje tego typu rozwiązanie. To jest na zasadzie: każda propozycja logiczna jest odrzucana, bo my mamy rację, bo po nas tylko potop.

Kto z państwa jest za przyjęciem 14. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Kto z państwa jest za przyjęciem 15. poprawki, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę przyjął.

Komisja wnosi o jej odrzucenie. Kto z państwa jest za przyjęciem 16. poprawki, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę odrzucił. Komisja wnosi o jej odrzucenie. Pytanie zadaje poseł Dariusz Piontkowski, klub Prawo i Sprawiedliwość. Pytanie do ministra. Z jednej strony totalna opozycja mówi o tym, że Polska stała się śmietnikiem Europy. czyli ściągamy za dużo odpadów, a z drugiej strony jednocześnie próbuje doprowadzić do tego, aby cena za przywóz odpadów była zdecydowanie niższa niż w innych krajach europejskich, aby można było spokojnie sprowadzać wszelkiego rodzaju odpady, jakie tylko sobie można zażyczyć.

To wyraźnie pokazuje, w którą stronę tak naprawdę totalna opozycja próbuje iść.

Proszę. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Otóż w tej poprawce posłowie Platformy Obywatelskiej proponują obniżenie proponowanej przez nas kwoty opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia na import odpadów.

Uważam, że zmniejszanie proponowane przez Platformę jest całkowicie nieuzasadnione, dlatego że bylibyśmy niemalże konkurencyjni do przywożenia odpadów, gdyż stawka takiej opłaty w Niemczech wynosi do 6 tys. euro, a więc i tak 14 tys. zł proponowane przez nas to znacznie mniej, a zmniejszenie tego do kwoty z propozycji Platformy byłoby wręcz zachętą, żeby to do nas sprowadzać te odpady. Głosujemy. Kto z państwa jest za przyjęciem 17. poprawki, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę odrzucił. W 18. poprawce do ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów wnioskodawcy proponują zachować dotychczasowe brzmienie art. 11. Komisja wnosi o jej odrzucenie. Pytanie zadaje poseł Gabriela Lenartowicz, klub Platforma Obywatelska. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Trochę mnie to dziwi, że najpierw przez 2 lata wyrażacie zgody na import odpadów niebezpiecznych, na dwukrotnie wyższą masę odpadów, a teraz nagle - szlaban, nawet jak to ma uzasadnienie, jeśli chodzi o utylizację polskich odpadów. Te liczby, które przytacza poseł Piontkowski, to jest manipulacja, bo ta większa ilość importowanych odpadów pochodziła z czasów, kiedy nie było zielonej listy i trzeba było wydawać zgody. W tej chwili od ubiegłego roku te odpady nie wymagają wydania zezwolenia. Po prostu kłamiecie i uciekacie od odpowiedzialności. Jeśli uważacie, że import odpadów niebezpiecznych jest zbyt duży, to decyzje wydaje Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, który wam podlega. Wy po prostu nie chcecie [[Dzwonek]] brać odpowiedzialności i uważacie, że sami. Proszę bardzo. Panie ministrze, w związku z tym pytanie: Czy prawdą jest to, co padło przed chwilą z mównicy, że w ubiegłym roku sprowadzono do Polski więcej odpadów niż 7 czy 8 lat temu? Czy prawdą jest, że Polska, sprowadzając w ubiegłym roku 370 tys. t odpadów, w poprzednich latach zaledwie sto kilkadziesiąt tysięcy ton, sprowadzała tych odpadów zdecydowanie mniej niż nasi sąsiedzi?

Minister Henryk Kowalczyk odpowie na to pytanie. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Trudno dyskutować z liczbami.

A więc jeśli to jest zwiększenie, 377 tys. jest większe od 1600 tys., to naprawdę trudno dyskutować tu o innych faktach.

Dziękuję. Kto z państwa jest za przyjęciem 18. poprawki, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Sejm poprawkę odrzucił. W 19. poprawce do ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów wnioskodawcy proponują nadać nowe brzmienie art. 11b. Pytanie zadaje poseł Tomasz Szymański, klub Platforma Obywatelska.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Tą ustawą na pewno nie ograniczycie fali pożarów, bo, po pierwsze, nie wiecie co i dlaczego się paliło. Dlaczego traktujecie polskich przedsiębiorców po macoszemu? Dlaczego daliście im tylko 5 dni, a odliczając sobotę i niedzielę, de facto 3 dni na skonsultowanie tego projektu ustawy?

Po drugie, firmy recyklingowe, przetwarzające odpady. Właśnie, mówicie o odpadach. To jest surowiec, który jest niezbędny do dalszej produkcji. Dzięki tym właśnie surowcom możemy taniej uzyskiwać produkty dzięki temu, że emisja dwutlenku węgla, ale także energia, która jest niezwykle cenna. W tym momencie są realne oszczędności. Dziękuję panu posłowi.

Kto z państwa jest za przyjęciem 19. poprawki, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę odrzucił. Kto z państwa jest za przyjęciem 20. poprawki, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę przyjął. Komisja wnosi o jej odrzucenie. Jej przyjęcie spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 22. Pytanie zadaje poseł Dariusz Piontkowski, klub Prawo i Sprawiedliwość. Panie Ministrze! Ta poprawka ma doprowadzić do tego, aby dotychczasowe przepisy, które nie potrafiły doprowadzić do tego, aby gospodarka odpadami w Polsce była zgodna z oczekiwaniami obywateli, tzn. aby nie szkodziła środowisku i była korzystna dla zdrowia i życia ludzi. Ta poprawka ma doprowadzić teraz do tego, abyśmy przez kolejne 3 lata utrzymali przepisy, które pozwalały na funkcjonowanie, jak to określił jeden z wiceministrów, tzw. mafii śmieciowej.

Dziękuję. Kto z państwa jest za przyjęciem 21. poprawki, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Sejm poprawkę odrzucił. Komisja wnosi o jej przyjęcie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę przyjął.

Komisja wnosi o jej odrzucenie.

Sejm poprawkę odrzucił.

Kto jest przeciw?

Całość projektu ustawy. Pytanie zadaje poseł Gabriela Lenartowicz, klub Platforma Obywatelska. Panie Marszałku! Skrajną nieodpowiedzialnością jest nieznajomość tematu i formułowanie przepisów tak, że one są wbrew temu, jaki jest cel tej ustawy. Tak naprawdę szykanujecie uczciwych polskich przedsiębiorców, a wzmocnicie mafię, bo rozszerzycie szarą strefę. Niestety ten resort to jest narodowa katastrofa ekologiczna. Do czego się nie zabierzecie, to jest dramat. Najpierw puszcza, potem wycinacie drzewa, zabijane są foki, a teraz mamy gwałtownie rosnącą liczbę pożarów i manipulacje faktami, [[Poruszenie na sali]] bo fakty, które pan przytacza, dotyczą czasów, kiedy nie potrzeba było wykazu, nie potrzeba było zezwoleń.

Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo Ministrowie! Ochrona środowiska i ochrona powietrza, którym oddychamy, jest nadrzędna, panie pośle, jeżeli pan miał wątpliwości, że inaczej myślę, ale właśnie dlatego tę ustawę poprzemy, mimo że ona jest pełna drastycznych błędów i procedowano nad nią z lekceważeniem wielu stron, szczególnie uczciwych przedsiębiorców. Ale dajemy wam szansę, że poprawicie to w Senacie, tak jak obiecaliście.

Dziękuję. Głos ma poseł Dariusz Piontkowski, Prawo i Sprawiedliwość. Od kilku lat przedsiębiorcy, którzy legalnie działają w branży odpadowej, domagają się zmiany przepisów, tak aby wyrównać szanse między tymi, którzy działają w szarej strefie, a tymi, którzy próbują przestrzegać przepisów obowiązujących w Polsce. Ta ustawa wyraźnie wychodzi naprzeciw ich oczekiwaniom. W trakcie prac komisji wprowadziliśmy poprawki, które były realizacją postulatów środowisk, tak aby nie wylać dziecka z kąpielą. Pozwala również nie dopuścić do prowadzenia działalności gospodarczej przez tych, którzy już wcześniej złamali przepisy i są przestępcami, a na mocy kruczków prawnych potrafili tę działalność prowadzić dalej ze szkodą dla środowiska i obywateli. Ta ustawa wprowadza dodatkowe kary dla tych, którzy łamią przepisy, a więc działa na korzyść obywateli. Wysoka Izbo! Ja uważam, że w tej Izbie powinno się wypowiadać w sposób bardzo rzetelny, logiczny i racjonalny. Nawet jak poseł Tarczyński zajmuje się czym innym, to warto też mówić. Problem polega na tym, że chyba. Problem polega na tym, że przepisy wprowadzone na mocy tej ustawy nie są przepisami, które uniemożliwiałyby działalność gospodarczą. Nie ma czegoś takiego. Natomiast ważną rzeczą jest, żebyśmy sobie wyjaśnili, dlaczego doszło do takiego procederu palenia śmieci w Polsce, co było tego przyczyną - czy to były takie względy, że np. ktoś przekraczał prawo, czy też po prostu stworzone zostało specjalne prawo pozwalające na bezkarny import śmieci do Polski. Dlatego też mam pytanie do pana ministra środowiska. Po pierwsze, kiedy odpowiecie na moją interpelację w tej sprawie i na inne pytania dotyczące tego procederu?

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Na początku pragnę podziękować wszystkim klubom za konstruktywną współpracę przy pracach nad tą ustawą, chociaż ostatnie wypowiedzi przedstawiciela klubu Platformy Obywatelskiej nie świadczyły o tym, żeby była jakakolwiek konstruktywna praca. Ale w czasie prac komisji zdarzały się momenty konstruktywnej pracy. Ja wiem, że najlepiej, jakby zostało tak, jak było, żeby śmieci można było przywozić bez żadnej odpowiedzialności, bo tak niestety było do tej pory.

To jest pierwsza przyczyna i pożarów, i porzuceń, i kłopotów samorządów. Oczywiście zdarzało się to przez wiele, wiele lat. Szanowni Państwo! Przez te wszystkie lata nikomu nie przyszło do głowy, że system jest ułomny, że system jest nieszczelny, że system pozwala. My dyskutujemy też o jakichś zezwoleniach zagranicznych. System pozwalał na to, żeby obok zezwoleń, które rzeczywiście w tym momencie są nieistotne - te zgodnie z prawem zwiezione odpady w celu odzyskania surowców wtórnych są niegroźne. Natomiast pod płaszczykiem tych zezwoleń były sprowadzane odpady, niestety niebezpieczne, odpady komunalne, czyli te, których wszyscy chcieli się pozbyć. A więc w tym przypadku od tego czasu uszczelniamy system. Ta ustawa tego nie rozwiązuje, to jest oczywiste, ale przynajmniej zabezpiecza nas przed dalszym przywożeniem w sposób nieograniczony odpadów, przed porzucaniem odpadów. Zwracam się do pani poseł Lieder z Nowoczesnej. Skoro ta ustawa - a zamierzacie ją poprzeć, za co bardzo dziękuję - jest tak zła, fatalna i ma tyle błędów, to dlaczego klub Nowoczesna nie złożył ani jednej poprawki, żeby spróbować chociaż trochę naprawić tę ustawę? Skoro zamierzacie poprzeć ustawę, a krytykujecie zapisy szczegółowe, to trzeba było złożyć pewne poprawki.

dobro naszego środowiska będzie uwzględnione i ta ustawa zyska poparcie. Proszę. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z państwa posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy z druku nr 2676, wraz z przyjętymi poprawkami, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Powracamy do rozpatrzenia punktu 8. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw. Dodatkowe sprawozdanie to druk nr 2677-A. Proszę panią poseł Annę Paluch o przedstawienie tego sprawozdania. Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W trakcie drugiego czytania projektu ustawy zawartego w druku nr 2662 złożono 15 poprawek.

Wysoka Izbo! Generalnie komisja nie zgodziła się na poprawkę ustrojową, na ten pakiet poprawek prowadzących do tego, żeby służby inspekcyjne podlegające wojewodzie wyjąć z administracji zespolonej wojewody. Przypomnę, że funkcje wojewody jako zwierzchnika służb w zakresie zarządzania kryzysowego są komplementarne z kompetencjami inspekcji, i to był powód, dla którego się na to nie zgodziliśmy. Wysoka Izbo! A propos tych uwag, które padały, o jakoby skandalicznym trybie procedowania przypomnę, że do dwudziestego drugiego, wobec powszechnego oburzenia Polaków na płonące wysypiska, rząd przygotował szybko pakiet tych dwóch ustaw, nad którymi teraz procedujemy. Komisja pracowała nad nimi kilka dni i dopiero dzisiaj, czyli 5 lipca, nad nimi dyskutujemy, więc myślę, że jak na ustawy, które mają usunąć stan, który bulwersuje większość Polaków, to jest zupełnie przyzwoite, dobre tempo, umożliwiające dobrą pracę. Proszę. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy.

Nad nimi głosować będziemy łącznie. Komisja wnosi o ich odrzucenie. Pytanie zadaje poseł Bogusław Sonik, klub Platforma Obywatelska. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że ta nowelizacja powoduje, że Inspekcja Ochrony Środowiska będzie wyposażona w uprawnienia policyjno-prokuratorskie, dochodzeniowo-śledcze. Instytucja ta nie jest przygotowana do prowadzenia takich działań. Na dodatek jeszcze nie powinno się łączyć funkcji kontrolnych z funkcjami ścigania.

Głos ma poseł Dariusz Piontkowski, Prawo i Sprawiedliwość. Szanowni Państwo! Kilka minut temu przegłosowaliśmy ustawę, która zaostrza przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej. Po to jednak, aby sprawdzić, czy przedsiębiorca rzeczywiście właściwie wykonuje prawo, trudno nie stworzyć dla Inspekcji Ochrony Środowiska dodatkowych uprawnień, tak aby mogła na bieżąco kontrolować, co dzieje się w tych dużych magazynach czy składowiskach, gdzie przetwarzane są odpady. Ta poprawka ma doprowadzić do tego, żeby Inspekcja Ochrony Środowiska była instytucją taką jak dotychczas, tzn. bezradną, taką, która nie potrafi zaradzić patologiom, która nie potrafi udowodnić przedsiębiorcy, że łamał prawo, że nielegalnie sprowadzał odpady albo je po prostu podpalał. I dlatego inspekcja została wyposażona m.in. w możliwość monitorowania, choćby za pomocą dronów, tego, co dzieje się na terenie składowiska. Dotychczasowa praktyka pokazała również, że Policja czy prokuratura niestety nie są dobrze przygotowane do ścigania tego typu przestępstw.

Kto z państwa posłów jest za przyjęciem poprawek 1. i 15., proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawki odrzucił.

Pytanie zadaje poseł Bogusław Sonik, klub Platforma Obywatelska. Szanowni Państwo! 20 lat administracji Inspekcji Ochrony Środowiska przyniosło takie wnioski, że należy skończyć z podwójnym podporządkowaniem tej inspekcji i podporządkować ją całkowicie, w sposób pionowy, Ministerstwu Środowiska, gwarantując w ten sposób, że żadne lokalne lobby nie będą miały wpływu na działalność tej inspekcji, a na dodatek będzie ona skutecznym narzędziem do kontrolowania w całej Polsce.

Zresztą, panie ministrze, jest wprowadzona pewnego rodzaju zmiana, dlatego że wyjmuje się z obecnych wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska laboratoria, które obecnie będą podporządkowane ministerstwu ochrony środowiska. Dziękuję. Kto z państwa jest za przyjęciem wymienionych poprawek, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawki odrzucił. Kto z państwa jest za przyjęciem 5. poprawki, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę odrzucił. Kto z państwa jest za przyjęciem 6. poprawki, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę przyjął. Z nią łączy się poprawka 9. Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawki przyjął. Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki. Jej przyjęcie spowoduje bezprzedmiotowość poprawki 12. Pytanie zadaje poseł Gabriela Lenartowicz, klub Platforma Obywatelska. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ta poprawka wynika z niekompetencji i jest zwyczajnie niezgodna z prawem, ingeruje w uprawnienia samorządu i każe niezgodnie z prawem władać terenami, do których nie ma się tytułu prawnego.

Ale odrzucamy, były. Nawet jeśli w ramach komisji przyznaliście rację, to ideologicznie je odrzucacie i wkładacie nam w usta zupełnie inne kwestie.

Kto z państwa jest za przyjęciem 11. poprawki, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę przyjął.

Kto z państwa jest za przyjęciem 13. poprawki, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę przyjął.

Kto z państwa jest za przyjęciem 14. poprawki, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę odrzucił. Pytanie zadaje poseł Bogusław Sonik, klub Platforma Obywatelska.

Pytanie zadaje poseł Dariusz Piontkowski, Prawo i Sprawiedliwość. Panie Ministrze! Czy ta ustawa jest realizacją postulatów przedsiębiorców, aby stworzyć w Polsce skuteczną inspekcję ochrony środowiska, inspekcję, która będzie dobrze finansowana, będzie zatrudniała odpowiednią liczbę pracowników, tak aby móc kontrolować także tych, którzy w ogóle prowadzą działania niezgodne z prawem i gromadzą odpady, nie mając na to żadnych zezwoleń, i doprowadzić potem do tego, aby takie osoby skazano prawomocnymi wyrokami? Czy ta ustawa pozwoli inspektorom ochrony środowiska wykorzystać dodatkowe zapisy prawne, które były przewidziane w poprzedniej ustawie o odpadach? Czy ta ustawa pozwoli w końcu stworzyć w Polsce system stałego monitoringu powietrza, ale być może także w niedługiej perspektywie - wody, i laboratoriów, które będą miały certyfikaty na terenie całego kraju?

Dziękuję. Głos ma minister środowiska Henryk Kowalczyk.

Wysoka Izbo! Otóż odpowiadając na pytanie pana posła Sonika, powiem, iż ustawa była konsultowana z wojewódzkimi inspektorami ochrony środowiska. Tak więc nie jest prawdą, że nie była konsultowana.

Zwiększa również uprawnienia kontrolne z wykorzystaniem wielu narzędzi, m.in. wprowadza możliwość kontrolowania samochodów, której do tej pory nie było. A więc te narzędzia, które otrzymuje Inspekcja Ochrony Środowiska, pozwolą na wdrożenie ustawy o odpadach tak, aby te przepisy, bardziej rygorystyczne, szczelne, były rzeczywiście egzekwowane i dotrzymywane. Przystępujemy do głosowania na całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 2677, wraz z przyjętymi poprawkami, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw. Powracamy do rozpatrzenia punktu 15. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2017 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium. W dyskusji zgłoszono poprawkę do projektu uchwały. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 2656-A. Proszę pana posła Andrzeja Szlachtę o przedstawienie sprawozdania komisji. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Premierze!

Komisja Finansów Publicznych na posiedzeniu w dniu 5 lipca rozpatrzyła ten wniosek i w głosowaniu go odrzuciła. Wcześniej Komisja Finansów Publicznych rozpatrzyła wniosek zgłoszony przez panią poseł Izabelę Leszczynę dotyczący negatywnej oceny wykonania części 19 budżetu. Reasumując, Komisja Finansów Publicznych rekomenduje Wysokiej Izbie przyjęcie w całości komisyjnego projektu uchwały w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. oraz w sprawie udzielenia absolutorium dla Rady Ministrów. Komisja wnosi o uchwalenie projektu uchwały zawartego w sprawozdaniu w druku nr 2656. Komisja przedstawia również wnioski mniejszości, a także w dodatkowym sprawozdaniu poprawkę, nad którymi głosować będziemy w pierwszej kolejności. W 1. wniosku mniejszości oraz tożsamej poprawce wnioskodawcy proponują nadać nowe brzmienie projektowi uchwały. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Przyjęcie tego wniosku mniejszości i poprawki spowoduje bezprzedmiotowość pozostałych propozycji.

Panie i Panowie Posłowie! Mam do państwa pytanie: Czy leci z nami pilot? Nie ma pana premiera Morawieckiego, który był ministrem finansów w roku 2017. To lekceważenie Wysokiej Izby. Remontowaliśmy tylko stare uzbrojenie. Nie zakupiono żadnego śmigłowca, ale jest pięć samolotów dla władzy. Proszę Państwa! Zgadnijcie, ile wydano? Nie możemy poprzeć tego budżetu. Szanowni państwo, ponad 30 opinii opisowych, czyli negatywnych.

Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Pani Minister! Chciałam zapytać, gdzie na nadwyżka.

Ano pewnie dlatego, że Polska ma jeden z najgorszych wyników w Unii Europejskiej. 12 krajów Unii Europejskiej pokazało, że jak się chce, to można wypracować nadwyżkę.

A Polska?

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

W 2. wniosku mniejszości wnioskodawcy proponują dodać punkt dotyczący wykonania budżetu państwa w części 19. Do pytania zgłosił się pan poseł Michał Szczerba, klub Platformy Obywatelskiej. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Rozmawiamy o wykonaniu budżetu państwa na rok 2017, ale nie będę marnował naszego czasu, mojego czasu, żeby przypomnieć państwu, w jakich warunkach był uchwalany ten budżet 16 grudnia w sali kolumnowej. Te gorszące obrazki, to, jak prowadziliście to głosowanie, zostaną z wami na zawsze. Ale przejdę teraz do tego, co jest clou, co wyszło z raportu Najwyższej Izby Kontroli. Rok 2017 jest rokiem rekordowym. W roku 2017 dwunastokrotnie wzrosły wydatki na premie dla najważniejszych urzędników państwowych. Mamy to czarno na białym - w raporcie NIK-u.

Panie Marszałku! To prawda.

Ale tego było wam za mało. Na transport wydaliście ponad 2 mln więcej w KPRM-ie, chociaż samochody służbowe przejechały o 130 km mniej. Naprawdę to trzeba umieć. Koszty waszego transportu są siedmiokrotnie wyższe niż koszty używania taksówek w Warszawie.

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 2. wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał?

Wysoki Sejmie! który w okresie dobrej koniunktury nie zbudował żadnych buforów na gorsze czasy. Indianie już wiedzieli, że jak upolowali bizona latem, to połowę musieli zostawić na zimę. To dlatego 20 państw Unii Europejskiej miało w zeszłym roku deficyt niższy niż 1%, a 12 państw miało nadwyżkę. Tymczasem Polska?

Jak wy się nie wstydzicie i jak wy to w ogóle robicie? Po tym rządzie nie będzie już śladu, ale niestety zostawi Polskę bezbronną wobec wahań w gospodarce.

Wysoka Izbo!

A jak wyglądała polityka senioralna? Kilka złotych waloryzacji. nie poparliście projektu nawet jednorazowego wsparcia, leki za darmo to swoista atrapa. Czy były pieniądze?

gdzie piszecie nową historię dla Polaków.

Panie Marszałku! Pani Minister! Dobre zdanie, które charakteryzowałoby sytuację ubiegłego roku, jest takie: Zastali Polskę murowaną, a zostawili drewnianą. Tak naprawdę chciałam zapytać, gdzie ten plan Morawieckiego i kiedy zobaczymy pierwsze jego rezultaty. bo miało nastąpić ożywienie w inwestycjach, cały rok czekaliśmy, tymczasem na koniec roku wyszło, że mamy najniższą stopę inwestycji prywatnych od 15 lat. Do tego, że firmy już wstrzymują się od inwestowania, w zasadzie można powiedzieć, że przywykliśmy. Ale to, że mamy w I kwartale ujemną dynamikę inwestycji firm krajowych, to już jest naprawdę zadziwiające, bo to trzeba umieć.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ja mam tę bardzo komfortową sytuację, że nie muszę się wyzłośliwiać, nie muszę robić wielkiej polityki z czegoś, co jest matematyką. Dwa dodać dwa jest cztery. Jeżeli po stronie przychodów i dochodów Skarbu Państwa udało się zwiększyć te sumy - z czego się bardzo cieszymy - to należy dążyć do tego, aby dwa dodać dwa było cztery, inaczej mówiąc, aby się zmniejszało zadłużenie państwa. Zwiększyliśmy podatki, zwiększyliśmy daniny publiczne, natomiast nie zmniejszyliśmy wydatków. Wynik jest taki, że niestety nasze zadłużenie cały czas rośnie. Nasze dzieci i długi. Długi też. Nasze dzieci i wnuki będą spłacały ich coraz więcej.

Pytanie zadaje pan poseł Tadeusz Cymański, klub Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku! 21 lat jestem tutaj, jestem z parlamentem związany, ale nigdy. Mówię to dlatego, żeby podać pewien szczegół. W końcowej fazie tej znakomitej dyskusji, na obszarze opozycji nie było ani jednego. Nigdy. Był jeden, było dwóch, trzech, ale zawsze ktoś był. Ja wiem, że status materialny ucierpiał, ale żeby aż tak? Trzeba powiedzieć wyraźnie: Najwyższa Izba Kontroli z tego miejsca, ustami prezesa, rekomendowała Wysokiej Izbie przyjęcie sprawozdania. Jest to instytucja, która nie oszczędzała was, a myśmy z tego korzystali, a dzisiaj nie oszczędza nas i sprawozdania, pytania stawia twarde. To jest ostatnia instytucja, która ma ogromny szacunek. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu uchwały w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów w brzmieniu z druku nr 2656, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Powracamy do rozpatrzenia punktu 18. porządku dziennego: Przedstawiony przez prezesa Rady Ministrów dokument: „Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie przedstawionej informacji, który poddam pod głosowanie. Odrzucenie tego wniosku będzie oznaczało, że Sejm informację przyjął do wiadomości.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam pytanie do pana premiera i proszę o odpowiedź na piśmie. Dlaczego się dzieje tak, że w czasach koniunktury gospodarczej drugi rok z rzędu strefy, zamiast się rozwijać, się zwijają?

Czy to jest efekt tego, że wymieniliście prawie 100% managementu w strefach, czy też propagandy, którą pan premier uprawia, mówiąc: jedna strefa w całej Polsce?

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Trudno się nie zgodzić z panem posłem Cymańskim, że polityka PiS-u doprowadziła do sytuacji, kiedy ostatnią instytucją, do której mamy zaufanie, jest Najwyższa Izba Kontroli. Dziękujemy panu prezesowi Kwiatkowskiemu. bo miałem okazję wczoraj rano odprowadzić do pracy pierwszą prezes Sądu Najwyższego. Na koniec pytanie. Dlaczego państwo nie reagowaliście, kiedy okazywało się, że po raz pierwszy od początku nakłady w specjalnych strefach inwestycyjnych spadały?

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie informacji zawartej w druku nr 2591, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek o odrzucenie informacji odrzucił. Powracamy do rozpatrzenia punktu 19. porządku dziennego: Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2017 roku wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2017 roku oraz komisyjnym projektem uchwały. Sejm przeprowadził pierwsze czytanie i przystąpił do drugiego czytania projektu uchwały. Wobec propozycji przystąpienia do głosowania po doręczeniu paniom i panom posłom zestawienia zgłoszonych poprawek zgłoszono sprzeciw. Propozycję tę poddam zatem pod głosowanie. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem propozycji przystąpienia do głosowania po doręczeniu zestawienia zgłoszonych poprawek, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm propozycję przyjął. Zestawienie zgłoszonych poprawek zostało doręczone do druku nr 2643. W 1. poprawce wnioskodawcy proponują nadać nowe brzmienie projektowi uchwały. Pytanie zadaje pan poseł Artur Dunin, Platforma. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Czy to prawda, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wie o tym, że pan prezes Kurski żąda od Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego pieniędzy za puszczanie transmisji z paraolimpiady? Czy to prawda, że zamiast funkcji społecznych kasa, kasa, kasa dla Kurskiego? Pytanie zadaje poseł Witold Zembaczyński, klub Nowoczesna. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Konstytucyjnie w art. 213 mamy ujęte, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji musi stać na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji. Tymczasem interes publiczny pod waszym nadzorem w telewizji narodowej już dawno zbankrutował, a rozplenił się wyłącznie interes partyjny i ten wielki i nabrzmiały interes partyjny dynda sobie na tym ekranie i przysłania wszystkie obiektywne przekazy. Do tego rzetelność dziennikarska, obiektywizm w wydaniu np. „Wiadomości” to jest dosłownie biały kruk.

Pytanie zadaje pan poseł Krzysztof Paszyk, klub Polskiego Stronnictwa Ludowego. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Wczoraj byliśmy świadkami wypowiedzi pana premiera Morawieckiego w Brukseli, w Strasburgu w Parlamencie Europejskim, który dowodził, że dziennikarze nie mają jakichkolwiek ograniczeń w dostępie do mediów publicznych, opozycja nie ma żadnych ograniczeń w dostępie do mediów publicznych. To chciałem dzisiaj większość sejmową zapytać: Czy to oznacza, że w najbliższym czasie zaproszenie do mediów publicznych, do kontynuowania swojego programu otrzyma pan red. Tomasz Lis? Przystępujemy do głosowania. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. W 2. poprawce wnioskodawcy proponują nowe brzmienie treści uchwały. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 2. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały zawartym w sprawozdaniu komisji.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Otóż Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w sposób rażący nie zakwestionowała cenzorskich zapędów prezesa Telewizji Polskiej Jacka Kurskiego, który cenzurował wielokrotnie, ale najbardziej spektakularnym przekładem jest wyeliminowanie Julii Wyszyńskiej.

To jest po prostu skandaliczne, niedopuszczalne.

To jest niedopuszczalne.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Jak patrzę na was, to zawsze mi się przypomina takie zwierzątko z bajki Adama Mickiewicza: Już był w ogródku, już witał się z gąską. I tak było również w przypadku Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Co się działo i co się stało 11 grudnia 2017 r.

Co zrobiła ta sama rada. ten sam przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 10 stycznia? Tak działacie. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu uchwały w brzmieniu z druku nr 2643, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał?

Sejm podjął uchwałę w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2017 r. Powracamy do rozpatrzenia punktu 20. porządku dziennego: Informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2017 roku wraz z komisyjnym projektem uchwały. Sejm przeprowadził pierwsze czytanie i przystąpił do drugiego czytania projektu uchwały. Wobec propozycji przystąpienia do głosowania po doręczeniu paniom i panom posłom zestawienia zgłoszonych poprawek zgłoszono sprzeciw. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem propozycji przystąpienia do głosowania po doręczeniu zestawienia zgłoszonych poprawek, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał?

Sejm propozycję przyjął. Zestawienie zgłoszonych poprawek zostało doręczone do druku nr 2644. Jej przyjęcie spowoduje bezprzedmiotowość pozostałych propozycji. Do pytania zgłosiła się pani poseł Izabela Śledzińska-Katarasińska.

Panie i Panowie Posłowie! Mam pytanie do przewodniczącego Rady Mediów Narodowych, pana posła, pana redaktora Krzysztofa Czabańskiego. Wczoraj z rozbrajającą szczerością przyznał, że rada zajmuje się tylko i wyłącznie obsadzaniem zarządów, rad nadzorczych i rad programowych spółek. Niczym innym. A na co i jak te zarządy tam rządzą, to już rady nie interesuje. A więc mam takie pytanie. Ponieważ według mnie już te wszystkie konfitury zostały rozdane, te wszystkie posady zostały przydzielone, to w takim razie kiedy pan przewodniczący poseł, redaktor poda to biuro kadr ministerstwa propagandy dobrej zmiany do dymisji? Pora powiedzieć, panie prezesie: zadanie wykonane. Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. W 2. poprawce wnioskodawcy proponują nadać nowe brzmienie projektowi uchwały. Jej przyjęcie spowoduje bezprzedmiotowość pozostałych propozycji. Przystępujemy do głosowania. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Do pytania zgłosił się poseł Robert Winnicki, poseł niezrzeszony. Wysoka Izbo! Jak funkcjonuje Rada Mediów Narodowych w praktyce? W praktyce wygląda to tak. Pan poseł Czabański promuje ustawę w Sejmie, ustawę o zniszczeniu, o likwidacji jednej z branż rolniczych.

Co robi pan poseł Czabański? Pan poseł Czabański jako organ nadzorujący funkcjonowanie mediów publicznych na Twitterze zapowiada, że w sprawie tego programu, który poszedł nie po jego myśli, będzie interweniował u prezesa telewizji. Proszę państwa, to jest rażący konflikt interesów. Zrobiliście z telewizji publicznej tanią, tępą propagandówę i nawet tego nie ukrywacie, i macie olbrzymi konflikt interesów z tym, co robicie. To jest wbrew jakimkolwiek zasadom etycznym. Kto jest przeciw?

Wysoka Izbo! Kiedy partia rządząca tworzyła Radę Mediów Narodowych, zwróciłem uwagę z tego samego miejsca na absurd, jaki przy okazji tego się pojawił, czyli na to, że tworzyliśmy Radę Mediów Narodowych, jednocześnie nie posiadając w ogóle mediów narodowych. Ten absurd tak naprawdę trwa nadal i ten absurd drenuje kieszeń naszego podatnika do cna tylko po to, żeby tak naprawdę dublować zadania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Kiedy wiceprzewodniczący stowarzyszenia skutecznie zgłosił się do Rady Mediów Narodowych ze skargą na działalność i bojkotowanie stowarzyszenia w Warszawie przez warszawski ośrodek Telewizji Polskiej i Radio dla Ciebie, ta Rada Mediów Narodowych przesłała tę skargę gdzie? Do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Wydajemy pieniądze tylko po to, żeby kilku posłów rządzącej koalicji mogło tytułować się ministrami. Wzywam do natychmiastowej likwidacji Rady Mediów Narodowych [[Dzwonek]] i przywrócenia status quo. Pytanie zadaje pan poseł Krzysztof Mieszkowski, klub Nowoczesna. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Nigdy nie zgadzam się z panem Robertem Winnickim, ale dzisiaj po raz pierwszy - tak. Otóż Rada Mediów Narodowych jest oczywiście organem niepotrzebnym, absurdalnym, groteskowym w naszej rzeczywistości demokratycznej. Ale ona ma jedno bardzo poważne zadanie. Obsadzanie stanowisk to jest bardzo ważna polityczna decyzja. Przed nami wybory samorządowe. Rada Mediów Narodowych będzie służyła kreowaniu rzeczywistości medialnej przed tymi wyborami. Niedawno zostały powołane osoby, które od kilku dni czy od kilku tygodni pełnią funkcje szefów rad programowych. Chyba nie ma, panie Czabański - i proszę mi na to odpowiedzieć - ani jednej osoby niezwiązanej ze środowiskiem PiS w tym gronie. Czy to jest prawda, czy nie?

Wysoka Izbo!

tych, którzy nie idą po linii partyjnej PiS-u.

I coraz więcej właśnie środowisk niezależnych, konserwatywnych, prawicowych, narodowych i katolickich to widzi - widzi, jak bardzo ciasna, wąska i nieprzyszłościowa jest wasza wizja. Pytanie zadaje poseł Michał Kamiński, klub Polskiego Stronnictwa Ludowego. Mam pytanie do pana przewodniczącego Rady Mediów Narodowych jako wybitnego - i mówię to bez ironii - dziennikarza. Czy pana zdaniem, panie przewodniczący, w dzisiejszym wydaniu „Wiadomości” telewizyjnych Polacy powinni się dowiedzieć, jak najbliższy doradca premiera Netanjahu ocenia politykę zagraniczną polskiego rządu w kontaktach z Izraelem? Czy „Wiadomości” telewizyjne powinny dzisiaj podać, że zdaniem tego, kto negocjował z rządem pana Morawieckiego, rząd pana Morawieckiego skulił ogon przed premierem Netanjahu?

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu uchwały w brzmieniu z druku nr 2644, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał?

Sejm podjął uchwałę w sprawie informacji o działalności Rady Mediów Narodowych w 2017 roku. Powracamy do rozpatrzenia punktu 21. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 2664-A. Proszę pana posła Bogdana Rzońcę o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji. Panie Marszałku! Przedstawiam sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania.

Komisje wnoszą o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 2664. Komisje w dodatkowym sprawozdaniu przedstawiają również poprawki, nad którymi Sejm głosować będzie w pierwszej kolejności.

Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie. Komisje wnoszą o ich przyjęcie. Do pytania zgłosił się pan poseł Krzysztof Truskolaski, klub Nowoczesna. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W tej ustawie chcecie dać ludziom mieszkania na 9 lat czy nawet na 15, tak jak proponuje jedna z tych poprawek. A co po tych 15 latach? Gdzie ci ludzie po tych 15 latach się wyprowadzą? Ta ustawa dezaktywizuje społeczeństwo. Ta ustawa nie zachęca do tego, aby człowiek mieszkający w tym mieszkaniu zarabiał więcej. Bo co, jeżeli najemca dostanie propozycję lepiej płatnej pracy lub jeżeli najemca dostanie propozycję podwyżki?

Pytanie zadaje pan poseł Cezary Grabarczyk, klub Platformy. Panie Marszałku! Mieszkanie to rzecz ważna, dla rodziny najważniejsza, ale trzeba szukać różnych sposobów, aby zaspokajać potrzeby mieszkaniowe Polaków. Państwo likwidujecie program „Mieszkanie dla młodych”, program, który pozwolił pozyskać mieszkanie ok. 300 tys. polskich rodzin. Jednocześnie kuglujecie państwo w propozycjach ustawowych.

Skąd?

Kto jest przeciw?

Sejm poprawki przyjął. Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie. Do pytania zgłosiła się pani poseł Krystyna Sibińska, klub Platformy Obywatelskiej. Wysoka Izbo! Niby PiS coś chce dać, ale z drugiej strony straszy karami. Nie wystarczą wam oświadczenia, będziecie żądać zaświadczeń, jeśli któryś urzędnik będzie miał wątpliwości. A jak zaświadczeń będzie mało, to uruchomicie wszystkie służby, żeby sprawdzić tego najemcę, ale nie tylko najemcę, całą jego rodzinę. Więcej zaufania do obywateli. Proszę o poparcie tej poprawki.

Ja państwu postaram się szybko wytłumaczyć, jak działa PiS. Podatek od nieruchomości komercyjnych, druga stawka podatku od najmu mieszkań, podatek bankowy obciążający kredyty hipoteczne - to są trzy podatki, które wprowadziliście, które obciążają budownictwo mieszkaniowe w Polsce i najem w takich budynkach. Pensja dla was, premia dla was i jeszcze pieniądze dla znajomych prezesa. A potem macie 50 zł i mówicie obywatelom, że coś im dajecie na czynsz. Właśnie na tym polega wasze rządzenie. Nie dajmy się okłamywać, to nie są żadne pieniądze, które dajecie. Pytanie: Według jakiego klucza będą dzielone?

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawki odrzucił.

Do pytania zgłosił się pan poseł Mirosław Suchoń, klub Nowoczesna. Panie Marszałku! Kiedy niemalże 2 lata temu Prawo i Sprawiedliwość wprowadzało płacę minimalną, wprowadzało godzinową stawkę minimalną, z tej trybuny szła taka propaganda, że teraz oto Polacy będą godnie zarabiać i będzie ich stać na wszystko.

Dzisiaj zabieracie im te pieniądze, wyciągacie Polakom pieniądze z kieszeni i udajecie, że coś im dajecie. Tymczasem wyciągacie pieniądze z kieszeni, potrącacie swoje na premie i tę resztę, która zostaje, w postaci takich socjalistycznych programów próbujecie.

Wysoka Izbo! Nie mogę słuchać tego, co tutaj pan poseł przed chwilą mówił. Proszę państwa, inteligentnych ludzi rozpoznajemy po tym, jak zarabiają pieniądze, a mądrych po tym, jak wydają.

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę odrzucił. Komisje wnoszą o odrzucenie tej poprawki.

Wysoka Izbo! W 2016 r. rząd przyjął uchwałę, w której przyjął narodowy program mieszkaniowy. Od tego czasu upłynęły już prawie 2 lata i mamy wielką klapę. Media donoszą, że firmy budujące tanie mieszkania na wynajem upadają. Media donoszą, że najemcy są zaskoczeni wysokością niskich czynszów, które są w istocie czynszami komercyjnymi.

Panie ministrze, skąd ten upór? Pytanie zadaje pani poseł Paulina Hennig-Kloska, klub Nowoczesna. Panie i Panowie Posłowie! Pan poseł miał rację, byliśmy w rachunkach niedokładni, zapomnieliśmy przecież o obietnicy, którą złożyliście wyborcom, obniżenia VAT-u do starych stawek, czyli do podatku od najmu nieruchomości komercyjnych, który obciąża mieszkania, drugiej stawki podatku od dochodów z najmu, podatku bankowego, który wprost doliczany jest do kredytów hipotecznych.

To są konkretne pieniądze obywateli, które im zabieracie każdego dnia. Nie macie prawa nigdy więcej mówić, że cokolwiek im dajecie. Polska nie jest krajem płynącym ropą. Tu pieniądze do budżetu dają obywatele. Przystępujemy do głosowania. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Przed przystąpieniem do głosowania nad całością projektu ustawy do pytania zgłosiła się pani poseł Małgorzata Chmiel, klub Platformy Obywatelskiej. Szanowni Państwo! Projekt dopłat jest dowodem na to, że przyznajecie się do porażki programu M+ w systemie KZN-u. Chciałam się zapytać, co będzie z najemcami tych mieszkań, kiedy skończy im się okres dopłat.

Wysoka Izbo! Alexis de Tocqueville powiedział, że demokracja kończy się wtedy, gdy parlament zauważy, że można obywateli przekupić ich własnymi pieniędzmi. Państwo nie tylko to zauważyli, państwo uczynili sobie z tej zasady modus operandi. Dlaczego nie dać obywatelowi wędki? Państwo najpierw zabierają obywatelowi rybę poprzez podnoszenie kolejnych podatków, a później łaskawie dają pół tej ryby. A my mówimy prosto: Jeżeli chcemy, by młodzi ludzie się bogacili, by Polacy mogli godnie zarabiać i żeby ich było stać na własne mieszkanie, to musimy dać im wędkę, czyli obniżyć koszty pracy, czyli przede wszystkim obniżyć opodatkowanie pracy i przestać im zabierać 40% pensji. Proponujemy obniżenie kosztów pracy, opodatkowania pracy, dlatego w całości będziemy głosować za odrzuceniem tego [[Dzwonek]] kłamliwego projektu. Panie Marszałku! Wspieranie budowy mieszkań pod wynajem jest kwestią niezwykle ważną. Państwo powinno stworzyć kompleksowy program mieszkaniowy. Nowoczesna popiera program budowy mieszkań pod wynajem, ale nie w tej postaci. To rozwiązanie nie wspiera ciężkiej pracy Polaków i nie zachęca ich do zarabiania, tylko zachęca ich do kombinowania i dezaktywizuje nasze społeczeństwo. Rozwiązanie tego problemu może być proste. Jeżeli przestaniecie na Polaków nakładać setki podatków, które generują tylko i wyłącznie wzrost kosztów naszego życia, to na pewno Polacy będą mieli pieniądze na własne M. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto się wstrzymał?

Sejm uchwalił ustawę o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania. Powracamy do rozpatrzenia punktu 22. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 2700. Do pytania zgłosiła się pani poseł Genowefa Tokarska, klub PSL.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ta ustawa, Wysoka Izbo, pozwala na blokadę przedsiębiorcom, klientowi każdego rachunku w banku lub w SKOK-u na okres do 72 godzin bez możliwości zaskarżenia i bez wiedzy, bez informacji o tej blokadzie. W związku z tym pytam, czy Krajowa Administracja Skarbowa poniesie odpowiedzialność za pomyłki w blokadach środków przedsiębiorców. Bank, który ma być niemy i nie może informować, czy Krajową Administrację Skarbową? Jeszcze drugie pytanie: Czy rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, sympatyczny były poseł ziemi lubelskiej, będzie mógł poinformować swoich podopiecznych, jakie prawo przedsiębiorcom [[Dzwonek]] zgotował PiS?

Co jest? Udało się. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! To bardzo ważny z punktu widzenia bezpieczeństwa polskich przedsiębiorców projekt. Tak jak już przed chwilą tutaj usłyszeliśmy, administracja podatkowa bez powiadomienia, bez możliwości odwołania będzie mogła zablokować konto przedsiębiorcy na 72 godziny. Jeszcze raz powtórzę: bez postanowienia i bez prawa zaskarżenia tej decyzji. To jest naruszenie podstawowych zasad konstytucyjnych. To jest naruszenie art. 78 konstytucji, czyli prawa do zaskarżenia, zaufania obywatela do państwa, art. 2, i wreszcie zasady proporcjonalności. I to nie jest tylko moja opinia.

Panie Marszałku!

Już w tym roku wzrost upadłości wynosi 21%, a przewiduje się, że docelowo upadnie 30% więcej firm w stosunku do roku ubiegłego, a już w roku ubiegłym był niezły wzrost. Co to powoduje? Oczywiście przede wszystkim problemy z płynnością, split payment, wstrzymywanie im VAT-u, ale też z rentownością, bo rosną koszty pracy, są nowe opłaty i podatki. Oczywiście są problemy na rynku pracy. Problem ze znalezieniem pracownika kończy się niewykonaniem kontraktu.

W czasie pierwszego czytania mówiłem o tym, że jesteśmy na wojnie, na wojnie podatkowej, natomiast ta propozycja, czyli blokowanie kont przedsiębiorców, te 72 godziny bez postanowienia, bez możliwości zaskarżenia, to jest po prostu przegięcie. Nie powiem co. Każdy przedsiębiorca od momentu, kiedy pan prezydent podpisze tę ustawę, może żyć w ciągłej niepewności, czy będzie mógł dokonać płatności, a co za tym idzie, czy upadnie, czy nie. Jeżeli dojdzie do sytuacji, w której przedsiębiorcy upadną, ludzie trafią na bruk, ich kontrahenci nie dostaną pieniędzy. To może powodować bardzo niebezpieczny proceder. Byliśmy za tym, żeby procedować nad tą ustawą w komisji, żebyście się państwo opamiętali, żebyście nie kręcili bata na przedsiębiorców.

Powracamy do rozpatrzenia punktu 23. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 2687-A. Proszę panią poseł Annę Czech o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji. Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić dodatkowe sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw, druki nr 2333, 2687 i 2687-A. W drugim czytaniu zgłoszono osiem poprawek.

Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 2687. Komisja w dodatkowym sprawozdaniu przedstawia również poprawki, nad którymi Sejm głosować będzie w pierwszej kolejności.

Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Z pytaniem zgłosiła się pani poseł Anna Nemś, klub Platformy. Wysoka Izbo! Partnerstwo publiczno-prywatne jest bardzo ważnym źródłem pozyskiwania funduszy na inwestycje publiczne. Jest to ważne źródło w całej Europie, tylko niestety nie w Polsce. W Polsce, podobnie jak strefy ekonomiczne, PPP jest w całkowitym odwrocie. Dzisiaj ta ustawa, którą państwo przedstawiacie, tej sytuacji nie zmieni. Próbujemy ją poprawić. W 1. poprawce dajemy możliwość, aby podmiot publiczny mógł wystąpić z wnioskiem o opinię na temat zasadności realizacji przedsięwzięcia PPP nie tylko do ministra do spraw rozwoju regionalnego, ale również do właściwego marszałka. Marszałkowie w tym zakresie mają duży potencjał dotyczący opiniowania formy realizacji tego przedsięwzięcia. Będzie to też oznaczało większą samodzielność jednostek samorządu terytorialnego i nieangażowanie władz centralnych, aby miały czas na inne ważne czynności. Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Przystępujemy do głosowania. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Przystępujemy do głosowania.

Sejm poprawkę odrzucił. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Wysoka Izbo! W tej poprawce proponujemy zapewnienie ochrony płatności podwykonawców przez partnera prywatnego.

Proszę państwa, ja mam pytanie w tej sytuacji: A gdzie jest rzecznik MŚP, rzecznik, który ma bronić praw przedsiębiorców? 2 tygodnie temu dostał nominację polityczną - prosto z ławy poselskiej na urząd. Pewnie teraz jest zainteresowany gromadzeniem gadżetów, a tu, proszę państwa, co ustawa, to problemy dla przedsiębiorców, tak samo jak w przypadku przed chwilą głosowanej ordynacji podatkowej.

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił.

Przystępujemy do głosowania. Kto się wstrzymał?

Komisja wnosi o ich przyjęcie. Do pytania zgłosiła się pani poseł Anna Nemś, klub Platformy. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W poprawce tej chcielibyśmy, aby minister do spraw rozwoju regionalnego przedkładał sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie PPP nie tylko Radzie Ministrów, ale również właściwej komisji sejmowej. Taką sytuację mamy w strefach właśnie, takie sprawozdania są.

Mam nadzieję, że państwo poprzecie tę poprawkę i zagłosujecie za. Kto się wstrzymał?

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę odrzucił. Przed przystąpieniem do głosowania nad całością projektu ustawy do pytania zgłosiła się pani poseł Anna Nemś, klub Platformy. Wysoka Izbo! W partnerstwie publiczno-prywatnym dzięki podziałowi zadań, odpowiedzialności i ryzyka osiąga się najbardziej efektywne ekonomicznie sposoby dostarczania usług publicznych. Każda ze stron, zarówno strona publiczna, jak i strona prywatna, czerpie korzyści.

Szanowni państwo, w roku 2017 wszczęto ile? 16 postępowań. W latach poprzednich było to 50, 60. Podmiot prywatny nigdy nie zaryzykuje swoich pieniędzy w sytuacji niepewności i braku stabilizacji. Czy ta procedowana ustawa coś zmieni? Nie zmieni. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 2687, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał?

Powracamy do rozpatrzenia punktu 24. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych, Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Trzeciego Protokołu do Porozumienia ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy, sporządzonego w Strasburgu dnia 6 marca 1959 r. Komisje wnoszą o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 2546. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 2546, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Wszyscy byli za.

Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. W dyskusji zgłoszono wniosek o skierowanie projektu ustawy dodatkowo do Komisji Finansów Publicznych, Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Propozycją zaopiniowaną przez Prezydium Sejmu jest, aby Sejm skierował ten projekt ustawy do Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w celu rozpatrzenia. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję zaopiniowaną przez Prezydium Sejmu przyjął, a wniosek o dodatkowe skierowanie tego projektu ustawy poddam pod głosowanie. Sprzeciwu. Sprzeciw przeciwko czemu? No przecież właśnie będziemy nad tym głosować. A, jest pytanie, w międzyczasie jeszcze wpłynęło. Pani poseł Krystyna Sibińska, klub Platformy. Wysoka Izbo! Zmiana będzie skutkowała również utrwaleniem wizerunku Wód Polskich jako rzetelnego kontrahenta w dłuższej perspektywie czasu. To jest cytat z uzasadnienia tego projektu uchwały. Sami w to nie wierzycie, bo wczoraj, kiedy ta ustawa była procedowana, na sali nie było nikogo z PiS-u. Nie było pani premier Szydło, która z tej mównicy tak bardzo broniła tej ustawy. Nie było pani poseł Paluch, która tak sprytnie przeprowadziła tę ustawę przez Sejm.

Tak się wstydzicie tej ustawy, że chcecie to wrzucić do jednej komisji. Chcecie, zgodnie z receptą waszego premiera, dżumę leczyć cholerą, ale wam to nie wyjdzie. Nie naprawicie tej ustawy, nie poprawicie wizerunku, a my to wyjaśnimy w komisji śledczej. Pani poseł, jeszcze chwileczkę.

Rozumiem. Wysoka Izbo! Ja trochę posłów PiS rozumiem. Oni po prostu chcieli wykluczyć z prac nad tą ustawą jedną swoją posłankę i dlatego chcieli zawęzić prace tylko do jednej komisji, ale sprawa jest naprawdę bardzo poważna. Państwo musicie wiedzieć, że to tak naprawdę dotyczy funkcjonowania Wód Polskich i musi się tym zająć komisja finansów. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości.

Nie otrzymali tych pieniędzy.

Wysoka Izbo! Pani poseł powiedziała, że Wody Polskie są uczciwym kontrahentem, więc pomyślałem, że muszę wyjść i zapytać.

Czy otrzymali już te podwyżki czy nie? Drodzy państwo, tutaj chodzi również o to, że skoro ministerstwo zawiera porozumienie z pracownikami, na podstawie którego mają oni dostać podwyżki, to jeżeli oni tych pieniędzy nie dostali, to narażacie państwo na straty również w postaci konieczności zapłacenia im odsetek ustawowych. Jeżeli przychodzi minister i zawiera porozumienie, na podstawie którego pracownicy mają otrzymać podwyżkę wynagrodzenia, to to się nie liczy? Robi się z gęby cholewę?

Kto się wstrzymał?

Kto się wstrzymał?

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 33. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2683 i 2690) Proszę panią poseł Annę Paluch o przedstawienie sprawozdania komisji. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Komisja proponuje wszystkie te poprawki przyjąć. Jeżeli Sejm nie odrzuci poprawki Senatu, uważa się ją za przyjętą. W punktach porządku dziennego dotyczących rozpatrywania poprawek Senatu głosować będziemy nad wnioskami o odrzucenie poprawek Senatu.

Przystępujemy go głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 1. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę przyjął. Przystępujemy go głosowania. Kto jest przeciw?

Sejm poprawkę przyjął. Przystępujemy do głosowania. Kto się wstrzymał?

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 34. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2681 i 2704) Proszę pana posła Bogdana Rzońcę o przedstawienie sprawozdania komisji. Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Głosować będziemy zgodnie z zasadami stosowanymi w poprzednim punkcie porządku dziennego. Przystępujemy do głosowania. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Wszyscy byli przeciw.

Proszę pana posła Bogdana Rzońcę o przedstawienie sprawozdania komisji. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Senat przyjął w tym przypadku dwie poprawki i proponujemy przyjęcie tych poprawek, czyli też głosowanie na czerwono. Głosować będziemy zgodnie z zasadami stosowanymi w poprzednim punkcie porządku dziennego. Z poprawką tą łączy się poprawka 2. Komisja wnosi o ich przyjęcie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawki przyjął. Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie uchwały Senatu w sprawie ustawy o tachografach. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 36. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o własności lokali (druki nr 2684 i 2695) Proszę pana posła Ryszarda Bartosika o przedstawienie sprawozdania komisji. Panie Marszałku! Państwo Ministrowie! Wysoka Izbo! Senat przyjął dwie poprawki. Komisje wnoszą o przyjęcie tych poprawek. Głosować będziemy zgodnie z zasadami. Senat proponuje skreślić wyrazy „chyba, że w budynku po tej dacie przeprowadzono roboty budowlane wymagające pozwolenia na budowę” Do pytania zgłosiła się pani poseł Małgorzata Chmiel, Platforma Obywatelska.

Szanowni Państwo! Cieszymy się, że przyjęliście te poprawki, które myśmy sugerowali, ponieważ to już trzeci raz jest poprawiany ten sam przepis. Czy nie lepiej było od razu posłuchać tego, co my mówimy? Czy wy państwo myślicie, że chcemy wam dokuczyć? My chcemy po prostu stanowić dobre prawo i naprawiać. A więc następnym razem bardzo proszę posłuchać tego, co my mówimy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę przyjął. Komisje wnoszą o przyjęcie tej poprawki. Przystępujemy do głosowania. Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę przyjął. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 37. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2682 i 2694) Proszę pana posła Janusza Śniadka o przedstawienie sprawozdania komisji. Pana posła Janusza Śniadka proszę o przedstawienie. Wysoka Izbo! Senat po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych, druk nr 1933, wprowadził do niej 10 poprawek natury legislacyjno-redakcyjnej. Komisja Polityki Społecznej i Rodziny po rozpatrzeniu poprawek Senatu wnosi do Wysokiej Izby, niespotykanie jednomyślnie, o przyjęcie wszystkich poprawek Senatu.

Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę przyjął. Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.

Nikt nie był za, przeciw - 310, wstrzymało się 100. Sejm poprawkę przyjął. Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki. Przystępujemy do głosowania. Kto się wstrzymał?

Przystępujemy do głosowania. Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę przyjął.

Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nikt nie był za, przeciw - 409, 1 się wstrzymał. Sejm poprawkę przyjął. Przystępujemy do głosowania.

Sejm poprawkę przyjął. Przystępujemy do głosowania. Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę przyjął. Senat proponuje inne brzmienie ust. 1.

Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę przyjął. Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki. Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę przyjął. Przystępujemy do głosowania. Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę przyjął. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 38. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (druki nr 2685 i 2691) Proszę pana posła Wojciecha Murdzka o przedstawienie sprawozdania komisji. Wysoka Izbo! Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, druk nr 2685. Po rozpatrzeniu wszystkich poprawek zgłoszonych przez Senat - tych poprawek było 31 - komisja wnosi o przyjęcie wszystkich poprawek. Dziękuję bardzo. Głosować będziemy zgodnie z zasadami przyjętymi poprzednio. Senat zgłosił do ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie. Przystępujemy do głosowania.

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Wszyscy byli przeciw. Sejm poprawki przyjął.

Komisja wnosi o jej przyjęcie. Okej. Kto się wstrzymał?

Komisja wnosi o jej przyjęcie. Przystępujemy do głosowania.

Przeciw - 410, 1 się wstrzymał. Sejm poprawkę przyjął. Komisja wnosi o ich przyjęcie. Kto się wstrzymał? Sejm poprawki przyjął.

Komisja wnosi o jej przyjęcie. Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę przyjął. Senat proponuje odpowiednio dodać wyrazy „spółek cywilnych osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku” Kto się wstrzymał? Głosowało 411 posłów. Wszyscy byli przeciw. Sejm poprawkę przyjął.

Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę przyjął.

Przystępujemy do głosowania. Kto się wstrzymał? Sejm poprawki przyjął. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 39. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2686 i 2715) Proszę pana posła Krzysztofa Kubowa o przedstawienie sprawozdania komisji. Wysoka Izbo! Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii na posiedzeniu w dniu 5 lipca rozpatrzyła poprawki Senatu. Głosować będziemy zgodnie z zasadami stosowanymi poprzednio.

Kto się wstrzymał?

Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie. Kto się wstrzymał?

Kto się wstrzymał? Za - 2, przeciw - 406, wstrzymał się - 1. Sejm poprawkę przyjął. Powracamy do rozpatrzenia punktu 29. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Podczas drugiego czytania projektu ustawy, w związku ze zgłoszeniem do niego poprawek, wobec propozycji ponownego skierowania tego projektu do Komisji Nadzwyczajnej w celu przedstawienia sprawozdania zgłoszono sprzeciw. Pod głosowanie poddam propozycję skierowania projektu ustawy do Komisji Nadzwyczajnej w celu przedstawienia dodatkowego sprawozdania. Odrzucenie tej propozycji oznaczać będzie, że Sejm przystąpi do trzeciego czytania po doręczeniu paniom i panom posłom zestawienia zgłoszonych poprawek. Do pytań zgłosiła się pani poseł Krystyna Sibińska, klub Platformy. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Od dzisiaj planowaniem przestrzennym i realizacją inwestycji powinni zajmować się teolodzy, politycy, historycy, bo takie osoby, nie umniejszając ich kompetencjom w innych dziedzinach, są w komisji deregulacyjnej. Dlatego zgłosiliśmy sprzeciw, ponieważ od zawsze inwestycjami mieszkaniowymi, wszystkimi propozycjami dotyczącymi budownictwa mieszkaniowego zajmowała się Komisja Infrastruktury, a jeśli chodzi o planowanie przestrzenne, stanowienie prawa miejscowego, projekty zawsze trafiały do komisji samorządu. Dzisiaj to wyszło taką dziwną drogą. Komisja deregulacyjna zajmuje się stanowieniem prawa mówiącego o tym, że nowe inwestycje będą budowane w oparciu o uchwały rad gmin. Nijak się to ma do deregulacji, naprawdę.

Wysoka Izbo! Szanowni państwo, mówimy o ustawie, która w niektórych kręgach już jest nazywana ustawą deweloper+. I to powinno dać państwu do myślenia, już tylko to. z zaskoczenia została skierowana do komisji, i to nie komisji merytorycznej, Komisji Infrastruktury, która mogłaby merytorycznie powiedzieć, co w tej ustawie jest, tylko trafiła do komisji do spraw deregulacji, chociaż ta ustawa z tą komisją, z deregulacją nie ma absolutnie nic wspólnego, chyba że za deregulację uważać coś, co wprowadza ta ustawa, czyli możliwość obejścia planów zagospodarowania przestrzennego, to rzeczywiście jest to deregulacja.

Panie Premierze! Jesteśmy przeciwni jako klub ponownemu skierowaniu tego ważnego projektu do komisji deregulacyjnej. Prawidłowymi odbiorcami tego projektu powinny być dwie komisje: Komisja Infrastruktury i komisja samorządu. Panie marszałku, jeszcze jedna ważna kwestia - została złamana procedura. Otóż pan marszałek zobowiązał nasze dwie komisje do wyrażenia opinii dla komisji do spraw deregulacji.

Kto z pań i panów posłów jest za ponownym skierowaniem tego projektu do Komisji Nadzwyczajnej, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

W pierwszej kolejności pod głosowanie poddam wniosek o odrzucenie projektu ustawy w całości. Jego przyjęcie spowoduje bezprzedmiotowość pozostałych propozycji.

Szanowni Państwo! Platforma Obywatelska zgłosiła wniosek o odrzucenie projektu w całości, dlatego że ustawa przygotowana przez PiS, specustawa mieszkaniowa, która miała służyć obywatelom, to ustawa deweloperska. To nie jest ustawa obywatelska, ale właśnie deweloperska. Ustawa w żaden sposób nie gwarantuje budowania mieszkań czynszowych, społecznych czy komunalnych, pozwala za to na budowanie apartamentów i ekskluzywnych osiedli. Ustawa zezwala na dewastowanie przestrzeni, wprowadza przepisy obciążające gminy działaniami deweloperów, stawia interes prywatny ponad publicznym, stwarza przestrzeń do działań nieprzejrzystych i zachowań korupcjogennych, ma negatywną opinię Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, jest także sprzeczna z ideą, o której mówił sam PiS. Projekt miał być skierowany do osób o niskich i średnich dochodach, a jest skierowany do deweloperów. Wysoka Izbo! Nowoczesna również złożyła wniosek o odrzucenie tej ustawy. Ta ustawa powinna być odrzucona, a CBA powinno się zająć sprawdzeniem procesu legislacyjnego. Trzeba sprawdzić, kto tak naprawdę wpływał na ministerstwo, żeby robić przy okazji tej ustawy różnego rodzaju przekręty. Pozwalacie na mocy tej ustawy unieważnić de facto plany zagospodarowania przestrzennego i zrealizować sobie inwestycję, jaką chcecie. To jest po prostu skandaliczny przepis, za którym zapewne ktoś musi stać. Bo nie boicie się i w art. 5 wprost wypisujecie, kto prawdopodobnie za tym stoi: właściciele gruntów PKP i gruntów wojskowych, a więc tych, które teraz są wprost zależne od ministra Błaszczaka i od ministra Adamczyka. Panie Ministrze! W Ministerstwie Infrastruktury nieraz dochodziło do działań korupcjogennych, już za pana czasów. Głos zabierze przedstawiciel Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju sekretarz stanu Artur Soboń. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Otóż ta ustawa nie likwiduje planów zagospodarowania przestrzennego. Plany zagospodarowania przestrzennego obowiązują. Tyle mamy terenów objętych planami zagospodarowania przestrzennego w miastach, bardzo często szczególnie w dużych miastach, gdzie ten proces tworzenia planu zagospodarowania przestrzennego trwa długo, latami, i gdzie co trzeci plan zagospodarowania przestrzennego nie obejmuje nawet 1 ha terenu i nie jest żadnym planowaniem przestrzennym, tylko załatwianiem pojedynczych interesów. Może łatwiej jest bez planów zagospodarowania przestrzennego łowić w mętnej wodzie, bo prezydenci, burmistrzowie wydali.

W Warszawie pani prezydent Warszawy z Platformy Obywatelskiej wydała ich 1473, w Lubinie - 707, prezydent Poznania wydał 852, prezydent Łodzi - 1969, prezydent. Krakowa - 1936, prezydent Gdańska - 309, prezydent Bydgoszczy - 303. Ja tak mogę wymieniać w nieskończoność. To jest. To oni wprowadzają chaos urbanistyczny, z którym my kończymy, bo my po raz pierwszy w tej ustawie wprowadzamy standardy urbanistyczne i wprowadzamy konieczność realnego. planowania przestrzennego, tak aby można było zagospodarować pod budownictwo mieszkaniowe tereny, które są dostępne, tereny pokolejowe, powojskowe, tereny rolne, tereny poprzemysłowe, tereny popocztowe, po to żeby budować szybciej, żeby budować taniej, żeby budować więcej. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie projektu ustawy w całości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Do zadania pytania zgłosiła się pani poseł Krystyna Sibińska, klub Platformy. Wysoka Izbo! Jeśli to mają być tanie mieszkania, to zmieńcie definicję inwestora i dopiszcie, że inwestor to jest taka osoba, która będzie budowała w formie budownictwa czynszowego, komunalnego bądź społecznego. Jeśli tego nie zmienicie, to potwierdzicie tylko tezę, że umówiliście się z deweloperami po to, żeby ułatwić im budowanie na ich terenach. I tylko po to będziecie to robić, żeby wypełnić tabelki ze slajdów premiera Morawieckiego.

Panie Premierze! Wysoka Izbo! Pan minister przed chwilą powiedział, że plany zagospodarowania przestrzennego zostają. Konstytucja jest, ale jej nie przestrzegacie. Robicie wszystko, żeby obejść ich zapisy. Plany zagospodarowania przestrzennego będą, ale deweloperzy będą hasać po tych planach, jak tylko będzie im się podobało.

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił.